Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju. Od kilku lat toczy się w Polsce dyskusja o potrzebie i kierunkach zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Zmiany dokonywane w ostatnich latach nie obejmują tylko kwestii organizacyjnych, najbardziej widocznych w dyskusji publicznej. Wprowadzane są również zmiany w przepisach proceduralnych wyznaczających sposób postępowania przed sądami mające na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowań. Mimo tego działalność sądów w dalszym ciągu częściej spotyka się z krytyką niż z aprobatą. Według szerokiego badania CBOS poświęconego temu zagadnieniu odsetek Polaków, którzy na podstawie własnych doświadczeń wyrażali dezaprobatę wobec działalności sądów, wynosił 50%. Połowa badanych negatywnie oceniała więc funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w tym co ósmy twierdził, że działa on zdecydowanie źle. Według ostatnich danych działalność wymiaru sprawiedliwości ocenia pozytywnie 29%, a negatywnie 41% respondentów. Największymi bolączkami wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest, po pierwsze, brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a przynajmniej brak zaufania w takim stopniu, w jakim byśmy tego oczekiwali. Na drugim miejscu można wymienić opieszałość wymiaru sprawiedliwości, czyli przedłużające się, skomplikowane postępowania, których obywatele bardzo często nie są w stanie zrozumieć i które prowadzą do pogłębiania poczucia niesprawiedliwości. Nie zawsze jest to spowodowane kwestiami, które rozpatrywane są przez sąd, ale właśnie sposobem działania wymiaru sprawiedliwości. Przewlekłość wynika po części z liczby spraw, ale po części także z przyjętego modelu i sposobu postępowania. Procedury prawne wciąż pozostają dla zwykłych obywateli niezrozumiałe, a długotrwałe oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy, na wyrok czy postanowienie nie sprzyja budowaniu poczucia sprawiedliwości. Jest to jeden z poważniejszych problemów rzutujących nie tylko na funkcjonowanie struktur wymiaru sprawiedliwości, ale również na ogólną ocenę sprawności funkcjonowania państwa. Zdaniem wielu prawników i przedstawicieli instytucji państwowych potrzebne nam jest pilne podjęcie działań mających na celu odciążenie sądów, skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie i odbiurokratyzowanie procesu wymierzania sprawiedliwości. W marcu tego roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda utworzył w Kancelarii Prezydenta specjalny zespół kierowany przez pana prof. Piotra Kruszyńskiego, a złożony z przedstawicieli m.in. ministra sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, przedstawicieli Kukiz’15, osób, które posiadają doświadczenie zarówno naukowe, jak i procesowe, doradców i ekspertów. Celem tego zespołu było zidentyfikowanie potrzeb wymiaru sprawiedliwości pod względem wykorzystania instytucji sędziów pokoju. Idea ponownego wprowadzenia sędziów pokoju do wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie jest całkowicie nowa, gdyż dyskusja dotycząca wykorzystania tej instytucji w odpowiedzi na współczesne problemy władzy sądowniczej toczy się już od kilku lat. Na ziemiach polskich sędziowie pokoju funkcjonowali już w XIX w., na początku XX w., a także w odrodzonej Rzeczypospolitej. Postulując wprowadzenie instytucji sędziego pokoju, przywołuje się doświadczenia krajów systemu common law, takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, ale także krajów, w których obowiązuje system kontynentalny, tj. Szwajcarii oraz Belgii. W każdym z tych krajów pozycja sędziów pokoju jest różna. Historycznie rzecz ujmując: sędziów pokoju wprowadzono w celu odformalizowania i przyspieszenia procesu orzeczniczego. Jedną z dróg ku temu jest zmniejszenie kognicji sądów, czyli przekazanie części spraw, które dziś prowadzą sądy powszechne, utworzonym na podstawie zaproponowanej przez pana prezydenta regulacji sądom pokoju; drugą jest wprowadzenie w przypadku sądów pokoju uproszczonych procedur, które z racji charakteru spraw, jakie będą rozstrzygane w sądach pokoju, spowoduje, że sprawy zostaną rozpatrzone wnikliwie, ale i szybko. Inicjatywa ustawodawcza prezydenta Rzeczypospolitej składa się z dwóch ustaw: ustawy o sądach pokoju i ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju. Co one zawierają? Przede wszystkim ustanowienie sądów pokoju jako sądów najniższego szczebla w ramach sądów powszechnych, które odciążą sądy rejonowe. Czynności podejmowane przez sądy pokoju będą mieściły się w granicach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Sądy pokoju będą rozstrzygały sprawy mniejszej wagi, wyłącznie karne i cywilne. Skąd będą brali się sędziowie pokoju? Będą to osoby zainteresowane tym, żeby zostać sędziami pokoju, i które spełnią odpowiednie, przewidziane ustawą warunki. W pierwszej kolejności Krajowa Rada Sądownictwa będzie rozpatrywała kandydatury pod względem spełnienia kryteriów ustawowych, a następnie wszystkie te osoby, które w przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa będą te warunki spełniały i będą mogły zostać sędziami pokoju, będą poddawane weryfikacji wyborczej. Będą przeprowadzane wybory, w których lokalna społeczność zdecyduje ostatecznie o tym, kto zostanie sędzią pokoju. Tym samym zostanie poszerzony udział czynnika społecznego w kreowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wybory będą powszechne i bezpośrednie, proces głosowania Osoby, które zostały wybrane, zostaną przedstawione przez Krajową Radę Sądownictwa prezydentowi Rzeczypospolitej, który będzie powoływał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju. Sędzia pokoju pełniący urząd w oparciu o mandat pochodzący z wyboru niewątpliwie ma szansę cieszyć się dużym autorytetem i wzbudzać zaufanie społeczności lokalnej. Co istotne, sędziom pokoju zostaną stworzone warunki niezbędne do zachowania przez nich niezawisłości, analogiczne do tych, jakie konstytucja i ustawy przyznają sędziom zawodowym. W tym miejscu należy podkreślić, że mimo nowatorskiego charakteru proponowanej regulacji zaprojektowano ją w sposób przystający do aktualnych wymogów ustrojowych określonych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Odstępstwa są jednak dopuszczalne, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, wyjątki muszą być uzasadnione konstytucyjnie legitymowanym celem i mieścić się w granicach realizacji tego celu. Instytucja powierzenia pełnienia czynności sędziowskich osobom niebędącym sędziami służyć powinna przede wszystkim lepszej realizacji podmiotowego prawa określonego w art. 45 konstytucji, czyli prawa do sądu. Po drugie, muszą być spełnione wszystkie istotne materialnie warunki, od których uzależniona jest bezstronność, niezawisłość i niezależność sądu. Inaczej mówiąc, niezależnie od nazwy stanowiska służbowego status osoby, której powierzono pełnienie czynności sędziowskich, musi odpowiadać wzorcowi niezawisłości wynikającemu z konstytucyjnych przepisów dotyczących statusu sędziego. Z tego powodu projekt maksymalnie zbliża status sędziego pokoju do statusu sędziego w zakresie przyznanych praw, ale również obowiązków. Kandydat na sędziego pokoju będzie zobligowany posiadać wykształcenie prawnicze i co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej, bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa, a więc działalnością legislacyjną. Sędzia pokoju będzie musiał mieć ukończone 29 lat najpóźniej w dniu wyborów i mieć nie więcej niż 70 lat w dniu objęcia stanowiska sędziego pokoju. Sędziowie pokoju będą pełnili swoją funkcję przez okres 6-letniej kadencji. Projekt przewiduje możliwość pełnienia urzędu przez sędziego pokoju wyłącznie przez jedną kadencję, jednakże jeżeli sędzia pokoju pełni urząd przez mniej niż 4 lata wskutek przyjęcia mandatu lub wyboru w wyborach uzupełniających w toku kadencji sędziów pokoju, będzie mógł zostać w takiej sytuacji wyjątkowo wybrany na drugą kadencję. Projektowana regulacja dąży do zagwarantowania sędziom pokoju immunitetu. Ponadto sędziowie pokoju, analogicznie jak sędziowie zawodowi, nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia, być członkiem partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów lub niezawisłości sędziów pokoju. Wynagrodzenie sędziów pokoju będzie określone na poziomie wynagrodzenia asesora sądowego, które - przypomnę - wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego. Nie tylko sędziowie pokoju, lecz również sądy pokoju będą funkcjonowały kadencyjnie. Kadencja wszystkich sądów pokoju będzie wspólna i trwać będzie 6 lat. Termin rozpoczęcia nowej kadencji sądów pokoju, przypadający nie później niż 2 miesiące po wyborach sędziów pokoju, określi minister sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, w drodze rozporządzenia. Sądy pokoju zostaną związane organizacyjnie z sądami rejonowymi poprzez, co do zasady, tożsamość siedziby i obszaru właściwości sądu pokoju i sądu rejonowego, dyrektora i prezesa sądu pokoju, którymi będą odpowiednio dyrektor i prezes sądu rejonowego. Sąd rejonowy będzie rozpatrywał środki odwoławcze od orzeczeń sądu pokoju, czyli zachowana i utrzymana oczywiście zostanie konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania. Projekt zawiera również ukształtowane analogicznie do pozostałych szczebli sądów powszechnych zasady finansowania sądów pokoju i zatrudniania asystentów sędziego oraz urzędników i pracowników sądowych. W sprawach cywilnych do właściwości sądów pokoju będą należały sprawy o zawezwanie do próby ugodowej, o alimenty oraz rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Do właściwości sądów pokoju w sprawach karnych z kolei przekazano występki określone w Kodeksie karnym. Tutaj mogę podać tytułem przykładu m.in. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego czy prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień, po zakazie, zakłócanie miru domowego, rozpijanie małoletniego, napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej, zakłócanie przebiegu zgromadzenia, posługiwanie się cudzym dokumentem, także występki, jeżeli wartość mienia będącego przedmiotem przestępstwa albo wyrządzonej przestępstwem szkody nie przekracza 10 tys. zł. Uwzględniając to kryterium, byłyby to takie występki jak kradzież czy kradzież z włamaniem, ale w przypadku mniejszej wagi, przywłaszczenie, oszustwo w przypadku mniejszej wagi, zniszczenie mienia ruchomego czy paserstwo umyślne. Z kolei w sprawach o wykroczenia orzekanie przez sądy pokoju będzie stanowiło regułę. Sprawy te właściwie w całości znajdą się w jurysdykcji sądów pokoju. Do kognicji sądów pokoju, tak jak państwo widzicie, przekazano więc drobne sprawy o niewielkim stopniu skomplikowania. Ich rozpatrywanie przez sędziów pokoju odciąży inne sądy powszechne i pozwoli im skoncentrować się na rozpoznawaniu spraw bardziej skomplikowanych. Osiągniemy więc efekt przyspieszenia rozpoznania spraw nie tylko w tych sprawach, które bezpośrednio w uproszczonej procedurze zostaną skierowane do rozstrzygnięcia do sądu pokoju, ale także w tych wszystkich innych sprawach, gdzie moce przerobowe będą mogły być skierowane na rozpoznanie i podjęcie tych spraw, które dzisiaj oczekują na rozpoznanie. W projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju zawarto regulacje zmierzające do wprowadzenia w poszczególnych ustawach zmian niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania sądów pokoju. Przyjęto, że ustawa o sądach pokoju wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Z kolei wejście w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju podzielono na odpowiednio długie etapy. Najszybciej wejdą w życie przepisy umożliwiające działalność pełnomocnika do spraw utworzenia sądów pokoju. Celem działania pełnomocnika będzie opracowanie planu podziału terytorium Rzeczypospolitej na okręgi wyborcze, przygotowanie planów utworzenia sądów pokoju oraz podjęcie czynności zmierzających do zapewnienia sądom pokoju odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych. Najbardziej odłożono w czasie wejście w życie zmian dotyczących postępowania przed sądami pokoju oraz przyznających szczególne uprawnienia byłym sędziom pokoju, tj. możliwość przystępowania do zawodowych egzaminów prawniczych bez konieczności odbycia aplikacji.

Mówimy tutaj przecież o osobach, które będą miały już duże doświadczenie i które wcześniej miały to trzyletnie doświadczenie, i mają spełniony wymóg wykształcenia prawniczego. Rozszerzenie udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości mieszczące się w konstytucyjnych ramach art. 175 i art. 182 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest dużym wyzwaniem ustrojowym, technicznym i finansowym, niemniej w ostatecznym rozrachunku i perspektywie okaże się korzystne dla społeczeństwa. Nie do przecenienia są walory edukacyjne takiego rozwiązania, poczucie wspólnej odpowiedzialności za wymierzoną sprawiedliwość oraz poczucie sprawiedliwości wymierzanej innym obywatelom przez obywateli - niezawodowych sędziów. Celem powołania sądów pokoju jest wzmocnienie sądownictwa, tak by obywatele utożsamiali się z instytucjami wymiaru sprawiedliwości i mieli do sędziów zaufanie. Zwracam się do Wysokiego Sejmu w imieniu pana prezydenta o podjęcie prac nad wniesionymi projektami ustaw oraz rzetelną, merytoryczną dyskusję, której efektem będzie prawo stanowiące odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości, tak aby stał się on bliższy obywatelom, aby odzyskał akceptację społeczną i aby sądy w Polsce były uważane za sprawiedliwe. Przedstawienie Wysokiej Izbie projektów ustaw prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postrzega jako kolejny krok zmierzający do osiągnięcia tego celu. Biorąc pod uwagę te okoliczności, wnoszę o poparcie przez Wysoką Izbę przedstawionych (Dzwonek) projektów ustaw. Dziękuję bardzo uprzejmie, panie ministrze. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana posła Arkadiusza Myrchę o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy zawartego w druku nr 1378. Zapraszam, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej mam przyjemność i zaszczyt przedstawić uzasadnienie projektu objętego drukiem nr 1378, stanowiącego o wprowadzeniu do sądownictwa powszechnego nowej instytucji, tzw. obywatelskiego sędziego handlowego. Mówienie o tym, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, szczególnie w sądownictwie, nie jest dobra, jest truizmem. Wszyscy obserwujemy od kilku lat pogłębiającą się zapaść organizacyjną. Ale co gorsza, obserwujemy spadek zaufania ogólnie do wymiaru sprawiedliwości. Nie są to tezy, które wyjmujemy z kapelusza. Są to tezy potwierdzone twardymi danymi publikowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Są to tezy wynikające z cyklicznie przeprowadzanych badań, w szczególności przez CBOS.

Ale problemy są także, powiedzmy sobie, drobniejsze, organizacyjne, które podnoszone są w doktrynie, które podnoszone są przez praktyków.

Wiemy, że instytucja ławnika, która jest co do zasady dobra, wymaga korekt, wymaga zmian, o czym będę jeszcze w swoim wystąpieniu mówił.

Mówię tu właśnie o sprawach gospodarczych. Kiedy sięgniemy do statystyk, zauważymy, że jeszcze w 2011 r. średni okres oczekiwania na rozstrzygnięcie w sądach rejonowych w wydziałach gospodarczych wynosił 3,6 miesiąca. W 2020 r. jest to już 8 miesięcy. Wzrost jest gigantyczny, ale szkodę ponoszą przedsiębiorcy, strony postępowania. Podobnie jest w postępowaniach toczących się przed sądami okręgowymi. Dlaczego o tym mówię? To jest o tyle ważne, że nawet najlepszy wyrok, który został wydany przez najlepszego sędziego, nie będzie miał szans powodzenia, jeżeli strony postępowania, czyli obywatele, nie będą ufały temu sędziemu, nie będą ufały, że wyrok, który zapadł na sali posiedzeń, jest wyrokiem sprawiedliwym, że należy się z nim pogodzić i po prostu go zrealizować. Jeżeli będzie on kontestowany, jeżeli będzie kwestionowana wiedza sędziego, jego fachowość, to wtedy taki wymiar sprawiedliwości nie będzie spełniał swojej elementarnej zasady, czyli właśnie wymierzania tej sprawiedliwości. Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych nie jest też niczym nowym. Podobne instytucje funkcjonują w krajach europejskich. Projekt, który prezentujemy, jest częściowo zaczerpnięty z modelu austriackiego, który wprost posługuje się terminem sędziów handlowych. Cała tendencja w XXI w., jeżeli chodzi o reformowanie wymiaru sprawiedliwości, ukierunkowana jest na to, żeby ten tzw. czynnik społeczny, mówiąc wprost, żeby obywatele mieli trochę większy wpływ na to, co dzieje się na sali rozpraw, niż to miało miejsce dotychczas, żeby nie byli tylko stronami, uczestnikami postępowania, świadkami, ale także żeby byli tym głosem, czasami głosem rozsądku, czasami głosem doświadczenia, tak niezbędnego do orzekania w praktycznie wszelkich sprawach.

Ten projekt ustawy, co ważne, znajdujący się w pełni w ramach zarysowanych przez naszą ustawę zasadniczą, będzie poprawiał wszystkie te newralgiczne obszary.

Jest to instytucja nowa, dedykowana w szczególności właśnie postępowaniom gospodarczym, bo to jest odpowiedź na jeden z postulatów, który pojawia się w doktrynie, w orzecznictwie, a mianowicie postulat profesjonalizacji ławników. Często mamy do czynienia z sytuacją, że ławnicy orzekający na sali rozpraw nie mają takiej prawniczej czy fachowej wiedzy w sprawach, w których uczestniczą. Sędzia ma wiedzę prawniczą, zna procedury, zna materię, ale jemu też brakuje tej wiedzy. Postuluje się, żeby następowała taka profesjonalizacja ławników, żeby oni byli szkoleni w tych dziedzinach, w których orzekają: prawo karne, wykroczenia, sprawy rodzinne. Przyjmujemy ten model gospodarczy, bo tutaj może nie w łatwy sposób, ale w sposób taki namacalny jest możliwość wprowadzenia tej profesjonalizacji czynnika społecznego.

Bo jeżeli przedsiębiorcy, którzy kierują swój spór do sądu - a wiemy, że przedsiębiorcy do sądu idą chyba w ostateczności, podejmują próby ugodowe, czy to w formie arbitrażu, czy przed innymi instytucjami, albo w takim normalnym, zwyczajnym, codziennym życiu - jeżeli kierują tam swój spór o często duże, poważne sprawy, to potrzebują mieć zaufanie, potrzebują mieć zrozumienie w składzie orzekającym. I zobaczą, że obok fachowego sędziego, który zadbał o prawidłowość procedur, który będzie doskonale znał materię, zobowiązania, Kodeks spółek handlowych, będą jeszcze siedzieli przedsiębiorcy, którzy zapewnią ducha tego rozstrzygnięcia, którzy nakierują tego sędziego i jego doświadczenie życiowe na spory, które nurtują polskich przedsiębiorców. Wprowadzenie tej instytucji do wymiaru sprawiedliwości ma też być formą pewnej aktywizacji społeczności lokalnej.

Sadzając je na sali rozpraw jako głos doradczy, od razu sprawiamy, że zaufanie do wymiaru sprawiedliwości do wydawanych wyroków może wzrosnąć.

Proponujemy wprowadzenie instytucji sędziego handlowego do rozstrzygnięć podejmowanych w sądach okręgowych w pierwszej instancji, tam bowiem z mocy przepisów rozstrzygane są sprawy najbardziej skomplikowane ze względu na najwyższą wartość sporu.

Co ważne, wprowadza się też górną granicę wieku w ślad za rozstrzygnięciami. Miałem wczoraj spokojniejszy wieczór. górną granicę wieku, wzorowaną na rozstrzygnięciach dla ławników opisanych w ustawie o sądach powszechnych. Istotny jest wybór sędziów handlowych. Proponujemy, żeby sędziowie handlowi wybierani byli przez sejmiki województw, przez radnych tych sejmików, czyli przez samorządowców, którzy cieszą się ogromnym zaufaniem, mają mocną, bezpośrednią legitymację od swoich mieszkańców. To radni sejmikowi odpowiedzialni byliby za przeprowadzenie transparentnego procesu wyborczego.

To zapewni nie tylko większą transparentność, ale także większy mandat zaufania do wybranego sędziego handlowego. W przeciwieństwie do sędziego zawodowego wybór ten nie byłby dożywotni.

Jest to obwarowane pewnymi bezpiecznikami. Przede wszystkim, co najważniejsze, takie odwołanie mogłoby nastąpić nie z inicjatywy samych radnych, ale tylko i wyłącznie na wniosek prezesa sądu okręgowego, po zaopiniowaniu tego wniosku przez kolegium sądu, tak żeby ta decyzja faktycznie nie była arbitralna.

Projekt ustawy też w sposób jednoznaczny te kwestie przesądza, w szczególności że sędziowie handlowi nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić innej działalności (Dzwonek), której. Pojawiają się pytania i wątpliwości osób, które zapoznały się z projektem: a co w takiej sytuacji, jeżeli przedsiębiorcy wykorzystywaliby swoje stanowisko do wyciągania pewnych informacji od innych przedsiębiorców, którzy toczą spór przed sądem.

Ba, jest dużo większe zaufanie do tego typu rozstrzygnięć niż do rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pragnę zaapelować, żebyśmy spokojnie nad tym projektem procedowali, bo jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości czy natury konstytucyjnej, czy natury praktycznej, to oczywiście jesteśmy skłonni do przyjęcia jakichś zmian i poprawek. Niemniej jednak miejmy odwagę wymiar sprawiedliwości zmieniać w sposób odważny, ale nie, jak często na tej sali sejmowej słyszymy, w sposób szalony. Dziękuję serdecznie. Proszę pana posła Krzysztofa Paszyka o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy zawartego w druku nr 1762. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Panie, Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów i Konserwatyści projektu dotyczącego powołania sądów pokoju. Na początek może kilka słów o okolicznościach, w jakich ten projekt powstał. Nie jest to projekt napisany tylko w gronie naszych posłów czy ekspertów, ten projekt urodził się w drodze daleko idących konsultacji społecznych. Dzięki uprzejmości pana marszałka Piotra Zgorzelskiego kilkukrotnie tu, w parlamencie, odbyły się posiedzenia okrągłego stołu dotyczące właśnie potrzeb i miejsc, gdzie te zmiany w sądownictwie są najbardziej potrzebne. W tych konsultacjach również, co chciałbym bardzo podkreślić, wzięły udział organizacje zrzeszające osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości, osoby, które bezsilnie przez wiele ostatnich lat próbowały walczyć o sprawiedliwość, ale ten system wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo im nie do końca na to pozwalały. Dzięki tym wielu godzinom rozmów właśnie wskazano na to, że przywrócenie do sądownictwa polskiego instytucji sądów pokoju i sędziów pokoju jest jedną z tych najbardziej oczekiwanych właśnie przez osoby, które zderzyły się z wieloma utrudnieniami, z wieloma barierami, jeśli chodzi o dostępność, jeśli chodzi o możliwości walki o sprawiedliwość przed polskimi sądami. Dzięki temu powstał projekt ustawy, który mam przyjemność zaprezentować. Projekt ten wywodzi się, tak jak to padło z ust obydwu przedmówców prezentujących również bardzo podobne projekty, po pierwsze, właśnie z braku zaufania, z pewnej niemocy, jeśli chodzi o dostęp do wymiaru sprawiedliwości, do sądów, po drugie, ze zjawiska, które obserwujemy z niezwykłym zaniepokojeniem, tj. wydłużających się i to właściwie w każdej kategorii spraw, wydłużających się terminów rozpatrywania spraw przed polskimi sądami. Wiele osób właśnie z tych przywołanych przeze mnie środowisk pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości bardzo zaufało dzisiaj rządzącym, którzy odpowiadają za wymiar sprawiedliwości.

Przechodząc do projektu, który mam przyjemność zaprezentować, powiem, że jego założeniem jest to, aby sądy pokoju odciążyły sądownictwo powszechne poprzez przejęcie znacznej części spraw należących do właściwości sądów rejonowych, zapewniając w ten sposób szybsze i bardziej sprawne prowadzenie postępowań sądowych. Rokrocznie rośnie przewlekłość postępowań przed sądami rejonowymi. O ile w 2015 r. terminy rozpraw były wyznaczane z 3-miesięcznym okresem oczekiwania, o tyle obecnie termin oczekiwania na rozprawy zwiększył się ponaddwukrotnie.

Projektowane rozwiązanie zakłada powołanie sądów pokoju we wszystkich powiatach, miastach na prawach powiatu i dzielnicach gminy Warszawa.

Proponuje się, aby kandydaci na sędziów pokoju byli wybierani w wyborach powszechnych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, powiatów oraz dzielnic gminy Warszawa. Sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach powszechnych odbywających się wraz z wyborami samorządowymi. To jest rozwiązanie, które ma racjonalizować koszty wyboru sędziów. Osoba wybrana przez obywateli będzie siłą rzeczy o wiele bardziej niezależna od pozostałych władz, posiadając własny mandat wyborczy, a tym samym poparcie obywateli, niż osoba powoływana przez zamknięte gremia.

To też jest wyróżnik na tle pozostałych projektów. Uważamy, że zapewni to sprawność funkcjonowania projektowanej instytucji oraz szybkie załatwianie prowadzonych postępowań, co jest jednym z założeń projektodawców. Projekt zakłada, że sądy staną się sądami I instancji w sprawach najprostszych, o najniższym ciężarze gatunkowym. Proponujemy przekazanie sądom pokoju następujących kategorii spraw: spraw o wykroczenia; spraw karnych zagrożonych karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku; jak również następujących spraw cywilnych: o prawa majątkowe, świadczenie, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł; spraw, o których mowa w dziale II tytułu II Kodeksu cywilnego, tj. o roszczenia z rękojmi lub gwarancji, jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 2 tys. zł; sporów z powództwa najemcy lokalu mieszkalnego przeciwko wynajmującemu; spraw określonych w art. 144 Kodeksu cywilnego, tj. spory sąsiedzkie o tzw. immisje; sporów z czynów niedozwolonych, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, a dochodzone przez powoda roszczenie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; sporów o naruszenie posiadania, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł; sporów o wydanie własności i o ochronę własności, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. Kandydaci na sędziów pokoju nie będą uprawnieni do prowadzenia kampanii wyborczej, bowiem mogłoby to stać w sprzeczności z ich niezawisłością. Sądy pokoju mają zostać usytuowane w strukturze organizacyjnej sądów rejonowych. Wyraża się to w przyjętej konstrukcji, wedle której będą one miały siedzibę w siedzibie sądu rejonowego, zaś ich finansowanie będzie dokonywane z budżetu państwa w części przekazanej corocznie na finansowanie sądownictwa powszechnego.

W tym zakresie proponuje się jednak modyfikację polegającą na określeniu wyższej granicy wieku, czyli 35 lat. Przewiduje się, że funkcjonowanie sądów pokoju spowoduje znaczne przyspieszenie postępowań prowadzonych przez sądy powszechne. W ocenie autorów projektu zaproponowane w nim rozwiązania, zwłaszcza wybór kandydatów na sędziów pokoju w wyborach powszechnych, spowoduje zwiększenie zaufania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Dotychczas wprowadzane reformy wymiaru sprawiedliwości wielokrotnie uzasadniane są potrzebą przybliżania wymiaru sprawiedliwości do ludzi i zwiększania udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Uzasadnienie takie nie zmienia jednak faktu, że ustawy uchwalane przez Sejm w ostatnich latach w żaden sposób nie spełniały tej funkcji. Projektowana ustawa ma być też swego rodzaju odpowiedzią ustawodawcy na dokonaną w 2001 r. na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego likwidację kolegiów do spraw wykroczeń i przekazanie rozpoznawanych przez nie spraw wydziałom karnym sądów rejonowych. Ten zabieg pozostawał oczywiście w zgodzie z konstytucją, w której wymiar sprawiedliwości został powierzony wyłącznie sądom. Tymczasem kolegia do spraw wykroczeń były organami pozasądowymi i jako takie nie mieściły się w konstytucyjnej konstrukcji władzy sądowniczej. Niemniej zabieg ten spowodował powstanie znacznego obciążenia sądów rejonowych, wpływając na postępującą w kolejnych latach przewlekłość postępowań sądowych. Celem długofalowym, który postawił sobie projektodawca jako konsekwencję projektowanych regulacji, stanowiącym niejako efekt celu doraźnego w postaci przyspieszenia postępowań sądowych, jest osiągnięcie znacznego wzrostu zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Zaufanie to będzie możliwe do odbudowania jedynie w sytuacji, gdy obywatele uzyskają rzeczywisty wpływ w procesie wskazywania kandydatów na sędziów pokoju oraz gdy postępowania sądowe ulegną przyspieszeniu. Na takie rozwiązania oczekują obywatele, co wynika z licznych sondaży i badań społecznych. W imieniu wnioskodawców chcę powiedzieć, panie marszałku, Wysoka Izbo, że liczymy na dobrą, konstruktywną dyskusję nad wszystkimi projektami oraz na to, że nie ulegną one jakiemuś długotrwałemu mrożeniu na kolejnym etapie i że będziemy mogli w realnym, niedługim terminie doprowadzić do powstania całościowej ustawy dotyczącej sądów pokoju. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Na pewno będziemy procedowali nad tymi projektami w pokoju. Bardzo proszę panią poseł Annę Marię Żukowską o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy zawartego w drukach nr 1763 i 1763-A. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! Rozmawiamy dzisiaj głównie o sądach pokoju, a także o sędziach handlowych. Ale porozmawiajmy szerzej o wymiarze sprawiedliwości. Skąd wzięła się potrzeba tych wszystkich projektów? Wymiar sprawiedliwości - mimo tego, co deklarowało Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie, że to jest naczelnym celem zmian, które przeprowadza - nie działa, nie funkcjonuje sprawnie. To dotyka każdego obywatela, na najniższym poziomie. W wielu sprawach, sprawach istotnych życiowo, takich jak sprawy w sądzie w wydziałach pracy, na pierwszą rozprawę oczekuje się minimum rok. A to dotyczy np. zwolnień z pracy, kiedy pracownik chce udowodnić, że został niesłusznie zwolniony, m.in. np. dyscyplinarnie, i nie ma takiej szansy przez ponad rok. To nie poprawia w żaden sposób życia Polek i Polaków. W przypadku zwykłych zdarzeń, takich jak stłuczka, też te rozprawy są zwoływane dopiero po bardzo długim czasie, np. właśnie po roku, kiedy świadkowie już nic z tego nie pamiętają. To naprawdę nie ma sensu. To nie działa, to po prostu nie działa. Te zmiany, które przeprowadzacie, niszczą polską praworządność, niszczą naszą demokrację, a w żaden sposób nie pomagają panu Kowalskiemu - panu posłowi też Kowalskiemu, który tutaj siedzi przede mną i słucha.

Dlatego wszystkie te projekty w moim rozumieniu zmierzają do poprawy tej sytuacji. Nasz projekt jest projektem, który został przedłożony - znaczy, przedłożone były założenia do tej ustawy - jeszcze w poprzedniej kadencji. Złaszaliśmy go jako pierwsi. Chodzi o to, żeby wprowadzić tę instytucję, wprowadzić coś, co rzeczywiście pomoże Polkom i Polakom dochodzić sprawiedliwości w sposób szybki i w sposób efektywny. Przyspieszenie postępowań, odciążenie sądów właśnie od tych spraw bagatelnych jest istotą projektu przedłożonego przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Ma to również wzmocnić demokratyczny wymiar legitymacji wymiaru sprawiedliwości, żeby obywatele i obywatelki czuli, że te orzeczenia są rzeczywiście w ich imieniu, że te orzeczenia są dla nich i że wymiar sprawiedliwości nie jest odległy, nie jest nieosiągalny, tylko jest tu, blisko, w mojej gminie. Dlatego proponujemy, żeby wyłanianie sędziów pokoju odbywało się z udziałem społeczności lokalnych, czyli mieszkańców, którzy popierają danego kandydata, i ten wybór miałby się dokonywać przez rady gmin. Kandydaci, którzy spełnialiby warunki, które zaraz wymienię, musieliby przedłożyć minimum 50 podpisów za poparciem swojej kandydatury i ta kandydatura byłaby rozpatrywana przez radę gminy. Jakie wymagania przewidujemy dla kandydatów? Przewidujemy, po pierwsze, wiek między 31. rokiem życia a 65. rokiem życia, wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie minimum 1 roku w zakresie legislacji - to może być praca w organach samorządowych, to może być wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego. Co więcej, uważamy, że rada gminy, która powinna przeprowadzić publiczne przesłuchanie kandydatów, powinna wyłonić w głosowaniu tajnym dwóch, dwoje spośród nich i przedstawić te kandydatury zgromadzeniu ogólnemu sądu rejonowego właściwego terytorialnie dla danej gminy, po to żeby zachować ten element, że to sędziowie wybierają sędziów. My tu nie będziemy legitymizowali, jak w jednym z tych projektów, neo-KRS-u. To sędziowie mają się wybierać i się powoływać.

Uważamy, że ślubowanie, które sędzia pokoju składa wobec prezesa właściwego sądu rejonowego, również powoduje takie nawiązanie łączności między powszechnym wymiarem sprawiedliwości a sędziami pokoju - którzy oczywiście zgodnie z naszym założeniem nie są sędziami w rozumieniu konstytucji. To są osoby, które podobnie jak asesorzy sądowi wykonują ograniczoną liczbę powierzonych im zadań, w bardzo ograniczonym zakresie. W związku z tym naszym zdaniem nie ma tutaj konieczności zmiany konstytucji. Absolutnie nie widzimy takiej potrzeby, w naszym projekcie też tego nie przewidziano.

Proponujemy województwo opolskie i województwo kujawsko-pomorskie.

Chcielibyśmy sprawdzić, jak to działa, żeby móc ewentualnie poprawić pewne niedociągnięcia, które najpewniej by pojawiły. Zawsze tak jest z nowymi rzeczami, które się wprowadza.

Myślę, że będziemy w stanie pracować nad tymi ustawami w komisji. Chciałabym, żeby to była praca cywilizowana - tu zwracam się do przewodniczącego mojej komisji pana Marka Asta - żeby to nie było o godz. 2 w nocy, żebyśmy mogli sobie spokojnie porozmawiać o tych projektach, bo jak widzę, z wielu środowisk politycznych płynie potrzeba zmiany idącej w tym kierunku. Różnimy się na pewno, jeżeli chodzi o zakres tego, o tryb wyboru - to jest moja główna bolączka odnośnie do projektu pana prezydenta - niemniej jednak widzimy tę potrzebę. Widzi ją bardzo dużo różnych środowisk politycznych: lewica, prawica, centrum, PSL.

Dziękuję serdecznie.

Ja też.

Otwieram dyskusję.

Dobrze mówię? Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec zgłoszonych projektów ustaw o sędziach pokoju. Tak jak na tej sali już padło, jest to instytucja niezwykle oczekiwana i zapewne oczekiwana z życzliwością przez środowiska prawnicze, środowiska polityczne. Przede wszystkim jest oczekiwana przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego jest oczekiwana? Wynika to z niedoskonałości naszego wymiaru sprawiedliwości, bolączek, które nasze sądownictwo dotykają, przede wszystkim oczywiście przewlekłości postępowań wynikających też z natłoku spraw, wpływu spraw do sądów powszechnych, szczególnie spraw o drobnym charakterze. Dotyczy to zarówno spraw cywilnych, jak i spraw karnych.

Ona od dziesiątek lat funkcjonuje w systemie anglosaskim, ale też - jak w uzasadnieniu do projektu prezydenckiego wskazano - w niektórych państwach europejskich, np. w Szwajcarii, zbliżone rozwiązania są przyjmowane. Istota tej instytucji, istota sędziego pokoju przede wszystkim polega na tym, że pochodzi on z powszechnego wyboru - i to też państwo wielokrotnie podkreślaliście, że to stanowi jego atut, to, że posiada mandat z wyboru, mandat społeczny do sprawowania swojej funkcji. On musi wynikać też oczywiście z zaufania do osoby, która ten mandat będzie sprawować. Ale to jest też postulat obywateli, którzy powiadają: no chcemy mieć zaufanie do sędziów, którzy mają rozstrzygać o naszych sprawach, o sprawach życiowych, mają rozstrzygać pomiędzy nami spory. Stąd też istotnie można się zapytać: Dlaczego do tej pory nie udało się znaleźć konsensusu pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi, aby tę instytucję do polskiego porządku prawnego wprowadzić? Tak jak powiedziałem, samo rozwiązanie w postaci sądów pokoju, sędziów pokoju jest oczekiwane i wyrazem wyjścia naprzeciw temu oczekiwaniu społecznemu jest fakt, że dzisiaj debatujemy nad nie tylko przedłożeniem prezydenckim, ale również projektami zgłoszonymi przez kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej i Lewicy. Trzeba powiedzieć, że oczywiście najpełniejszy projekt został złożony przez prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie zarówno opisu samej instytucji sędziego pokoju, jak i procedur, które są opisane w tym drugim projekcie - Przepisy wprowadzające. Trudno się też nie zgodzić z tymi propozycjami, które w projekcie są zawarte, co do zarówno powszechności wyborów, jak i zakresu spraw, którymi sędzia pokoju czy sądy pokoju mają się zajmować, a także warunków, jakim powinien odpowiadać sędzia pokoju. Można się zastanawiać nad tym, czy tylko i wyłącznie jedna kadencja, bo sędzia pokoju, który 6 lat wykonuje dobrze swoją pracę, zyskuje zaufanie mieszkańców swojego rejonu, okręgu, w którym orzeka, czy nie byłoby dobrze, aby miał szansę być wybrany na kolejną kadencję.

Będzie na to czas podczas prac w komisji. Najbardziej zbliżony do projektu prezydenckiego jest projekt Koalicji Polskiej. Myślę, że w przypadku wielu rozwiązań będzie zgoda, będzie można wiele dopracować i w zasadzie nie widzę jakiejś dużej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma projektami, w szczególności, że jeden i drugi zakłada powszechny wybór sędziów pokoju. Projekt Lewicy zakłada wybór pośredni - i to jest jakby słabość tego projektu, bo wybór pośredni nie odpowiada już temu oczekiwaniu społecznemu, że lokalna społeczność będzie wybierała swojego sędziego pokoju. Można nawet dyskutować, czy kryterium mieszkańców, czy kryterium spraw, które są w sądzie, którymi sąd rejonowy jest obciążony, które będą przypadały na sędziego pokoju. Ale tak jak powiedziałem, to już szczegóły. Natomiast projekt Koalicji Obywatelskiej w istocie dotyczy jednak zupełnie innej instytucji.

Zdajemy sobie sprawę, że w tym pionie sądownictwa też są problemy, jest też przewlekłość postępowań i duża komplikacja materii, którymi te sądy się zajmują. Mając na uwadze i oczekiwania społeczne, i chęć rozwiązania tych problemów, które leżą u podstaw złożenia projektów o sędziach pokoju, w imieniu klubu wnoszę o przekazanie projektów do dalszego procedowania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Dzisiaj pracujemy nad ustawą, która, mam wrażenie, jest efektem pewnej obsesji pana prezydenta Dudy, obsesji, która zmierza w stronę nie tylko zniszczenia niezależnych od polityków sądów, ale nade wszystko do pozbawienia Polaków dostępu do profesjonalnego wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa jest niekonstytucyjna, ale do tego prezydent przyzwyczaił nas już od pierwszych tygodni swojej kadencji. Polska konstytucja nie przewiduje sądów pokoju, a obywatele mogą w wymiarze sprawiedliwości uczestniczyć, ale nie sprawować go samodzielnie. Dzisiaj nie potrzebujemy kolejnej niekonstytucyjnej, niechlujnej, źle przygotowanej ustawy. Dzisiaj najważniejszą sprawą dla Polski jest likwidacja tzw. Izby Dyscyplinarnej oraz neo-KRS-u. Projekt, o którym rozmawiamy, jest efektem brudnego politycznego dealu i zasłoną dymną dla PiS-owskiego uporu i kunktatorstwa. Prezydent powinien teraz wnieść projekt ustawy realizującej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Atutami nowego prawa, jak słyszymy od projektodawców, miały być bezpośrednie wybory sędziów pokoju. Tyle że to jest kłamstwo. Po wyborze sędzia pokoju będzie bowiem weryfikowany przez upolitycznioną neo-KRS i powoływany lub nie przez prezydenta. Jakby tego było mało, to prokurator będzie mógł zablokować każdą kandydaturę. Wystarczy, że rozpocznie postępowanie wobec kandydata i w ten prosty sposób wyeliminuje niewygodnego kandydata na sędziego pokoju. Jeśli ktoś sądzi, że nie będzie takiej pokusy w politycznie i ręcznie sterowanej prokuraturze Ziobry, to jest naprawdę fantastą. Wybory sędziego pokoju będą farsą, populistyczną przykrywką dla dewastacji niezależności wymiaru sprawiedliwości, bo przecież taki cel ma ta ustawa. Jeśli myślicie państwo, że celem tej ustawy jest wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości obywateli cieszących się poparciem lokalnych społeczności, to was oszukano. Największe szanse na sprawne przeprowadzenie kampanii wyborczej będą mieli kandydaci posiadający silne wsparcie struktur, także partyjnych, które pomogą zebrać pieniądze, zorganizują szkolenia, zorganizują spotkania z kandydatem. Ustawa przewiduje ponad 4 tys. nowych etatów nieprofesjonalnych sędziów. To ludzie, którzy, nie miejmy złudzeń, przynajmniej w części będą wskazywani przez lokalnych polityków obecnej władzy. Co więcej, sami politycy, członkowie partii, będą mogli kandydować na sędziów pokoju. Dopiero po wyborze, po 14 dniach będą mogli zrezygnować z członkostwa. Jak Piotrowicz, Pawłowicz przechodzili z ław poselskich do Trybunału, tak np. lokalni działacze prosto z foteli radnych przejdą do sądów pokoju i nadal będą wdzięczni swojej partii. Miało być szybciej, sprawniej, jednak ta ustawa pogłębi tylko chaos w wymiarze sprawiedliwości. Niekonstytucyjność wielu przepisów tej ustawy i udział upolitycznionej neo-KRS w wyborze sędziów sprawią, że obywatel, wychodząc z sądu pokoju, nie będzie miał pewności, czy wyrok wydał sędzia, czy to w ogóle wyrok, czy to jest świstek papieru, który z powodzeniem będzie można kwestionować w postępowaniach przed niezależnymi sądami. O czym będą decydowali sędziowie pokoju? Oskarżenie o kradzież to jest bardzo poważna sprawa. Można trafić do więzienia, stracić dobre imię na lata, można tu przegrać całe życie. Czy oddalibyśmy swoje życie i zdrowie w ręce felczerów, a nie lekarzy? W sprawach cywilnych to są np. alimenty. Czy chcielibyście opowiedzieć, dlaczego były mąż nie chce łożyć np. na dziecko jakiejś byłej, nie wiem, PiS-owskiej radnej, której minister sprawiedliwości może zdjąć obowiązek zachowania tajemnicy? Prezydencki projekt ustawy o sędziach pokoju to jest po prostu prawny bubel, który nikomu życia nie ułatwi. 70 stron regulacji, wyłączeń, wyjątków, błędy legislacyjne, wewnętrzne sprzeczności. Naprawdę wstyd, że po tylu miesiącach z Pałacu Prezydenckiego wychodzi projekt, który ma mniejszą wartość niż papier, na którym został wydrukowany. Tylnymi drzwiami wprowadzacie po prostu zwiększony nadzór polityczny nad wymiarem sprawiedliwości. Neo-KRS będzie tych sędziów weryfikował, prezydent powoływał, jak mu się spodobają, a minister Ziobro będzie przenosił, zwalniał z tajemnicy, wydawał polecenia administracyjne. Wysoki Sejmie! Powtórzę: dzisiaj Polacy nie potrzebują kolejnej niekonstytucyjnej, niechlujnej i szkodliwej ustawy.

Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pani marszałek. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedłożone prezydenckie projekty dotyczące sędziów pokoju są wyrazem magicznego myślenia, że oto dorzucimy jakieś rozwiązanie i będzie cud, i wszystko się rozwiąże. Otóż nic bardziej mylnego. Jeżeli ktoś myśli, że poprawi sytuację w wymiarze sprawiedliwości rozwiązaniami bazującymi na małych wymaganiach merytorycznych, małym lub żadnym doświadczeniu proceduralnym zamiast na profesjonalizmie i specjalizacji sędziów, to jest w błędzie. Tym projektem prezydenckim PiS robi wszystko, by zniszczyć niezależność sądów, a twierdzenie, że sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, to, proszę państwa, czysta fikcja i chwyt reklamowy, by przekonać obywateli do pomysłu. Art. 3 projektu o sądach pokoju mówi o wyborach powszechnych, ale w art. 20 i 21 jest mowa o powołaniu na stanowisko sędziego pokoju, na wniosek KRS, przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzi się zatem pytanie, kto tak naprawdę powołuje sędziów. W art. 12 pkt 24 ustawy - Przepisy wprowadzające dodaje się do Kodeksu wyborczego przepisy dotyczące powszechnych wyborów sędziów pokoju.

Taki zapis powoduje, że prezydent będzie miał możliwość odmowy powołania kandydata mimo uzyskania przez niego poparcia w wyborach powszechnych. Czy to będzie jedna, dwie czy trzy kadencje, to i tak będzie to naruszenie art. 179, z którego wynika, że sędziowie powoływani są na czas nieoznaczony, co również jest wyrazem niezawisłości. Tak więc ok. 4 tys. wybranych osób przejdzie przez neo-KRS, a to oznacza, że państwo PiS robi wszystko, by zniszczyć niezależność sądów i upolitycznić te wybory. Jakby tego było mało, kandydować na sędziów pokoju mogą osoby należące do partii politycznych. Osoba, która została wybrana, dopiero w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów powinna złożyć oświadczenie o rezygnacji z przynależności do partii politycznych. Projektodawcy, uzasadniając te projekty, powołują się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., ale, powołując się na to orzeczenie, cytują wygodny dla nich fragment uzasadnienia. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że nie ma znaczenia, czy chodzi o sprawy mniejszej, czy większej wagi. W każdym przypadku sąd powinien być niezależny, a sędziowie niezawiśli. Skoro sędziowie mają być wybierani w wyborach powszechnych, a następnie rozstrzygać w sprawach na terenie swoich okręgów wyborczych - pamiętajmy przy tym, że obywatele mogą dokonywać wpłat na kampanię - to czy będzie można uznać, że będą sądem niezależnym? To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, o którym powiedziałam, jest swoistym memento dla projektodawców opiniowanych ustaw w zakresie konsekwencji powoływania do życia instytucji niezgodnej z konstytucją. I jeszcze jedno, proszę państwa - koszty. Ok. 4 tys. sędziów pokoju, mniej więcej 1300 asystentów i ponad 7800 pracowników administracji. Wiecie państwo, jaki to będzie koszt w ciągu 10 lat? Gdyby chociaż część przeznaczyć na wymiar sprawiedliwości, na zwiększenie liczby pracowników administracyjnych dobrze opłacanych, na jednego asystenta dla sędziego, na odpowiednią liczbę referendarzy i sędziów, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i ilość wpływających spraw, to naprawdę sądy działałyby dobrze. Dobra procedura, dobra informatyzacja, profesjonalizm sędziów, wręcz specjalizacja, bo trudno, by sędzia znał się wszystkim - to są drogi do rozwiązania problemów wymiaru sprawiedliwości. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli mówimy o czynniku społecznym, to mamy dzisiaj ławników.

Mediacja, proszę państwa, to bardzo ważny sposób rozwiązywania problemów wymiaru sprawiedliwości. Lepsza najgorsza ugoda niż najlepszy wyrok, bo jest zawierana pomiędzy stronami.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czas na Lewicę. Pan poseł Andrzej Szejna, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o sędziach pokoju ma przybliżyć sądy do obywateli. Ma stać się urzeczywistnieniem udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - w przeciwieństwie do działań Zbigniewa Ziobry, który doprowadził do częściowego wyeliminowania ławników z orzekania w czasie pandemii. Ustawa Lewicy i prezydenta ma być remedium dla wymiaru sprawiedliwości wobec zniszczeń, których przez ostatnie 6 lat dokonał Zbigniew Ziobro i jego ekipa. Dokonali oni destrukcji wymiaru sprawiedliwości. Ta destrukcja spotkała się z reakcją klubu Lewicy. Polacy mają prawo oczekiwać, że ktoś, kto będzie sądził ich sprawy, będzie również znał miejscowe realia, a nie że prezesa sądu odwoła czy powoła faksem minister sprawiedliwości. Zaskoczę was i zacytuję Kornela Morawieckiego, który kiedyś powiedział: „Być może polski wymiar sprawiedliwości wymaga więcej sprawiedliwości, a mniej prawa. Potrzeba więcej empatii. Ważna jest ludzka wrażliwość” To właśnie sędziowie pokoju mają wnieść empatię i ludzką wrażliwość do wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo mają wzmocnić demokratyczną legitymację wymiaru sprawiedliwości, sprzyjać zwiększeniu społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, wzmocnieniu jego autorytetu i akceptacji dla wydawanych orzeczeń. Dziś obywatel niewiarygodnie długo czeka na rozpoznanie sprawy przez sąd i jest to wina Zbigniewa Ziobry. Musimy coś z tym zrobić. A najprostszym i najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie sędziów pokoju. Zobrazuję dane statystyczne: przecież 11 miesięcy oczekiwania na przywrócenie do pracy bezprawnie zwolnionego członka związków zawodowych to o 11 miesięcy za wiele. Oczywiście nie mówimy o Warszawie, bo tu w tym terminie może nie odbyć się nawet pierwsza rozprawa. Nie ma spraw mniej lub bardziej ważnych, wszystkie są ważne i wszystkie powinny być szybko rozpatrywane. Wprowadzenie sędziów pokoju ma na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw, tym samym przywrócenie elementarnego poczucia sprawiedliwości. Zwiększenie liczby sędziów, do których ludzie będą mieć zaufanie, pozwoli na urealnienie środków ochrony prawnej. Projekt Lewicy i projekt prezydencki co do zasady są zbieżne, a różnice są niewielkie - przykładowo czas trwania kadencji, zakres spraw, którymi mają zająć się sędziowie, dodatkowe szkolenie przed rozpoczęciem pracy, które proponuje Lewica - poza dwoma zasadniczymi kwestiami: sposobem wyboru sędziów i ich liczbą. Lewica proponuje wybór sędziów pokoju poprzez zgromadzenie sędziów sądu rejonowego w jawnym głosowaniu spośród kandydatów przedstawionych przez radę gminy. Rada gminy lub upoważniona przez nią komisja przeprowadza publiczne przesłuchanie kandydatów. Podczas przesłuchania pytania mogą zadawać radni, mieszkańcy bez ograniczenia czasu. Lewica proponuje jednego sędziego pokoju na 30 tys. mieszkańców, a prezydent - jednego na 10 tys. mieszkańców. Wybory powszechne proponowane przez prezydenta mają wiele wad. Pierwsza, bardzo oczywista wada to koszty. Ile kosztują wybory, najpewniej wie pan minister Sasin, ale pamiętajmy, że głównym kosztem wyborów są pensje członków komisji. Według naszych szacunków koszt przeprowadzenia takich wyborów to ok. 300 mln. Nie upolityczniajmy tych wyborów, nie zmuszajmy, by w kampanii wyborczej kandydaci prześcigali się w obietnicach typu: skażę każdego, dożywocie za kradzież. Dość populizmu funduje nam na co dzień Zbigniew Ziobro. W naszej ocenie 1200 sędziów pokoju będzie stanowiło wystarczające wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości. Proponowane przez prezydenta 3800 sędziów jest liczbą nadmierną. Szanowni Państwo! W imieniu klubu parlamentarnego Lewica wnosimy o dalsze procedowanie nad przedłożonym projektem. Dziękuję. Proszę bardzo, pan poseł Krzysztof Śmiszek. Wysoka Izbo! W imieniu klubu Lewicy przedstawiam stanowisko naszego klubu w odniesieniu do poselskiego projektu ustawy o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wychodzi naprzeciw konstytucyjnej zasadzie wzmacniania prawa społeczeństwa obywatelskiego do uczestnictwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Powinni po prostu mieć realny wpływ na wymierzanie sprawiedliwości, czyli na kształtowanie stosunków społecznych oraz na stosowanie prawa. Od lat bolączką polskiego sądownictwa są przeciągające się procesy, długie wyczekiwanie na wyrok, czasami tak długie, że nawet otrzymanie orzeczenia niewiele zmienia sytuację prawną strony. Sędziowskie biurka uginają się coraz bardziej od nadmiaru spraw, a często postępowania gospodarcze przeciągają się z uwagi na wysoki stopień skomplikowania zagadnienia. Zaproponowany projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych z jednej strony jest ciekawą próbą oddania w ręce obywateli decyzji w postępowaniach o charakterze gospodarczym, z drugiej - to dobry przykład odciążania i wzmacniania potencjału polskich sądów i polskich sędziów. Jak podnoszą projektodawcy, projektowana ustawa stanowi propozycję urzeczywistnienia ogólnej normy konstytucyjnej o uczestnictwie obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Dlaczego obywatelscy sędziowie handlowi to interesująca propozycja? Żyjemy w bardzo szybko zmieniającym się świecie - nowe technologie, nowe techniki współpracy gospodarczej, nowe sposoby produkcji czy, ogólnie rzecz ujmując, niezwykle szybko zmieniające się uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Nie zawsze zawodowi sędziowie nadążają za tymi zmianami. Nie każdy jest w stanie śledzić zmieniające się trendy prowadzenia biznesu. Obecność w składzie orzekającym osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, może być jedynie wzmocnieniem dla profesjonalnych sędziów, którzy muszą mierzyć się z ciągle zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Funkcja obywatelskich sędziów handlowych w założeniu ma być sprawowana przez obywateli będących przedsiębiorcami i służyć uaktywnieniu tych osób jako członków społeczności lokalnej, a także stworzyć możliwość skorzystania z ich wiedzy oraz doświadczenia życiowego i zawodowego. To ciekawa propozycja, chociaż klub Lewicy będzie zgłaszał w trakcie prac parlamentarnych pewne zmiany czy pewne propozycje dodatkowych rozwiązań, np. w celu zagwarantowania pewności i szybkości postępowania dodatkowe kryterium wykształcenia prawniczego kandydata na obywatelskiego sędziego handlowego. Klub Lewicy, mając na uwadze takie wartości jak uczestnictwo czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie profesjonalnych sędziów poprzez dostarczanie im branżowej wiedzy z zakresu obrotu gospodarczego, popiera przedstawiony projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych i postulujemy przesłanie go do dalszych prac do odpowiedniej komisji sejmowej. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Teraz poproszę pana posła Jana Szopińskiego z klubu parlamentarnego Lewica. Panie pośle, ma pan 3 minuty, więc proszę się nie spieszyć. Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak powszechnie wiadomo, ustawa o sędziach pokoju z druku nr 1761 jest ceną, jaką PiS płaci panu posłowi Kukizowi za udzieloną pomoc. Chciałbym zadać pytanie pomysłodawcy wprowadzenia sędziów pokoju w ramach tego druku, bo nasi wyborcy pytają, czego spodziewacie się państwo po dopuszczeniu do orzekania ludzi bez doświadczenia i kierunkowego wykształcenia. I pytanie drugie, na które też oczekujemy odpowiedzi, żeby móc dobrze pracować nad tym projektem: Kto będzie rozstrzygał - używając nomenklatury partii rządzącej - o kryształowości charakterów kandydatów na sędziów? Chciałbym też zapytać, jaki będzie system weryfikacji ich wiedzy oraz kwalifikacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze!

Pozwolę sobie jedynie wskazać na pewne odrębności w ramach tej debaty.

Reasumując, chciałbym w imieniu Koalicji Polskiej - PSL, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów wnieść o skierowanie wszystkich czterech projektów do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Krzysztofa Bosaka, koło

Wysoki Sejmie! Bez wątpienia mamy do czynienia z kryzysem polskiego sądownictwa.

Natomiast projekty te są próbą poszukiwania wyjścia z kryzysu. Zanim zaczniemy mówić o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących powołania sędziów pokoju, chcę powiedzieć dwa, trzy słowa ogólnie. Wydaje mi się, że warto to powiedzieć, zanim będziemy omawiać dokładnie, kto powinien być na sędziego powołany, gdyż rola sędziego zaciera się. Coraz częściej sami sędziowie widzą swoją rolę nieco inaczej, bardziej politycznie, mniej jako pełniących pewną służebną funkcję wobec społeczeństwa, tzn. właśnie tych, którzy mają sprawnie i sprawiedliwie rozstrzygać spory na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a bardziej jako tych, którzy mają wspomagać obóz władzy, np. pracując na delegacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości i angażując się w rozgrywki w swoim własnym środowisku, albo jako tych, którzy mają zwalczać obóz władzy, dlatego że w jakichś kwestiach politycznych się nie zgadzają albo np. że mają stać na straży jakichś doktryn, jakichś koncepcji politycznych, które nie są skodyfikowane bezpośrednio w przepisach prawa, np. związanych z prawem międzynarodowym, związanych z prawem unijnym, związanych z pewnymi szczegółowymi możliwymi interpretacjami konstytucji, które jednak interpretacyjnie są zapisane w przepisach ustawowych, a nie konstytucyjnych, są po prostu kwestią pewnego mniemania, że jest tak albo że jest inaczej. Okazuje się, że niektórzy sędziowie są gotowi nawet wprost w uzasadnieniach wyroków sądu powoływać się na różne ideologie, dlatego że uważają, że ich rola jest taka, że mają np. stać na straży jakiejś konkretnej doktryny ideowo-politycznej przeciwko jakimś innym doktrynom ideowo-politycznym, podczas gdy nic o tym nie ma literalnie w przepisach prawa. To wszystko należy odrzucić. Nie jest możliwe zreformowanie sądów, jeżeli sędziowie lub ludzie aspirujący do zawodu sędziego będą okopywać się na ideologicznych stanowiskach i będą angażować się w walkę ideologiczną. Od tego jest parlament, od tego jesteśmy tutaj my, posłowie, żebyśmy spierali się o koncepcje polityczne, różne doktryny. Jeśli to się uda, to już będzie bardzo dużo. Teraz w kwestii reformy. Bez wątpienia mamy do czynienia z kryzysem sądownictwa. Główne problemy, na które zwracają uwagę ludzie, to może nawet bardziej niż niesprawiedliwość wyroków po prostu przewlekłość postępowań - smutny przykład to sprawy związane z kwestią czy to adopcji, czy praw rodzicielskich, potrafiące ciągnąć się dłużej, niż dziecko jest dzieckiem, bo mija po kilka lat, zanim zapadnie wyrok prawomocny, przechodzi to przez wszystkie instancje, więc jeżeli dotyczy to dziecka w wieku nastoletnim, to dziecko może osiągnąć pełnoletność, a sprawy jeszcze do końca nie są rozstrzygnięte, tak nie powinno być - niskie zaufanie społeczne i rzeczy, o których już mówiłem, czyli zaangażowanie polityczne, a nie czysto merytoryczne, zawodowe, sędziów. Główna wada, jaką widzę w tym projekcie, który jest tutaj przedstawiony, jest taka, że ten projekt ma się nijak do reform proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeżeli chcemy rozładować ten zator spraw, który powoduje, że tak wiele lat trzeba czekać na wyrok, to oczekiwałbym, oczekiwalibyśmy podejścia projektowego. To znaczy, że ktoś, kto przynosi konkretne projekty do Sejmu, pokaże nam, w jaki sposób np. w ciągu 2 lat, 5 lat albo dekady zaskutkuje to rozładowaniem obecnego zatoru spraw. Jeżeli mamy konkretną liczbę, np. mówi się, że ma być powołanych 3933 sędziów pokoju, to chciałbym też wyliczenia, jaką liczbę spraw ci ludzie rozpatrzą i o ile skróci się czas postępowania w innych sprawach, które nie będą przekazane sędziom pokoju. Takiego podejścia projektowego brakuje. Jeżeli założone jest wynagrodzenie na poziomie 80% pierwszego uposażenia sędziego sądu rejonowego i chcemy ludzi z wykształceniem prawniczym, z jakąś praktyką i w wieku minimum 29 lat, i jeszcze chcemy ten stan odnawiać co 6 lat, to skąd my tych ludzi weźmiemy? Skąd założenie, że uda się ich zrekrutować w takiej liczbie za takie pieniądze? Jeżeli chcemy, żeby ci ludzie byli względnie profesjonalni w tym swoim orzekaniu, żeby nabrali pewnego doświadczenia, żeby ta instytucja się zakorzeniła, to pomysł kadencyjności 6-letniej wydaje się nietrafiony.

Tymczasem sędziowie pokoju mają być zakorzenieni i wspierani przez sądy rejonowe. Na koniec słowo o propozycjach, które jako Konfederacja składaliśmy - przeorganizowanie pracy sędziów sądów powszechnych, zasada, by sędzia zajmował się jednocześnie tylko kilkoma sprawami i sprawnie i szybko je kończył, i wreszcie w szczególnych sprawach, w ramach realizacji art. 182 konstytucji, udział czynnika społecznego, w wydzielonych najważniejszych sprawach powołanie i wprowadzenie ław przysięgłych. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, panie pośle. Wysoka Izbo! Polska 2050 słynie z tego, że nie waha się sięgać po rozwiązania nowe i niestandardowe - ale nie po to żeby podążać za modą, tylko po to żeby poprawić życie Polek i Polaków. Wiem, że „sędziowie pokoju” to jest świetna nazwa, że budzi bardzo pozytywne emocje, bardzo pozytywne konotacje. Historię prawa miałem z prof. Adamem Lityńskim, jestem więc w tej niewielkiej grupie, która wie, może nie pamięta, ale wie, jak funkcjonowali sędziowie pokoju w Księstwie Warszawskim czy w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Prezentowane dzisiaj rozwiązania nawiązują jednak głównie do wzorców anglosaskich, ze swojej natury obcych polskiemu systemowi prawnemu. Mają szczytny cel - poprawić skuteczność wymiaru sprawiedliwości, przyspieszyć jego funkcjonowanie, odciążyć zawodowych sędziów. Ale nie mają szacunku dla polskiej tradycji oraz dla polskiej konstytucji - idą wbrew zasadzie nieusuwalności sędziów, burzą dwuinstancyjny tok postępowania. A przecież szybkość i sprawność postępowań sądowych można zapewnić już dziś, tu i teraz, i to stosunkowo niewielkimi środkami. W sądach jest dziś o połowę mniej asystentów sędziego niż samych sędziów. Gdyby, wzorem proponowanych projektów, każdy sędzia sądu powszechnego miał jednego czy dwoje asystentów, to postępowania z pewnością nabrałyby rozpędu. Podobnie pewnie zadziałałoby wzmocnienie kompetencyjne referendarzy sądowych czy inna prosta rzecz - zapewnienie godnych warunków pracy i płacy administracji sądowej. W naszym pomyśle na Polskę 2050 zaproponowaliśmy utworzenie sądów pierwszego kontaktu w każdym powiecie - zgodnych z ładem konstytucyjnym, obsługiwanych przez asesorów i ławników, działających w oparciu o uproszczoną procedurę, ze znacząco obniżonymi opłatami sądowymi. Z pewnością z tym projektem jeszcze wrócimy. Wśród prezentowanych rozwiązań sensownym punktem wyjścia do dalszych prac w naszej ocenie jest koncepcja Lewicy, z instytucją sprzeciwu wobec orzeczenia sędziego pokoju. Wychodzi ona ze słusznego założenia, że sędziowie pokoju nie są i nie będą sędziami w rozumieniu konstytucyjnym. Może nie w dwóch arbitralnie wybranych województwach, ale np. w kilkunastu powiatach wyselekcjonowanych w oparciu o statystyki dotyczące czasu trwania postępowań. Oczywiście w żaden sposób nie zmniejsza to wagi wyzwania, bo całość prac tak czy siak musiałaby się skończyć zmianą konstytucji po ewentualnym okresie pilotażu.

Polki i Polacy nie chcą podejmować się tej społecznej roli. Jesteśmy gotowi do dalszych prac nad projektami pod warunkiem zapewnienia ich zgodności z polską konstytucją. Ani projekt pana prezydenta, jakkolwiek dobrze dopracowany legislacyjnie i w wielu punktach ciekawy, np. w zakresie procedury wyborczej, ani koncepcja koleżanek i kolegów z PSL-u nie zapewniają tej zgodności. Równie istotnym hamulcem jest dalsze zwiększanie kompetencji upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa czy kalki z tzw. ustawy kagańcowej, czyli rozwiązania, za które nalicza się dziś Polsce 1 mln euro kary dziennie. Na marginesie, żaden z przedstawionych dziś projektów, o czym wspominał mój przedmówca, nie ma oceny skutków regulacji. Nie wiem, na jakiej podstawie szacowano liczbę spraw dla sędziów pokoju czy ich realne obciążenie. Mamy głęboką nadzieję, że w całej koncepcji sędziów pokoju nie chodzi o zaprowadzenie jakiejś formy sprawiedliwości ludowej, a po prostu o zwiększenie udziału Polek i Polaków w orzekaniu. Prawnicy wulgarnie nazywają to czynnikiem społecznym. Mocno wierzymy, że lekarstwo, które zostanie wypracowane przez Sejm, nie okaże się gorsze od samej choroby. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Jarosława Sachajkę, Kukiz’15. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Z uwagi na ograniczony czas wypowiedzi przedstawię stanowisko koła Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia w przedmiocie najistotniejszych regulacji zawartych w pięciu omawianych projektach dotyczących utworzenia sądów pokoju oraz obywatelskich sędziów handlowych. W pierwszej kolejności pragniemy podziękować panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za wszystkie dotychczasowe działania mające na celu wprowadzenie do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej instytucji sądów pokoju, w sposób znaczący wpływającej na rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Pragniemy również podziękować wszystkim klubom parlamentarnym zaangażowanym w proces legislacyjny w przedmiocie utworzenia sądów pokoju oraz zwiększenia udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ustawa o sądach pokoju jest realizacją propozycji Kukiz’15, wobec czego wyrażamy satysfakcję. Dla dobra ogółu Polaków wszyscy możemy współpracować przy jej uchwaleniu ponad podziałami politycznymi. Na wstępie należy podkreślić, że na pochwały zasługuje zdiagnozowanie przez projektodawców największego problemu postępowań przed sądami powszechnymi polegającego na przewlekłości prowadzonych postępowań.

Dlatego też utworzenie sądów pokoju, których właściwość przedmiotowa została ograniczona do spraw o stosunkowo niskim poziomie komplikacji, z pewnością jest racjonalnym rozwiązaniem tego problemu. Dodatkowo powiązanie sprawowania urzędu sędziego pokoju z procesem demokracji bezpośredniej znacząco wpłynie na zwiększenie zaufania Polaków do władzy sądowniczej. Ponadto prowadzi to do procesu utożsamiania się obywateli z wymiarem sprawiedliwości, co stanowi również niezbędny element rozwoju demokratycznego społeczeństwa. W celu zapewnienia sądom pokoju faktycznej możliwości sprawnego działania i rozwiązania problemu przewlekłości postępowań sądowych niezbędne jest optymalne określenie liczby stanowisk sędziów pokoju w zakresie ich właściwości miejscowej oraz ich strukturalne powiązanie z sądami rejonowymi. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na proces wyborczy, jeśli chodzi o sędziów pokoju, bowiem to od tej regulacji będzie uzależnione faktyczne poczucie wpływu Polaków na działania wymiaru sprawiedliwości. Uważamy, iż wybory powinny mieć charakter bezpośredni. Jednocześnie zasadna byłaby możliwość powiązania kadencji sędziów pokoju z kadencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzania wyborów sędziów pokoju w ramach jednych wyborów. Taka regulacja z jednej strony obniży koszt organizacji wyborów, zaś z drugiej strony pozytywnie wpłynie na frekwencję wyborczą, która zwiększy udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości i pozwoli większej grupie Polaków utożsamiać się z władzą sądowniczą. Chcielibyśmy również podkreślić, iż działalność sądów pokoju musi opierać się na pracy doświadczonych prawników, których status będzie możliwie zbliżony do statusu sędziego zawodowego. Z uwagi na wysokie wymagania i stosunkowo wąski krąg kandydatów należy pamiętać, iż forma wykonywania zawodu prawniczego w postaci sprawowania urzędu sędziego pokoju nie tylko powinna być atrakcyjna finansowo, lecz również powinna zapewniać stabilizację wraz z perspektywą czasową sprawowania tego urzędu.

Uważamy również, iż kandydat na sędziego pokoju nie powinien być członkiem partii politycznej w ciągu 3 lat przed wyborami oraz że nie powinno być ograniczenia w pełnieniu urzędu sędziego pokoju do jednej kadencji. Natomiast jeśli chodzi o kierunek, zakres i kompleksowość rozwiązań, to propozycja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to najlepszy projekt, w oparciu o który Wysoka Izba powinna wypracować docelową ustawę. Jednocześnie na zakończenie pragnę podziękować panu prof. Piotrowi Kruszyńskiemu, który już w ubiegłej kadencji razem z posłami Kukiz’15 opracował białą księgę dotyczącą sędziów pokoju, jak również przewodniczył zespołowi. Dziękuję serdecznie.

Proszę bardzo, pani poseł.

Nie podoba nam się on, bo nie podoba nam się, że minister sprawiedliwości rządzi prokuratorami. Nie podoba nam się, że stale wydłużają się postępowania sądowe i zbyt długo trzeba czekać na orzeczenia. Nie podoba nam się to, że nie wybieracie sędziów na wolne stanowiska sędziowskie. Nie podoba nam się to, że mimo postulatów pracowników administracyjnych, kuratorów nie podnosicie im wynagrodzeń, by stały się godziwie. Nam się taki wymiar sprawiedliwości, jak wy tworzycie (Dzwonek), nie podoba. Dziękuję serdecznie. Teraz pan poseł Sachajko powie, co mu się nie podoba. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Właśnie słuchałem i państwa wniosek o odrzucenie projektu prezydenckiego w pierwszym czytaniu pokazuje, że państwo jednoznacznie nie chcą żadnych zmian. No dobrze. Proszę państwa, wysłuchaliśmy.

Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Bardzo proszę. Można wszystko, tylko czasami uśmiech też by się przydał. Wysoka Izbo! Chodzi o zmiany, które kierunkują pewne myślenie zgoła inne, niż do tej pory, przez ostatnie lata towarzyszyło politykom. Chodzi o przejmowanie pewnej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez różne środowiska, przekazanie tej kontroli w większym stopniu obywatelom.

Jak słucham o kosztach wyborów bezpośrednich powiązanych z tymi procedowanymi ustawami, to trochę mnie to bawi, ponieważ jakbyście państwo policzyli, ile Polska płaciła w wyniku wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za skargi obywateli polskich na wymiar sprawiedliwości, to okazałoby się, że ta kwota jest zdecydowanie większa w ostatnich latach. Ubolewam tylko, że w tej dyskusji nie ma Ministerstwa Sprawiedliwości, bo przecież to Ministerstwo Sprawiedliwości powinno mieć tutaj głos opiniotwórczy i pokazać elementy, z którymi się zgadza lub się nie zgadza. Oczywiście jak najbardziej będziemy chętni do rozmów nad wszystkimi państwa projektami. One są trochę różne i dotykają różnych spraw, niemniej jednak powinniśmy dyskutować, np. nad sposobem wyboru. Oczywiście najbliżej Polskim Sprawom jest do projektu prezydenckiego i projektu Koalicji Polskiej, być może nawet bardziej do Koalicji Polskiej, ponieważ tam są te elementy pierwotne i zasadnicze, które idą najdalej, jeśli chodzi o demokratyzację. Boicie się państwo wyborów powszechnych, boicie się demokracji bezpośredniej. Skupmy się na tym, jak ludzi edukować, żeby to nie były kampanie plakatowe. Jak edukować, jak dostarczać ludziom wiedzę, żeby ich wybory były świadome, żeby dokonywali wyborów sędziów pod względem kwalifikacji, zaufania społecznego. Ludzie muszą się nauczyć, komu ufają, i dopiero później mogą weryfikować.

Już nie mówię o bardzo długim doświadczeniu, ale z całą pewnością sprawy, którymi będzie zajmował się sędzia, te drobne sprawy, ale tak naprawdę bardzo życiowe. Tymi sprawami musi zajmować się sędzia, który nie tylko czyta literę prawa, ale też zna życie, zna społeczność lokalną i potrafi w całą doktrynę swojego orzekania włożyć również empatię czy znajomość sytuacji życiowych. Oczywiście ważne jest, abyśmy podjęli dyskusję na temat sposobu wyboru, żeby było poczucie, że nie tylko i wyłącznie Krajowa Rada Sądownictwa poprzez różne kompetencje ma wpływ na to, kto ostatecznie zostanie sędzią pokoju, ale przede wszystkim żeby ludzie mieli poczucie, że oddali swój głos na kogoś, kogo znają lokalnie i wiedzą, że ta osoba tak naprawdę ma szansę, że żaden polityk w tym nie będzie uczestniczył. Ja się bardzo cieszę, że ta dyskusja się odbywa. Ona jest absolutnie potrzebna. Wymiar sprawiedliwości nie jest lepszy, chociaż wszyscy już teraz dokładnie widzą, że zmiany personalne z naszych na waszych, z waszych na naszych, których będziemy kontrolować, po prostu absolutnie nie działają. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia debata i że będzie ona rzeczowa. Ważne, że rozmawiamy, że będziemy przytaczać argumenty i że ludzie będą słuchać, czego tak naprawdę ta instytucja sędziów pokoju będzie dotyczyła, bo to jest element edukacji, do której my wszyscy jesteśmy zobowiązani jako politycy. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Proszę państwa, przechodzimy do zadawania pytań.

Zapraszam pana posła Janusza Kowalskiego. Proszę państwa, znacie moje liberalne podejście do tych spraw. Proszę pani, siedzę tutaj od 2 lat, znam te zapewnienia.

Jak wyjdę, to się ruszę, oczywiście. Panie Marszałku! Uzupełniając niewiedzę posłów Platformy Obywatelskiej i Lewicy, chcę jasno podkreślić, że za reformę sądownictwa od 4 lat odpowiada bezpośrednio pan prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, po zatrzymaniu reformy pana ministra Zbigniewa Ziobro w 2017 r. z polskiej strony z dobrymi chęciami, zakończył się niestety porażką, bo po stronie Brukseli tej dobrej chęci nie było i nigdy nie będzie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dzisiaj największy problem sądownictwa. Tym problemem jest oczywiście gangrena. Tą martwą tkanką w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sądownictwo, są upolitycznieni sędziowie, którzy chodzą na te wszystkie KOD-owskie urodziny z Donaldem Tuskiem, klaskają. Zamiast orzekać w sądach, bawią się w politykę (Dzwonek), chodzą na ustawki Platformy Obywatelskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie ministrze, z całą sympatią dla pana, przybył pan do Pałacu Prezydenckiego w todze z zielonym żabotem, ale niestety dziś zgubił pan po drodze ten etos prawniczy, bo przygotował pan absolutny bubel prawny. Prosty przykład: w ustawie o sądach powszechnych jest napisane, że sędzia urzęduje w todze z łańcuchem i orłem w koronie, a w pana ustawie jest napisane, że sędzia pokoju będzie urzędował w todze z łańcuchem z orłem, ale już bez korony, gdzieś pan zgubił koronę po drodze. W art. 18 jest napisane, że nie może być kandydatem na sędziego pokoju każda osoba, przeciwko której toczy się postępowanie. A co z domniemaniem niewinności? Możecie wytaczać te postępowania tylko po to, żeby zamknąć ścieżkę dostępu do tej funkcji. Więc tak naprawdę to jest ustawa o ścieżce kariery z awansu społecznego dla działaczy PiS. Jest wiele większych problemów, chociażby w kwestii alimentów. Sugerowanie, że to są proste sprawy i dawanie możliwości ministrowi sprawiedliwości ściągania tajemnicy w tej sprawie z sędziów pokoju (Dzwonek) jest kolejnym absurdem, który w tej ustawie nie może mieć miejsca. Takich problemów jest znacznie więcej. Sam wybór sędziów nie jest bezpośredni, panie marszałku, jest pośredni. Pan poseł Jan Szopiński, Klub Parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiemy już, że prezesami sądów pokoju będą prezesi sądów rejonowych, a wszystkimi aspektami ich działalności będzie rządził minister sprawiedliwości. Sprawy mają być przyznawane losowo, ale na przydział ma wpływ minister, dbając o proporcjonalność obciążenia sprawami. Zatem reasumując, ma być tak jak pewnie z reasumpcjami w naszym Sejmie do czasu osiągnięcia pożądanego wyniku głosowania, a tam losowania mogą być powtarzane. Wiemy też, kto może zostać sędzią pokoju - może być nim każdy niekarany magister prawa. Czy to dobre i jedyne kryteria, by dobrze sprawować urzędy sędziów pokoju, Polacy muszą odpowiedzieć sobie sami. Tymczasem ja uprzejmie proszę kancelarię pana prezydenta o uzasadnienie tych wymagań, które muszą wypełniać sędziowie pokoju. Uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Na początek pytanie do nieobecnego pana ministra sprawiedliwości, co sądzi o instytucji sędziów pokoju i czy w kontekście planowanej reformy spłaszczenia struktury sądów w Polsce w ogóle dopuszcza taką myśl. Pytanie do pana ministra reprezentującego pana prezydenta: Czy odbyły się jakiekolwiek rozmowy na linii Pałac Prezydencki - Ministerstwo Sprawiedliwości?

Jeśli chodzi o odpowiedź ministra Ziobro, ministra sprawiedliwości, bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Artur Dziambor, koło parlamentarne o nazwie Konfederacja. Wysoka Izbo! Na temat sędziów handlowych chciałem powiedzieć, że jest to rozwiązanie, które oczywiście jest od bardzo dawna oczekiwane przez środowisko, i jest to rozwiązanie jak najbardziej pozytywne, idące w bardzo dobrą stronę. Natomiast chciałem powiedzieć, że przede wszystkim wszelkie kroki, które mają usprawnić jakkolwiek działalność sądów - i to w tym przypadku akurat we wsparciu ze strony specjalistów - są pozytywne i należy je popierać.

Innymi słowy, o ile wzrośnie nam koszt utrzymania całego systemu i ile tacy sędziowie będą zarabiali za prowadzenie sprawy? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście obywatele nie mają żadnych wątpliwości, że dotychczasowe zmiany wprowadzane przez rząd PiS w obszarze sądownictwa spowodowały, że ono działa chyba najgorzej, przynajmniej od 1989 r. Coraz dłuższy czas oczekiwania, coraz mniejsze zaufanie, odpływ doświadczonych pracowników to skutek działalności zarówno rządu, jak i pana prezydenta.

Te projekty wychodzą naprzeciw oczekiwaniu takiego prostego rozwiązania sprawy. To pytanie do pana ministra, który jest przedstawicielem Kancelarii Prezydenta. Nowo powołani sędziowie zgodnie z projektem mają być weryfikowani przez upolitycznioną KRS, a później powoływani przez pana prezydenta. W jaki sposób pan prezydent to tłumaczy ludziom? Przecież oni powinni wybierać, a nie KRS. Dziękuję bardzo. Pierwsze dotyczy propozycji, którą złożyłem w trakcie omawiania projektów, aby powiązać wybory na sędziów pokoju z wyborami prezydenckimi. Wtedy mielibyśmy zapewnione to, że one będą rzeczywiście powszechne.

Taki sędzia nie będzie miał motywacji do tego, żeby rzeczywiście pracować tak, jak powinien pracować. Jeżeli byłyby to dwie kadencje i po drugiej kadencji on od razu mógłby być wybrany przez KRS do sądu, to wtedy widzimy jego zaangażowanie i nie ma tego niebezpieczeństwa, że to będzie tylko taki element w karierze prawnika. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Kazimierz Smoliński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szkoda, że dyskusja nad tak ważnymi i przełomowymi projektami w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości w pewnych momentach niestety była kompletnie niemerytoryczna.

Gdyby iść tym torem, to za chwilę powiemy, że Sejm jest upolityczniony. Mam pytanie do pana. Widzę, że posłowie nie rozumieją takich podstawowych sarkastycznych sformułowań, ale trudno, mogę to tłumaczyć.

Dobrze, wszystko na spokojnie. Bardzo proszę. Proszę zadać pytanie. Panie Ministrze! Mam pytania związane z projektem.

Czy kwestia pewnych wpłat czy braku ograniczenia przez jedną osobę wpłat nie może spowodować, że jedna osoba może sfinansować całą kampanię wyborczą? Tych pytań jest więcej. Czy w kwestii kadencji jest tutaj otwartość ze strony pana prezydenta na ewentualne zmiany w dalszym procedowaniu? Bardzo bym o to apelował. Tak jak mówię, popieramy wszystkie projekty, one powinny być przedmiotem obrad, ale bardzo proszę do nich podchodzić rzetelnie i obiektywnie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Odniosę się merytorycznie do projektów ustaw o sędziach pokoju. Chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na negatywne skutki tej regulacji. Mówię tu o stanie zamieszania prawnego i niepewności prawnej w zakresie spraw sądowych i zapadłych czy mających zapaść orzeczeniach wywołanych rewolucyjnymi zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ciągle istniejąca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - dla niektórych tylko na papierze - mówi wyraźnie, że wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe. Trudno w tym przepisie konstytucji doszukać się instytucji sądu pokoju. To oznacza, że każdy wyrok takiego sądu może być uznany za akt władzy państwowej, ale nie tej uprawnionej do wydania wyroku, tej wskazanej w ustawie zasadniczej mającej (Dzwonek) najwyższą moc prawną. Jak zatem ten przepis konstytucji pogodzić z celem wskazanym w uzasadnieniu projektu, którym ma być wzmocnienie sądownictwa, tak aby obywatele utożsamiali się z polskim wymiarem sprawiedliwości i mieli zaufanie do sędziów? Pani posłanka Karolina Pawliczak, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sędziowie pokoju, sprawiedliwość blisko ludzi - tak brzmi hasło na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sędziów pokoju. Ale wątpliwości jest bardzo wiele. Projekt ustawy zakłada bowiem, że na stanowisko nie mogą kandydować adwokaci, radcowie prawni czy aplikanci. Będą musieli zrezygnować z tych funkcji lub je po prostu zawiesić. Ale zakaz nie obejmuje prokuratorów w stanie spoczynku. Czy to oznacza, że PiS otwiera furtkę do obsadzania tych stanowisk przez prokuratorów Ziobry? Kandydaci będą zgłaszani do upolitycznionej KRS, która będzie sprawdzać, czy spełniają oni wymogi, co pozwoli na utrącanie niewygodnych dla władzy kandydatów. No i wreszcie co z zapisami konstytucji? Czy nie jest tak, że bez zmiany konstytucji nie można wprowadzać takiej instytucji? Zgodnie z art. 177 bowiem sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości (Dzwonek), a inne formy można stosować w ramach procedury przedsądowej. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska. Proszę, Jacku. Panie Marszałku! Panowie Posłowie!

Czy ocenia pozytywnie swoją decyzję, czy wręcz negatywnie?

Po drugie, jak pan prezydent ocenia aktualne propozycje, zapowiedzi reformy wymiaru sprawiedliwości, nad którymi pracuje się w Ministerstwie Sprawiedliwości, w kontekście również sędziów pokoju?

Poprosimy teraz pana posła Mariusza Goska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jest pan poseł? Nie ma. To poprosimy panią poseł Henrykę Krzywonos-Strycharską, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W sprawach o wykroczenie z powodu kierowania wniosków do sądu o ukaranie uczestników demonstracji, które zazwyczaj odnosiły się do obrony praw kobiet, niezawisłości sądów, obrony demokracji i wielu innych kwestii, dość często sędziowie, wydając wyrok, powoływali się na konstytucję i prawo międzynarodowe i uniewinniali te osoby. W związku z powyższym mam pytanie: Czy uważacie państwo, że sędziowie pokoju będą umieli zagłębić się w sprawy oraz konstytucję i prawo międzynarodowe, aby wydać sprawiedliwy wyrok? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Zdzisław Wolski, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo!

Najważniejszym zapewne warunkiem jest właściwy wybór sędziów pokoju - kompetentnych, merytorycznych i niezależnych. Mam pytanie do pana prezydenta.

Pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powołanie instytucji sędziów pokoju tak naprawdę odciąży w pierwszej kolejności sądy okręgowe, do których nie trafią te sprawy, które do tej pory w wyniku odwołania z sądów rejonowych trafiały. Otóż te sprawy zakończą się w sądzie rejonowym w pierwszej instancji, jeśli dobrze zrozumiałem projekt. Chodzi mi o środki odwoławcze, które przysługują normalnie, zwłaszcza te środki, które są środkami nadzwyczajnymi. Czy tutaj zachodzi jakaś istotna zmiana? To pierwsze pytanie.

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Nie ma posła Łąckiego. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Pani poseł Barbara Dolniak, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do przedstawiciela prezydenta. Dużo słyszeliśmy o konsultacjach. Chciałam zapytać, jakie konsultacje były prowadzone w związku z opracowanymi projektami. Jak szerokie były te konsultacje, czy w tym samym stylu, jak w przypadku projektów dotyczących KRS-u czy Sądu Najwyższego? A gdzie analiza skutków tych projektów?

Jak długo trwały i z kim były prowadzone? A gdzie analiza? Poza krótkimi, okrągłymi zdaniami, że były prowadzone konsultacje, nie ma żadnej analizy, są tylko i wyłącznie okrągłe zdania w tym uzasadnieniu. Jak to jest możliwe, że kandydować na sędziego pokoju może osoba, która należy do partii politycznej? Przecież to jest wprost wciąganie partii politycznych w proces kandydowania. Jak to jest możliwe? A co z kadencyjnością? Przecież wyraźnie mowa jest w konstytucji, że nie ma kadencyjności. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jedynym dorobkiem prezydenta Dudy i tego rządu, PiS-owskiego rządu, jest wydłużenie czasu postępowań sądowych z 4 do 7 miesięcy.

Szanowni państwo, chciałbym zapytać, pod kogo kroiliście tę ustawę. Doświadczenie, jakiego wymagacie od kandydatów na sędziów pokoju, to doświadczenie w zakresie czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa. Czy te kryteria były pisane pod asystentów i współpracowników Łukasza Mejzy? Bo idealnie się wpisują właśnie w wymagania wobec pracowników biur poselskich, radnych i innych politycznych kacyków, których macie pod dostatkiem.

Pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po 6 latach waszych rządów wciąż próbujecie tych samych sztuczek w niszczeniu wymiaru sprawiedliwości. Reforma Trybunału Konstytucyjnego miała usprawnić procedowanie. Efekt: TK rozpatruje mniej spraw niż przed zmianą, ale za to orzeka tak, jak tylko sobie PiS zażyczy. Zmiany w sądach powszechnych miały przyspieszyć pracę sądów, tymczasem spowodowały spowolnienie, a sędziowie są prześladowani i zastraszani. Dlatego kiedy przedkładacie kolejny projekt i uzasadniacie go usprawnieniem, to wiemy, że chodzi wam o chaos i dalsze podporządkowywanie sobie sądów. Dziś niezależni sędziowie uniewinniają obywateli protestujących przeciwko władzy. Czy sędziowie pokoju będą robić to samo, powołując się konstytucję? Nie sądzę. Ten projekt jest wam potrzebny tylko po to, żeby dobić politycznego targu z Pawłem Kukizem i utrzymać większość w Sejmie. Ostatnie zdanie, panie marszałku. Święte prawo obywateli i obywatelek do niezawisłego sądu sprzedajecie za utrzymanie się przy władzy. Nie ma i nie będzie na to zgody. Dziękuję. Pan poseł Dariusz Joński, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Halo, panie pośle, mam do pana uprzejmą prośbę. Akurat pana posła Jońskiego znam bardzo długo i nie chciałbym, żeby się stresował przez was. Dziękuję, panie marszałku. Pana marszałka też znam długo, więc też nie chciałbym, żeby pan marszałek się stresował tym, że ktoś rozmawia na sali. Co do projektu ustawy, fundamentalna, najważniejsza uwaga jest taka, że my mamy system sprawiedliwości zapisany w konstytucji i jakakolwiek zmiana wymaga również zmiany konstytucji. Dziwię się, że robi to pan prezydent, chociaż może już nie powinienem się dziwić. Ale trudno się nie zgodzić z prof. Ćwiąkalskim i prof. Zollem, byłym prezesem trybunału i byłym rzecznikiem praw obywatelskich, którzy podkreślają właśnie, że nie można uchwalić tej ustawy bez zmiany konstytucji.

Przez 10 lat będzie to prawie 9 mld zł.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Sędzia pokoju. Usłyszałam tutaj, że ludzi trzeba nauczyć zaufania. Przez 6 lat jesteśmy okłamywani, oszukiwani, manipulowani, przekupywani datkami. Nie da się, proszę państwa, szybko naprawić tej sytuacji. Sędzia pokoju sprawdziłby się na pewno w warunkach pełnej demokracji i samorządności, czego u nas niestety brakuje. Po 6 latach reformy sądownictwa nasze sądy są bezradne, spowolnione i upartyjnione, wszystko na korzyść cara Ziobry. Ponadto jest to wywiązanie się z umowy, handel z panem Kukizem za poparcie i głosy, bo prawdopodobnie nigdy nie zgodzilibyście się na taki absurd. Kolejna niewiadoma. Obecny stan naszego sądownictwa potrzebuje wsparcia, ale działań sprawdzonych, a nie kolejnej innowacji. Czy jednym z kryteriów wyboru sędziego będzie wspieranie PiS? Czy będzie to gwarancją niezawisłości? Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, przechodzimy do podsumowywania naszej dyskusji, pytań i stwierdzeń.

9. Bardzo proszę, pani minister. Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za udzielenie głosu, bo usłyszałam, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest obecne podczas dzisiejszej debaty. Jest obecne. Wsłuchiwało się we wszystkie argumenty i we wszystkie stanowiska i głosy w dyskusji. Dzisiaj debatujemy nad pięcioma projektami ustaw. Jak słusznie zauważyła pani poseł Anna Żukowska, to nie jest wyścig. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany ustrojowe, one muszą być przemyślane i dogłębnie przeanalizowane. Odnośnie do przedstawionych przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektów ustaw: o sądach pokoju i Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju chcę zaznaczyć, że rząd jeszcze nie zajął stanowiska, ale w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto już prace analityczne, które niewątpliwie będą skutkować opracowaniem kompleksowych uwag do tego projektu. Nie ulega wątpliwości, że sam projekt należy ocenić jako zawierający warte refleksji i pochylenia się nad nim rozwiązania wymagające jednak bardzo wnikliwej analizy i przygotowania bardzo szczegółowego stanowiska, które zapewne będzie prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w toku dalszych prac legislacyjnych. Ale już wstępna analiza projektu pozwala na poczynienie przynajmniej kilku uwag wymagających bez wątpienia wyjaśnienia w toku dalszych prac. Generalnie w odniesieniu do proponowanego katalogu spraw karnych można wyrazić zapatrywanie, że z uwagi na ich charakter powinny one jednak zostać wyłączone spod jurysdykcji sądów pokoju. Jako jeden z argumentów przemawiających za tą tezą należy wskazać konsekwencje wprowadzenia ograniczeń jurysdykcyjnych dla sędziów w odniesieniu do wymierzanych przez nich kar, tj. kary grzywny, kary ograniczenia wolności, [[Oklaski]] która trwa najdłużej 6 miesięcy, kary pozbawienia wolności trwającej najdłużej 3 miesiące. Zgodnie z projektem sprawa podlega przekazaniu właściwemu sądowi, jeżeli w toku postępowania przed sądem pokoju okaże się, że na podstawie okoliczności sprawy, w tym ujawnionych na rozprawie, sąd pokoju przewiduje możliwość wymierzenia kary wyższej niż 3 miesiące pozbawienia wolności. Projekt przewiduje również, że sąd pokoju może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że rozstrzygnięcie sprawy ze względu na jej przedmiot, zawiły charakter wymaga jej rozpoznania przez sąd rejonowy. W chwili obecnej trudno prognozować, jak ukształtuje się praktyka w momencie wejścia w życie ustawy, ale niestety realne jest zagrożenie, że sądy pokoju mogą często korzystać z praktyki przekazywania tego typu spraw sądom rejonowym, chociażby jeżeli wziąć pod uwagę ten argument, o którym mówiłam, iż sąd pokoju będzie miał prawo jedynie wtedy wymierzyć karę pozbawienia wolności, jeśli uzna, że powinna być wymierzona w granicy 3 miesięcy. Obawiamy się, że może to doprowadzić do złagodzenia wymiaru kary, a na takie rażące złagodzenie Ministerstwo Sprawiedliwości absolutnie nie może się zgodzić. W toku dalszych prac pod rozwagę należy poddać mechanizm przekazywania sprawy do sądu rejonowego choćby w sytuacji, którą przewiduje projekt, gdy przed sądem pokoju zaistnieje konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Wówczas sprawa nie będzie podlegała rozpoznaniu przez sąd pokoju. Po pierwsze, projektowana w tym liczba wyłączeń spraw spod właściwości sądu pokoju oraz sposób sformułowania tych wyłączeń mogą ostatecznie prowadzić do wielokrotnego przekazywania pomiędzy sądami akt, co ostatecznie będzie skutkowało wydłużeniem postępowania, a rozumiem, bo to wybrzmiało w czasie dzisiejszej debaty, że przewlekłość postępowania leży nam wszystkim na sercu i chcemy, aby okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy był jak najkrótszy. Tak jak zaznaczyłam na wstępie, projekty pana prezydenta są analizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, są godne uwagi i na pewno będziemy merytorycznie brać udział w toku dalszych prac i odnosić się do poszczególnych rozwiązań.

Odnosząc się do poselskiego projektu ustawy o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 1378, chciałabym zaznaczyć, że projekt został negatywnie zaopiniowany przez rząd.

Przepisy nie mówią, kto miałby tę wiedzę weryfikować i w jaki sposób miałaby być ona kontrolowana. Projekt wprowadza cenzus wieku: 29 lat, ale nie wprowadza cenzusu wykształcenia. Projekt ustawy przewiduje, że obywatelscy sędziowie handlowi przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami, z tym że nie mogą przewodniczyć na rozprawie czy naradzie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą.

Rząd zatem w stosunku do przedmiotowego projektu zajmuje negatywne stanowisko, gdyż utworzenie instytucji obywatelskich sędziów handlowych stoi w sprzeczności z wymogami konstytucyjnymi dotyczącymi statusu sędziów.

W jaki sposób wzrosną koszty postępowań w sądowych sprawach gospodarczych, w jaki sposób ewentualnie ci sędziowie mieliby być opłacani - te rozwiązania nie znalazły się w uzasadnieniu. Jeśli chodzi o poselski projekt ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 1762, to po pierwsze, założenie konstrukcyjne prowadzące do wykreowania uprawnień jurysdykcyjnych nowej kategorii sędziów niezawodowych uzasadnia w pierwszym rzędzie potrzebę wypowiedzi co do zgodności tych uregulowań z przepisami konstytucji Rzeczypospolitej, jak również w zakresie możliwości powoływania takiego sędziego na czas określony. Bez zmiany konstytucji nie jest bowiem możliwe przeprowadzenie takich zmian ustawodawczych, aby były zrealizowane kierunki zaproponowane w tej ustawie. Projekt podzielono na pięć rozdziałów: Organizacja sądów, Właściwość sądów pokoju,

Odnosząc się do propozycji rozwiązań zawartych w tym projekcie, wskazać należy na podstawowe wątpliwości właśnie w zakresie oceny zgodności z konstytucją tych propozycji, które przede wszystkim dotyczą kadencyjności, powołania na stanowisko sędziego oraz motywów, gdyż projektodawca, nawiązując do potrzeby projektowania regulacji, uwagę poświęca wyłącznie konieczności zachowania trybu powołania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co odpowiadać ma dochowaniu wymagań - tak przynajmniej ocenia to projektodawca - o których mowa w art. 179 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Za co najmniej wątpliwą z punktu widzenia systemu aksjologicznego wyrażonego dotychczasowymi przepisami dotyczącym tego, w jaki sposób sędziowie dochodzą do swojego zawodu - obecnie dzieje się to przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - można uznać propozycję regulacji polegającą na tym, że w razie rezygnacji z ubiegania się o ponowny wybór w wyborach na sędziego pokoju jest możliwe przeniesienie takiej osoby z urzędu na stanowisko sędziego sądu rejonowego, przy którym orzekał jako sędzia pokoju. Za wątpliwy z punktu widzenia normy przejściowej, o której jest mowa w art. 237 konstytucji, trzeba ocenić zawarty w uzasadnieniu projektu passus mówiący, że projektowana ustawa ma być też swego rodzaju odpowiedzią ustawodawcy na dokonaną w 2001 r. na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego likwidację kolegiów do spraw wykroczeń i przekazanie rozpoznawanych przez nie spraw wydziałom karnym sądów rejonowych. Stanowisko w zakresie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju, druk nr 1763, również nie zostało na chwilę obecną zajęte przez rząd. Mogę zaprezentować tylko stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, co niniejszym czynię.

Tak naprawdę regulacje te odnoszą się do zmiany przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeksu postępowania cywilnego czy też Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy art. 4 do 5 przewidują obowiązek składania przez ministra sprawiedliwości informacji o działalności sądów pokoju, natomiast przepis art. 5 przewiduje, że ustawa wchodzi w życie na obszarze województwa opolskiego i kujawsko-pomorskiego po upływie roku od dnia ogłoszenia, a w pozostałych województwach ustawa wchodzi w życie po upływie 3 lat od dnia ogłoszenia. Z taką regulacją absolutnie nie sposób się zgodzić. Nie ma bowiem możliwości, aby na terenie kraju na danym obszarze obowiązywał inny ustrój niż na pozostałym obszarze kraju. Nie można wprowadzać pilotażu w zakresie zmian ustrojowych dotyczących funkcjonowania sądów. Ponadto, zgodnie z projektowanym w tym projekcie przepisem art. 61 § 2 pkt 6 ustawy o ustroju sądów powszechnych, sędzia pokoju, który zajmował stanowisko sędziego pokoju przez co najmniej dwie kadencje, ma zyskać możliwość zgłoszenia swojej kandydatury w konkursie na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego. Takie rozwiązanie ma stanowić wprowadzenie kolejnej przesłanki, która zwalnia zainteresowanego kandydata na sędziego sądu rejonowego z wymaganych, co do zasady, obowiązku złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego lub zajmowania stanowiska asesora sądowego pełniącego obowiązki sędziego co najmniej przez 3 lata. Odnosząc się do tych propozycji, wstępnie należy zasygnalizować ponownie kwestię kadencyjności sędziów pokoju, sprzeczności projektowanych regulacji dotyczących mechanizmu wyboru kandydatów na sędziów pokoju przez rady gmin i zgromadzenie ogólne sędziów sądów rejonowych, z pominięciem aktu inwestytury pochodzącej od pana prezydenta, brak ochrony immunitetowej w ramach immunitetu formalnego, negatywne konsekwencje w zakresie płaszczyzny procesowej, zwłaszcza w tym obszarze, o którym już mówiłam, co do okresu obowiązywania w dwóch okręgach sądowych tej ustawy przez, jak to nazywa projektodawca w uzasadnieniu, okres pilotażowy.

Będziemy się pochylać nad rozwiązaniami. Nie jest tak, że uchylamy się od tej pracy, a moje niezajmowanie wcześniej stanowiska w dzisiejszej dyskusji było wynikiem tylko i wyłącznie tego, że czekałam na to, aż taki głos zostanie mi udzielony przez pana marszałka. Pytanie, które odnotowałam, a które zostało skierowane do pana ministra sprawiedliwości, to było pytanie zadane przez pana posła Paszka. Dotyczyło sędziów pokoju i spłaszczenia struktury, ale pan poseł poprosił o odpowiedź na piśmie i taka odpowiedź zostanie panu posłowi udzielona. Dziękuję bardzo, pani minister. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana ministra Pawła Muchę. Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Bardzo dziękuję za głosy, które zostały wyrażone w ramach tej debaty, w ramach dyskusji, a w szczególności za głosy aprobaty, bo te głosy zdecydowanie przeważały, jeżeli chodzi o wystąpienia klubowe, jeżeli chodzi o wystąpienia posłów. To jest rozwiązanie, które daje szansę na walkę z dwoma głównymi bolączkami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jakimi są brak zaufania do sądów i kwestia związana z przewlekłością postępowania.

Przypomnę, że o sądach pokoju stanowiła m.in. konstytucja marcowa i że sądy pokoju działały w odrodzonej Rzeczypospolitej, były bardzo dobrze oceniane. Inną rzeczą jest to, że później w trakcie zmian ustrojowych, prawnych zostały one wyeliminowane, ale absolutnie nawiązujemy nie tylko do tradycji anglosaskich i do modeli, które są w systemie kontynentalnym, europejskim, ale także do polskich tradycji prawnych. Były argumenty konstytucyjne. Szanowni państwo, oczywiście o konstytucyjności rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny, ale jeżeli padają argumenty natury konstytucyjnej, to powiem tak. Art. 175 konstytucji stanowi: „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne” Bardzo wyraźnie w tych projektach stanowimy, że sądy pokoju są elementem sądownictwa powszechnego.

Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Art. 182 polskiej konstytucji stanowi: „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa” To są te ustawy, tj. ustawa o sądach pokoju i ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju.

To wynika wprost z piśmiennictwa, z głosów, które pojawiają się w debacie publicznej, z komentarzy do konstytucji, z publikacji, które były wydawane nawet w tym roku, jeżeli chodzi o te kwestie. Wreszcie kwestionujecie państwo udział w procesie, jeżeli chodzi o gwarancję niezawisłości sędziowskiej, KRS-u. To już jest rzecz absolutnie kuriozalna.

Dzisiaj w polskim systemie prawnym orzekają asesorzy, i to musi pani marszałek, pani poseł, pani sędzia wiedzieć, orzekają ławnicy, a my chcemy wzmocnić udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Nie bójcie się państwo demokracji, nie bójcie się wyborów powszechnych, nie bójcie się tego, że obywatele będą decydować o sprawach obywateli - profesjonalnie przygotowani, wybrani bezpośrednio w wyborach przez społeczność lokalną. To są dobre rozwiązania. Ja nie rozumiem tych obaw dotyczących braku zaufania do ludzi czy braku zaufania do społeczeństwa i bardzo dziękuję tym z państwa, którzy takich wątpliwości nie mają. Przykro mi, że z tego apelu wyłamały się członkinie klubu, które miały wystąpienia już nie tak spokojnie i nie tak merytoryczne.

Absolutnie bardzo dziękuję za podobne postrzeganie tych problemów.

Widzę, że spojrzenie na te sprawy czy identyfikowanie tych problemów, tak jak to pan poseł przedstawiał, jest wspólne dla Koalicji Polskiej i dla pana prezydenta.

Jestem więc optymistą, jeżeli chodzi o głosy tych dwóch ugrupowań opozycyjnych, że jesteśmy w stanie pracować i merytorycznie dyskutować nad tymi projektami, udoskonalając je w toku debaty parlamentarnej.

Myśmy wskazali jedną kadencję, natomiast po to jest praca w komisji, żeby dzielić się argumentami, szczegółowo się do tego odnosić i przekonywać, które rozwiązania są najtrafniejsze. Starałem się bardzo krótko powiedzieć o tym, że trudno tutaj wskazywać na jakiekolwiek podstawy jakiegokolwiek kwestionowania konstytucyjności tych rozwiązań. To znaczy apeluję, żeby głos przedstawiciela wnioskodawów pana posła Myrchy był uwzględniony także przez państwa i żebyśmy nie rozmawiali na zasadzie obelg czy krzyków, tylko żebyśmy rozmawiali o problemach wymiaru sprawiedliwości merytorycznie. Jeżeli chodzi o kwestię dalszych szczegółowych pytań, pojawiło się kilka pytań dotyczących kampanii. Jeżeli chodzi o projektowany art. 490t Kodeksu wyborczego - to jest w ramach przepisów wprowadzających - my wprost stanowimy, to jest § 1, cytuję: Kampania wyborcza kandydata na sędziego ogranicza się do prezentacji sylwetki kandydata, w tym przedstawienia informacji o jego wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz działalności społecznej, w trakcie zebrań organizowanych jako zadanie własne przez gminy. W wyborach sędziów pokoju zakazuje się agitacji wyborczej z wyjątkiem działań określonych w przepisach niniejszego rozdziału. To jest bardzo specyficzna kampania. Mówimy, że to ma być w istocie rzeczy prezentacja kandydata.

Nie będzie więc tutaj elementów związanych z kampanią polityczną, tak nie stanowi ten projekt. Inną rzeczą jest, że padały tutaj zarzuty, iż nie ma limitu.

Tak nie jest, a mówimy o porządkowaniu bardzo ważnego wymiaru, wymiaru sprawiedliwości, o sprawach kluczowych dla ludzi.

Jak doliczymy inne składniki, to średnie czy przeciętne wynagrodzenie z dodatkami wynosi 15 tys. Myślę, że to jest godziwe wynagrodzenie, mieszczące się w standardzie konstytucyjnym. To wynagrodzenie, które przewidzieliśmy dla sędziów pokoju, jest wynagrodzeniem na poziomie asesorów sądowych. Jest to zawarte w uzasadnieniu. Wydaje nam się, że ta liczba 3900 sędziów jest absolutnie adekwatna do tych potrzeb, o których mówimy. Bardzo dziękuję za wystąpienie pana posła Jarosława Sachajki, który bardzo wyraźnie mówił o demokracji i obywatelskości. Tak, to jest projekt obywatelski. Zresztą jest na sali pan przewodniczący Paweł Kukiz, który tę inicjatywę panu prezydentowi zgłaszał. Myślę, że każdy, kto jest za obywatelskością, ten projekt będzie popierał, bo on oddaje władzę ludziom.

To jest absolutnie zmiana, którą partia, która ma w nazwie słowo „obywatelska”, powinna popierać. Tak wskazywałaby przynajmniej logika.

Bardzo dziękuję za to dotychczasowe wsparcie merytoryczne i tę współpracę w ramach zespołu przedstawicielowi ministra sprawiedliwości, dziękuję za te rozmowy, które odbywamy jako Kancelaria Prezydenta RP z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jedna rzecz.

Nie będzie wielokrotnego przekazywania spraw. Muszę uściślić, że taka sytuacja na gruncie tego projektu jest niemożliwa. Natomiast absolutnie będziemy czekać na te wnikliwe analizy i kompleksowe uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości, tak jak mówiłem, także ze strony państwa posłów i klubów. Będziemy je rozstrzygać.

Stąd nasza decyzja, żeby skierować te sprawy wykroczeniowe, te sprawy drobniejsze bezpośrednio do sądów pokoju i w ten sposób odciążyć cały wymiar sprawiedliwości.

Absolutnie trzeba będzie w ramach przepisów przejściowych dostosować to do tej struktury, ale przypomnę, że to pan minister Zbigniew Ziobro w marcu tego roku, publicznie się wypowiadając, mówił, że jest za sądami pokoju, mówił o tym, jak ogromne nadzieje wiąże z tym projektem, więc nie sądzę, żeby jakakolwiek sprzeczność mogła tutaj występować. To są dobre propozycje, to są przemyślane propozycje, nad którymi chcemy pracować. Bardzo proszę o taką rzetelną, merytoryczną uwagę (Dzwonek), bo obywatele czekają, żeby te zmiany weszły w życie, żebyśmy przeszli od słów do czynów, żeby to się stało obowiązującym prawem.

To de facto jest pewnym potępieniem. Proszę przedstawiciela wnioskodawców pana posła Arkadiusza. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu w ramach sprostowania, ponieważ pan minister powiedział, że nasze wystąpienia jako przedstawicieli klubu Koalicji Obywatelskiej były tylko emocjonalne, a nie merytoryczne. Widać pan minister nie słuchał, bo powoływaliśmy się np. na art. 179 konstytucji, który absolutnie nie przewiduje kadencyjności w przypadku sędziów.

To nie są przykłady dyskusji merytorycznej? Mówiliśmy o tym, że kandydować na sędziego pokoju może osoba, która należy do partii politycznej, co jest niedopuszczalne w przypadku sędziów czy asesorów w sądach powszechnych, bo takiej możliwości nie ma.

Bardzo proszę pana posła Arkadiusza Myrchę o zajęcie stanowiska w imieniu wnioskodawców. Dziękuję, panie marszałku. Panie Ministrze Mucha!

Taką bezpośrednią emanacją art. 182 konstytucji jest instytucja ławników, którzy są właśnie społecznym uchem, społecznymi doradcami zawodowego sędziego.

Odnoszę się do wystąpienia pani podsekretarz z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W projekcie ustawy przyjęliśmy założenie analogiczne do rozwiązań, które dotyczą wynagradzania ławników, czyli jest system dzienny diet jako formy sprawowania funkcji społecznej. Oczywiście jest on procentowo ustalany od wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów.

Naszą intencją jest to, żeby obywatelscy sędziowie handlowi nie rezygnowali ze swojej aktywności zawodowej.

Ale żeby też nie nadwyrężać zbytnio budżetu wymiaru sprawiedliwości, jest ustalony limit spraw, w których sędziowie handlowi mieliby orzekać w toku kadencji.

Będziemy wiedzieli, jak duże jest zainteresowanie, w ilu postępowaniach faktycznie braliby udział, ale byłbym spokojny.

Art. 182 mówi jednoznacznie, że obywatele, ten czynnik społeczny, mają uczestniczyć w wymiarze sprawiedliwości, a nie go przejmować.

Uważamy, że rozwiązanie przygotowane, jak powiedziałem już wcześniej, w gronie ekspertów, wypływające ze środowisk, które są żywo tym rozwiązaniem zainteresowane, faktycznie usprawni w sposób realny postępowania gospodarcze, a co najważniejsze zwiększy zaufanie do wyroków, które zapadają w sprawach gospodarczych.

Sądownictwo musimy zmieniać w sposób odważny, jak powiedziałem, ale nie w sposób szalony. Bardzo dziękuję panu posłowi za przedstawienie stanowiska wnioskodawców. Głos zabierze kolejny przedstawiciel wnioskodawców pan poseł Krzysztof Paszyk. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Króciutko, ponieważ tylko w jednym wąskim zakresie czuję się wywołany do odpowiedzi przez uczestników debaty, jaka odbyła się m.in. nad projektem Koalicji Polskiej - PSL, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów, a mianowicie aspekcie konstytucyjnym wprowadzanych zmian dotyczących sądów pokoju i sędziów pokoju. Tworząc naszą regulację, opieraliśmy się na brzmieniu art. 175 ust. 1 konstytucji, który stanowi, że sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest zarezerwowane dla, po pierwsze, Sądu Najwyższego, po drugie, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Dlatego też zaproponowaliśmy, aby sądy pokoju stanowiły czwarty obok sądów rejonowych, sądów okręgowych i sądów apelacyjnych element sądownictwa powszechnego usytuowany w niniejszej hierarchii przewidzianej przez konstytucję Rzeczypospolitej. A więc nie uważamy, aby tu był możliwy zarzut, by istniała jakakolwiek kolizja z brzmieniem konstytucji, a idąc dalej za głosami niektórych uczestników tej debaty - aby istniała konieczność zmiany konstytucji poprzedzającej ustanowienie sądów pokoju i sędziów pokoju.

Tak jak wspomniałem, nasz projekt powstał - i tu chylę czoło przed marszałkiem Piotrem Zgorzelskim - w toku długich, wyczerpujących konsultacji z udziałem różnych środowisk, stowarzyszeń reprezentujących także tych, którzy zostali dotknięci przez wymiar sprawiedliwości funkcjonujący w dzisiejszym stanie rzeczy.

Dziękuję bardzo. Czy jest na sali przedstawicielka wnioskodawców pani posłanka Anna Maria Żukowska?

Panie Marszałku!

Wiadomo, że sprawy, które są zastrzeżone do rozpatrywania przez określone sądy, nie będą mogły być rozpatrywane przez sędziów pokoju. Już o tym mówiłam. Zastrzeżenia zgłaszały też reprezentantki Koalicji Obywatelskiej.

Tutaj też pojawia się termin „sędzia”, a jak wiemy, ten sędzia handlowy nie byłby sędzią w rozumieniu konstytucyjnym.

Ta dwuinstancyjność w projekcie Lewicy jest jak najbardziej zachowana, ponieważ można zaskarżyć orzeczenie sędziego pokoju. Jako sąd I instancji orzekałby wówczas sąd rejonowy, więc ta dwuinstancyjność byłaby jak najbardziej zachowana.

Tak samo wyglądałoby to w ujęciu naszego projektu, jeżeliby został wniesiony sprzeciw. Pojawiła się kwestia kosztów wprowadzenia tych projektów. Nasze rozwiązanie, rozwiązanie proponowane przez Lewicę, jest w tym wymiarze, myślę, najbardziej oszczędne. Po pierwsze, byłyby to wydatki ze strony budżetu państwa, z części budżetowej: Sądy powszechne. To jest oczywiste. Jak mówiłam, ten sąd pokoju nie funkcjonowałby jako jakaś odrębna instytucja. On jak najbardziej funkcjonowałby w ramach sądu rejonowego.

Tylko tak dla zobrazowania skali tych wydatków przypomnę tzw. wybory kopertowe, które nie doszły do skutku. 300 mln zł rocznie to jest dużo. To znaczy według projektu pana prezydenta miałoby być ich dużo więcej niż według naszego.

Można tę część wymiaru sprawiedliwości powierzyć właśnie obywatelom, przedstawicielom obywateli, w trybie wyboru. To jest już dla nas kwestia kontrowersyjna, jeżeli chodzi o propozycję prezydencką, te wybory powszechne.

Oczywiście nie ukrywam, że naszym zdaniem najbardziej konstytucyjnym, niebudzącym kontrowersji projektem jest projekt klubu koalicyjnego Lewicy.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował poselskie projekty ustaw: o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 1378, o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 1762, o sądach pokoju, zawarty w drukach nr 1763 i 1763-A, do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów ustaw zawartych w drukach nr 1760 i 1761. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1795) Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Jana Sarnowskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Wysoka Izbo! Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zawiera rozwiązania, których głównym celem jest wdrożenie trzech dyrektyw unijnych dotyczących podatku akcyzowego, to jest dyrektywy horyzontalnej, dyrektywy alkoholowej i dyrektywy obronnej. Najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie to jest przede wszystkim elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, objęcie ich monitorowaniem za pomocą systemu EMCS. To jest ważna zmiana o charakterze uszczelniającym i usprawniającym obrót towarami akcyzowymi. Bardzo ważną zmianą, oczekiwaną przez rynek i wielokrotnie postulowaną przez przedsiębiorców, jest wreszcie wprowadzenie w Polsce preferencji podatkowej dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. Polega ona na obniżeniu do 50%, czyli o połowę, podstawowej stawki akcyzy, a także dodaniu do ustawy definicji małego, niezależnego producenta i wprowadzeniu systemu certyfikowania, który umożliwi korzystanie z tej preferencji. Obecnie taka preferencja dotyczy jedynie piwa. Zmiany te ułatwią prowadzenie działalności i rozwój przedsiębiorczości małych, lokalnych producentów napojów alkoholowych, w tym firm rodzinnych. Dzięki temu będziemy wspierać mały biznes i produkty made in Poland, na czym skorzystają polscy rolnicy i sadownicy, przede wszystkim producenci win, miodów pitnych oraz wódek regionalnych. To jest bardzo ważna informacja dla ponad 150 polskich winnic, dla kilkunastu producentów cydru, perry i miodu pitnego, ale również dla 62 tys. polskich sadowników, którzy mogą być zainteresowani przetwarzaniem swoich owoców w dobre polskie wyroby regionalne. Inne zmiany zawarte w proponowanej, przedłożonej ustawie to m.in. uelastycznienie sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą w innym kraju, a przeznaczonych dla konsumenta. W takim przypadku również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć akcyzę na terytorium kraju, bez konieczności korzystania z pośrednika. Ustawa zawiera też uproszczenia w zakresie zabezpieczeń akcyzowych. Dopuszczone zostanie np. wykorzystanie jednego zabezpieczenia zbiorczo na potrzeby całości działalności podmiotu posiadającego różne statusy akcyzowe. Wejście w życie tych rozwiązań, z uwagi na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wdrożenie całego szeregu uproszczeń, ale również obniżek podatków, a także tych nowych rozwiązań elektronizujących, będzie przynosić pozytywne skutki dla budżetu państwa, ale przede wszystkim właśnie dla przedsiębiorców. Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. O przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę panią poseł Ewę Szymańską. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedstawiony przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt zawiera przepisy wdrażające kilka dyrektyw, m.in. dyrektywy Rady Unii Europejskiej z 2017 r., z 2019 r., jak również z 2008 r., a także dwie dyrektywy z 2020 r.

Kodeks karny skarbowy, ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Trzy z wymienionych dyrektyw winny być zaimplementowane do naszego prawa do 31 grudnia tego roku, a jedna z nich - do 30 czerwca przyszłego roku. Przedłożony projekt ustawy przewiduje m.in. następujące zmiany: w ustawie o podatku akcyzowym przesunięcie terminu całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji do 1 stycznia 2023 r., doprecyzowanie w zakresie składania kwartalnych deklaracji dotyczących wyrobów zwolnionych z akcyzy i ze stawką zerową, przesunięcie terminu przyznania nowych kompetencji Inspekcji Handlowej, co ma związek z planowanymi przez Komisję Europejską zmianami, a także warunki zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych stanowiących deputat węglowy, zmiany stawek akcyzy na oleje opałowe, węgiel, koks, gaz ziemny i pozostałe paliwa gazowe opałowe. Proponowane zmiany w podatku akcyzowym dotyczą również pomiaru Plato w piwie, aktualizacji kodów na wina musujące i napoje musujące, certyfikacji małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych, doprecyzowania zwolnień z akcyzy skażonego alkoholu używanego do produkcji lekarstw, a także, jak już tu wspomniał pan minister, obniżenie o 50% akcyzy na niektóre napoje alkoholowe. Przewiduje się również zwolnienie z akcyzy wyrobów akcyzowych, które mają być wykorzystywane przez siły zbrojne państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji zadań Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zmiany w ustawie o VAT realizują również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący tzw. szybkiego VAT, dostosowując przepisy do prawa unijnego. Uogólniając, proponowane przepisy dostosowują krajowe prawo do prawa Unii Europejskiej, precyzują je i upraszczają, a także wprowadzają zmiany ułatwiające pracę i działalność zarówno podatnikom, jak i organom stosującym przepisy i kontrolującym ich stosowanie.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Marchewkę, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ten projekt ma na celu implementację i wprowadzenie do prawa krajowego prawa, które zostało zatwierdzone na szczeblu państw Unii Europejskiej. Chciałbym zwrócić natomiast uwagę na kilka zasadniczych kwestii, które z tego projektu wynikają. Pierwsza sprawa jest taka, że w ramach tego projektu wprowadzane są pewnego rodzaju preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. Na tych właśnie zaproponowanych zmianach mogą skorzystać zarówno rolnicy, jak i sadownicy. A te właśnie przepisy, przepisy ułatwiające, polegają na obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy. Ważne jest także to, że w tym projekcie dodawane są przepisy, które jasno definiują małego, niezależnego producenta i wprowadzają specjalnie dedykowany dla tej grupy przedsiębiorców system certyfikowania.

Sprawa druga jest taka, że obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terenie Unii Europejskiej, czyli tych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Ten dokument ma formę papierową.

Po trzecie, w projekcie zostały również uwzględnione rozwiązania, których celem jest przede wszystkim uelastycznienie sprzedaży wyrobów akcyzowych na odległość. Dzięki właśnie tym rozwiązaniom również sprzedawca, który wysyła wyroby z innego państwa członkowskiego, będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju, co może stanowić dla niego po prostu proceduralne ułatwienie. Jednak, abstrahując od przepisów, które zostały tutaj zawarte, i odnosząc się do akcyzy i do podatków, które państwo nakłada na obywateli, chcę zwrócić uwagę na pewną kwestię. Bardzo wiele ostatnio rząd opowiada o tym, jak to chce obniżać akcyzę - mówi się o energii elektrycznej, mówi się o paliwach - natomiast chcę zwrócić uwagę, że również w tej ustawie czy w tym projekcie wskazano na pewien ważny cel, czyli dostosowanie obowiązujących stawek akcyzy, oczywiście na niektóre wyroby energetyczne, do kursu euro, który w stosunku do polskiego złotego wzrasta, czyli do poziomu 4,58, gdyż trzeba zachować odpowiednie poziomy unijne. W związku z tym zostanie wprowadzona zmiana stawek na niektóre wyroby.

Oczywiście z potrzeby dostosowania do kursu euro, ale trzeba też powiedzieć jasno, że to wynika z deprecjacji złotego, który jest coraz słabszy w stosunku do euro. Jednym z powodów były po prostu celowe interwencje na rynku walutowym, które podejmował Narodowy Bank Polski, w celu obniżenia wartości złotego. Dzisiaj niestety konsumenci za to zapłacą, bo te stawki będą po prostu wyższe. Co więcej, panie ministrze - to jest też uwaga do rządu - ostatnio podnieśliście akcyzę na alkohol i papierosy, i to w momencie trudnym dla polskiej gospodarki.

A więc ta najwyższa inflacja za ostatni miesiąc wynosząca już prawie 8% (Dzwonek) i te ogromne wzrosty kosztów energii elektrycznej to oczywiście duże obciążenia, które muszą ponieść polscy przedsiębiorcy. Panie marszałku, już kończę - pozwoli pan, jeszcze dwa zdania dosłownie. A więc według tych wyliczeń resortu akcyza, zgodnie z waszymi założeniami, ma przynieść do budżetu w nowym roku dodatkowe 2 mld zł.

Myślę - nie wiem, czy rząd zwraca na to uwagę, ale uważam, że powinien - że właśnie wzrost cen na alkohole może być pewnego rodzaju prezentem dla grup przestępczych, które są zainteresowane powiększaniem swoich zysków z pominięciem zobowiązań podatkowych, które powinny być płacone na rzecz państwa. A więc legalna sprzedaż może się po prostu skurczyć, co z kolei może zagrozić wielu firmom, ale także rolnictwu.

Natomiast jesteśmy za tym, żeby ten projekt implementujący przepisy unijne trafił do drugiego czytania w ramach podkomisji, która będzie się nim zajmowała, i będziemy dalej nad nim procedować. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Marka Rutkę, który przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedłożony projekt jest kolejnym przykładem na to, że obecna władza bardzo często traktuje Wysoką Izbę jak maszynkę do głosowania, a nie miejsce rzetelnej legislacji, w którym powstaje prawo, do którego obywatel ma zaufanie i przekonanie. Mimo że Rada Ministrów przyjęła przedmiotowy projekt noweli akcyzowej już 23 listopada, to dopiero 29 listopada projekt dotarł do Sejmu i w ekspresowym tempie, jeszcze tego samego dnia został skierowany do pierwszego czytania. Warto dodać, że nie jest to jakiś skromny dokument, a liczący 53 strony akt prawny z 82-stronicowym uzasadnieniem. Myślą przewodnią projektu noweli akcyzowej było i jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. Proponowane zmiany wywołane są także tym, że z dniem 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej. Ze względu na zmianę przepisów nowej akcyzowej dyrektywy horyzontalnej ma nastąpić elektronizacja obecnie papierowych uproszczonych dokumentów towarzyszących. Nie do końca jednak wiadomo, co jest powodem, dla którego polskie eUDT-y w projekcie nowelizacji akcyzowej z angielskiego nazwane są e-SAD-ami, ale być może to efekt pośpiechu, do którego w Wysokiej Izbie już nas przyzwyczajono. Oczywiście podkreślić należy, że nowy model nabyć wewnątrzwspólnotowych niesie dużo dalej idące zmiany w modelu postępowania niż tylko ww. elektronizacja dokumentów towarzyszących. Jako zmianę na plus przyjąć należy, że dzięki przepisom komentowanej noweli akcyzowej przedsiębiorcy będą mogli w końcu, choć po spełnieniu szczególnych warunków, importować wyroby akcyzowe wprost do składu podatkowego. Nowe przepisy ułatwiają również handel wyrobami akcyzowymi na odległość, co wobec dynamicznego rozwoju tej branży, nie tylko zresztą wywołanego pandemią, należy przyjąć jako zmianę korzystną. Proponowane zmiany mają za zadanie uszczelnienie obrotu wyrobami akcyzowymi także pod kątem wymogów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W nowych regulacjach znaleźć można także przepisy normalizujące obszar zwrotu akcyzy. To zmiana, o której branża mówiła od dłuższego czasu, jednak nie wprowadzano jej w życie. W procedowanym projekcie wreszcie znalazła się długo oczekiwana przez branżę obniżka stawki akcyzy dla małych wytwórców napojów alkoholowych. Wskazane przepisy wprowadzają możliwość stosowania obniżenia stawki akcyzy o 50% w stosunku do stawek podstawowych, m.in. na wina wyprodukowane przez małego producenta wina, napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych oraz wyroby pośrednie wyprodukowane właśnie też przez małe podmioty. W procedowanym projekcie znalazły się także nowe kompetencje Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W noweli znalazły się przepisy wydłużające byt papierowych ewidencji akcyzowych, choć z drugiej strony trzeba przyznać, że zachowano je chyba tylko na wszelki wypadek, bo ewidencje są również w noweli z podwyżkami stawek. Przedmiotowa zmiana reguluje przypadki zwrotu dotychczasowych znaków akcyzy oraz ważności tych znaków naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych po wprowadzeniu nowego wzoru znaków akcyzy, w sytuacji gdy minister wprowadzi okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych znaków akcyzy. Zmiana ta, na plus, ułatwi podmiotom prowadzenie działalności gospodarczej. Bardzo dziękuję panu posłowi. Teraz zapraszam na mównicę pana posła Czesława Siekierskiego, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska.

Szanowni Państwo! Przedstawiona regulacja ma na celu harmonizację procedur akcyzowych i celnych w związku z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego i wprowadzenie nowej kategorii podmiotów.

Ponadto zostały także zapisane rozwiązania, które mają uelastycznić możliwość sprzedaży wyrobów akcyzowych na odległość.

To są rozwiązania, które w jakiś sposób w ciągu kolejnych lat uporządkują to czy dadzą pewne preferencje dla rozwoju małych firm w zakresie produktów regionalnych, które są w Polsce coraz bardziej popularne i są istotną formą dodatkowych dochodów dla małych producentów, w tym dla małych gospodarstw rolnych, albowiem rośnie produkcja winorośli, głównie w małych zakładach, w małych gospodarstwach. Jak państwo wiecie, Polska w przeszłości była liczącym się producentem spirytusu. Oczywiście tu się wszystko pozmieniało, bo wiele gorzelni zostało zlikwidowanych, ale dalej pozostajemy jednym z największych producentów w Unii i czwartym na świecie, jeżeli chodzi o produkcję wódek. To jest forma przetworzonego produktu, który daje wyższe korzyści na rynku.

Pojawiły się piwa smakowe.

Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Głos teraz zabierze pan poseł Mirosław Suchoń, który przedstawi stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050.

Bardzo uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Szanowni Państwo! Przedstawiony przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zmierza do wdrożenia do polskiego systemu prawa postanowień prawa europejskiego.

Głównym de facto celem wszystkich tych rozwiązań jest uproszczenie i elektronizacja procesu związanego z poborem akcyzy czy też usprawnienie monitorowania obrotu towarami objętymi akcyzą i ułatwienie sprzedaży wyrobów akcyzowych na odległość. Projekt przewiduje również preferencje podatkowe dla mniejszych wytwórców tych wyrobów. Dzięki przyjęciu projektowanych rozwiązań, w tym wynikających z dyrektywy horyzontalnej, będzie możliwe zagwarantowanie swobodnego przepływu wyrobów akcyzowych, a jednocześnie prawidłowego poboru podatku akcyzowego przez państwa członkowskie. Z tych powodów zmiany przewidują szereg regulacji dotyczących m.in. przedmiotu opodatkowania, podatników, ubytków, zwolnień, obrotu oraz kwestii związanych ze stosowaniem systemu MCS. Co ważne, tutaj uwaga do ministerstwa, termin wdrożenia trzech z tych czterech dyrektyw upływa 31 grudnia tego roku i naprawdę niezrozumiałe jest, panie ministrze, z jakich powodów rząd zwlekał do ostatniej chwili z przedstawieniem tych rozwiązań. To oceniamy bardzo negatywnie. W związku z powyższym składam wniosek o przekazanie projektu do komisji w celu szczegółowego omówienia proponowanych rozwiązań. Jednak, szanowni państwo, przy okazji procedowania nad tym projektem, który ma usprawnić kwestię akcyzy, widać, w jaki sposób rząd i nieodpowiedzialna działalność prezesa Narodowego Banku Polskiego, który świadomie działa na rzecz deprecjacji złotego, szkodzą obywatelom. W projekcie ustawy rząd przewidział podwyżkę akcyzy na olej opałowy, węgiel, koks i gaz ziemny, czyli de facto na ogrzewanie. To w oczywisty sposób uderzy w obywateli. Co prawda w uzasadnieniu rząd powołuje się na kwestie związane z minimalnym poziomem akcyzy związanym z kursem euro i na to, że należy go zaktualizować. Jednak deprecjację złotego bardzo silnie wspierali i rząd, i prezes Narodowego Banku Polskiego pan Glapiński. Panie Ministrze! W dobie szalejącej drożyzny, bardzo wysokiej inflacji (Dzwonek) dochodzącej już do 8% podwyższenie podatków z tytułu opału tuż przed zimą uderzy w ludzi. Jest to tym bardziej zaskakujące, że rząd ostatnio dużo mówi o tym, że ceny ogrzewania należy obniżyć, dlatego dzisiaj, panie ministrze, panie marszałku, Wysoka Izbo, żądamy procedowania nad projektami Polski 2050, które będą chronić Polaków przed drożyzną, oraz przedstawienia przez rząd ustaw, o których pan premier tyle opowiadał, i nadal opowiada, a konkretnych działań nadal nie ma. Czekamy, panie ministrze, i bardzo negatywnie oceniamy podnoszenie podatków na opał przed okresem zimowym. Na tym zakończyliśmy wystąpienia klubowe.

Jeszcze pani poseł. Dobrze. Ustalam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Rozumiem. W takim razie teraz pan poseł Jan Szopiński. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ustawy powstał, wierząc w słowa autorów, w celu uproszczenia procedur.

Czy urząd skarbowy naprawdę nie ma innych zajęć niż pilnowanie, kto i kiedy dokonał takiego zakupu, a ustawodawca jest przekonany, że podatnik nie ma pilniejszych obowiązków niż pilnowanie, czy ostatni zakup odbył się 360 czy może 365 dni temu? Czemu ma służyć ta biurokracja? Uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania pana posła Rafała Adamczyka.

Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To doprawdy zadziwiające, że w dobie szalejącej drożyzny, w dobie tak wysokiej inflacji, w dobie bardzo wysokich kursów walut i bardzo niskich wartości naszej narodowej waluty, za którą odpowiadają rząd - pana rząd, panie ministrze - i prezes Glapiński, państwo tłumaczą podwyżki akcyzy na opał tym, że kurs euro jest wysoki. To państwo za to odpowiadają, rząd za to odpowiada, odpowiada za to prezes Glapiński. Wypadałoby, panie ministrze, tutaj przyjść i przeprosić obywateli za to, że cały czas działacie na ich niekorzyść. Działacie specjalnie, żeby złoty tracił, i efektem tego są podwyżki, m.in. cen opału. I drugie pytanie, panie ministrze, o to zaniechanie, które wszyscy widzimy, czyli tak późne przedstawienie (Dzwonek) projektów ustaw. Dlaczego nie zrobiliście tego wcześniej? Czy na sali jest pan poseł Michał Szczerba? Nie widzę. Wobec tego pytanie zada pan poseł Janusz Cichoń. Wysoka Izbo! Chcę zwrócić uwagę na szczegółowe rozwiązanie związane z VAT, a tak naprawdę z wyrokiem ETS i próbą naprawienia reguł gry, jeśli chodzi o podatek od towarów i usług. W takiej formule i w takiej treści ten przepis będzie bardzo łatwo obejść. Nieuczciwe podmioty będą przewozić paliwo, na które nie będą wystawiać faktury, celując szczególnie w transporty lewego paliwa na początku miesiąca, a wówczas nie będzie podstaw do tego, aby żądać zapłaty podatku aż do 16. dnia kolejnego miesiąca. W międzyczasie paliwo się rozpłynie, zostanie sprzedane, np. w składzie. Dzisiejszy sens tego przepisu polega na tym, że fizyczna kontrola KAS-u, ulokowana na granicy, może w każdej chwili przejąć transport, jeśli nie zapłacono podatku z chwilą jego wwozu na terytorium Polski. Jeśli (Dzwonek) zmodyfikujecie ten przepis w taki sposób, jak proponujecie, to przewoźnik będzie utrzymywał, że nie ma faktury, bo nie została wystawiona, a może ją wystawić do 15. następnego miesiąca. Formalnie wszystko w porządku, ale tak naprawdę paliwo może się rozpłynąć.

Czasu macie niewiele, dlatego może trochę przydługo, ale to rzecz moim zdaniem istotna, biorąc pod uwagę szczelność systemu podatkowego. Proszę o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Marchewkę. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mamy do czynienia z najwyższą inflacją od ponad 20 lat. W tym miesiącu wzrost cen wyniósł prawie 8%. To jest sytuacja, która bardzo mocno uderza w portfele konsumentów, szczególnie przed świętami.

Wprowadziliście szereg nowych podatków i opłat, które dodatkowo przyczyniły się do wzrostu cen i usług, za które płacą każdego dnia obywatele. Mimo że zapowiadacie kolejne obniżki akcyzy, to - jak wynika wprost z tego dokumentu - w innych miejscach ta akcyzy wzrasta, co oczywiście uderzy po kieszeniach Polaków. Bardzo dziękuję. Pytanie zada teraz pani poseł Małgorzata Pępek. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Nowela zakłada m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. O wprowadzenie takiego rozwiązania apelowali winiarze i cydrownicy. Procedowana ustawa dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Jako kraj, który jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej i trzecim największym na świecie, powinniśmy wykorzystywać potencjał naszych producentów i wprowadzać rozwiązania wspierające mały biznes i produkty wytworzone w Polsce. Rządzicie już 6 lat, dlaczego nie wprowadziliście takich przepisów odpowiednio wcześniej?

Niedawno na alkohol, papierosy, olej opałowy, węgiel, gaz. Nie obchodzą was Polacy. Wolicie tylko ciągle podnosić akcyzę i liczycie na jak największe kolejne wpływy do budżetu. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Tomaszewskiego. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowni Przedstawiciele Rządu! Ustawa ta, jak wynika z uzasadnienia, jest implementacją prawa unijnego, ale także ma uprościć pewne procedury.

Prosiłbym uprzejmie o odpowiedź na piśmie, które z przepisów są pochodną tych konsultacji, a które zostały częściowo uwzględnione. Po drugie, ustawa wprowadza certyfikat małego przedsiębiorcy wina i napojów fermentacyjnych. Wczoraj omawialiśmy ustawę o wyrobach winiarskich, tam jest taka definicja: „drobny producent wina”

Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Nieodpowiedzialna polityka rządu i upolityczniony Narodowy Bank Polski doprowadziły do sytuacji, że inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat. To będą najdroższe święta od bardzo wielu lat. W związku z tym mam pytanie - i bardzo proszę o odpowiedź na piśmie, o przedstawienie na piśmie opracowań, bo rozumiem, że Ministerstwo Finansów dysponuje takim dogłębnym opracowaniem - jak te zmiany dotyczące akcyzy, ale także wszystkie te, które w ciągu ostatnich 2 miesięcy zostały wprowadzone, wpłyną na poziom inflacji w Polsce, która - powtarzam - jest najwyższa od ponad 20 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zada teraz pan poseł Wojciech Saługa. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W 2014 r. prezydent Putin objął embargiem import polskich jabłek i wtedy rozpoczął się bum na cydr. Mówiono, że to będzie takie nasze narodowe dobro, które będziemy wspierać, tym samym będziemy przeciwstawiać się wrogim działaniom prezydenta Putina.

Z roku na rok notujemy spadek sprzedaży. Robicie nareszcie, tak bym powiedział, jakiś ukłon w kierunku producentów, ale drobnych, małych.

Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Czesława Siekierskiego.

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pani poseł Paulina Hennig-Kloska. A do pana posła Janusza Korwin-Mikkego: jest możliwość zadania pytania poprzez. Panie Ministrze!

Dziś procedujemy nad ustawą, w której m.in. akcyza na gaz ma iść w górę. A więc jak to jest w końcu? Bo wygląda na to, że na kwartał akcyzę na środki opałowe chcecie obniżyć po to, żeby trwale ją podwyższyć. Uzasadniacie to osłabieniem się złotego. Ale efekt słabnięcia naszej waluty to polityka stosowana przez bank centralny i prezesa Glapińskiego. Pytanie, dlaczego za permanentne osłabianie złotego, do czego prezes Glapiński przyznawał się wielokrotnie w wywiadach, mają dzisiaj płacić Polacy. Proszę o doprecyzowanie (Dzwonek) tych wątpliwości, które rodzą się wokół waszej polityki energetycznej na najbliższe miesiące. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Korwin-Mikkego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam takie pytanie. Wczoraj uchwalaliśmy, wszystkie kluby poparły obniżkę podatków od małych producentów, dzisiaj mamy głosować nad dalszą obniżką, wymuszoną przez Unię, potem mamy mieć podwyżkę akcyzy, a za kilka dni rząd składa nowy pakiet ustaw, gdzie będzie się obniżało akcyzę. Chciałem spytać: Czy to nie jest po prostu wariactwo? Czy tam naprawdę nie można by nad tym normalnie procedować, czyli - krótko mówiąc - ustalić, że producent to jest producent, płaci podatek, i nie zajmować się, kto jest małym, kto jest średnim, kto jest dużym, tylko po prostu zwyczajnie ustalić raz na zawsze podatki, bo najgorsze są nieustanne zmiany, dla producentów najgorsze są nieustanne zmiany podatków.

Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Teraz pytanie zada pan poseł Artur Dziambor. Wysoka Izbo! Taki trochę wpis Schrödingera. Jest godz. 13.07 i właśnie w tym momencie omawiamy projekt ustawy, która ma obniżyć akcyzę, ułatwić biurokrację.

Tak więc, szanowni państwo. A w przyszłym tygodniu mamy jeszcze posiedzenie Sejmu, na którym będziemy rozmawiali o tym, jak będzie wyglądał pięknie świat po wprowadzeniu tzw. tarczy antyinflacyjnej, co do której wszyscy są zgodni, że ona będzie proinflacyjna, oczywiście poza ekipą z Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiam się, proszę państwa, po co. Może idźmy w tę stronę, przegłosujmy teraz tę ustawę, o której w tym momencie rozmawiamy, co do której wszyscy mamy zgodność, tak jak tutaj powiedział poseł Korwin-Mikke, a następnie odrzućmy podwyżkę akcyzy na papierosy i alkohol - już za 52 minuty będzie to głosowanie (Dzwonek) - a potem odrzućmy też to, co psuje waszą tarczę antyinflacyjną. Bardzo dziękuję. Na tym lista posłów zapisanych do pytań została wyczerpana. Proszę teraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Jana Sarnowskiego o odniesienie się do pytań i wystąpień klubowych. Wysoka Izbo! W pierwszych słowach chciałbym wyjaśnić kwestię procedowania nad tą ustawą. Tutaj trudno mówić o zaskoczeniu rynku przedsiębiorców czy producentów, ponieważ zmiany w dyrektywie, te, które mają być zaimplementowane, znane były już na początku tego roku.

Dlaczego wprowadzamy obniżkę dopiero teraz?

Ile podmiotów, ilu producentów cydru obejmie obniżka?

Padło tutaj bardzo dużo pytań dotyczących podniesienia wysokości akcyzy na gaz ziemny i węgiel. Chciałem gorąco podkreślić, że zmiany w przepisach mają charakter czysto formalny, ponieważ Polska wdrożyła 100% możliwości wyłączeń z tego podatku, na które pozwala dyrektywa. I tak z akcyzy zwolniony jest gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych gospodarstw domowych, organów administracji publicznej, jednostek Sił Zbrojnych, podmiotów systemu oświaty, żłobków, klubów dziecięcych, podmiotów leczniczych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznych i organizacji działalności pożytku publicznego, a także przedsiębiorców, służący do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych i ogrodniczych, w hodowli ryb, używany przez zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby gazowe. Bardzo trudno jest nawet określić liczbę podmiotów, które będą objęte tego rodzaju zmianą w przepisach. Również z tego powodu w ocenie skutków regulacji nie przewidzieliśmy żadnych dodatkowych wpływów budżetowych z tytułu tej konkretnej zmiany w prawie. Tak że bardzo trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek niespójności pomiędzy procedowanymi dzisiaj rozwiązaniami wynikającymi z pewnych wymogów prawa unijnego a generalną strategią rządu dotyczącą obniżek akcyzy. Jeśli chodzi o implementację zmian w podatku od towarów i usług w realizacji wyroku TSUE, to chciałbym gorąco podkreślić, że zmiany, które wdrażamy, są zgodne z wyrokiem i realizują jego treść. Ich wdrożenie przy zachowaniu efektu synergii z innymi wdrożonymi rozwiązaniami uszczelniającymi, takimi jak mechanizm podzielonej płatności czy SENT, czyli nasze narzędzie monitorowania również przy pomocy GPS-ów przewozu paliw, doprowadzi do tego, że zagrożenia rozszczelnieniem nie będzie. Polska w odpowiedzi na wyrok TSUE złożyła wniosek derogacyjny o udzielenie Polsce zgody na kontynuowanie zastosowania dotychczasowej szybkiej płatności VAT-u przy imporcie paliw. Oczekujemy na pozytywną odpowiedź Komisji w tym zakresie, tym bardziej że jest to zmiana korzystna dla przedsiębiorców i bardzo im potrzebna, prowadząca do zwiększenia bezpieczeństwa na rynku, jak również bardzo szeroko chwalona przez przedsiębiorców i w roku 2016, i teraz, podczas procedowania nad tą ustawą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 1795, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Wysoka Izbo!

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 1817. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, druk nr 1811. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu, oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1802 i 1801. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, - o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, - o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, - o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1794, 1807, 1800, 1815, 1805, 1804, 1798 i 1816. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Proszę państwa, bardzo proszę, pani poseł Urszula Nowogórska, Koalicja Polska, z wnioskiem formalnym.

Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Wczoraj dyskutowaliśmy na tej sali plenarnej nad projektem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Wszyscy doskonale wiemy, że strażacy i druhowie ochotnicy jadą tam, skąd wszyscy uciekają. Dzisiaj rano zdarzył się tragiczny wypadek. Strażacy z OSP Czernikowo wyjechali w trybie alarmowym do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Liciszewy koło Torunia. Ich samochód gaśniczy zderzył się z tirem. Proszę Wysoką Izbę o uczczenie minutą ciszy zmarłych tragicznie w wypadku.

Bardzo dziękuję, pani marszałek. Dziękuję państwu. Z wnioskiem formalnym pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica.

Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i wprowadzenie do porządku obrad punktu, w którym pan premier Kaczyński udzieli nam informacji o tym, czy służby specjalne wiedziały o działalności pana Łukasza Mejzy przed powołaniem go na stanowisko i - co ważne - czy wicepremier, przewodniczący komitetu do spraw bezpieczeństwa miał taką wiedzę. Jest to sprawa bez precedensu, żeby na najwyższe stanowiska w państwie wynosić człowieka, który mógł żerować na krzywdzie i cierpieniu ciężko chorych, nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodziców.

Panie Premierze! Ponieważ padł wniosek o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

U kogo nie działa? Proszę sprawdzić u pana posła urządzenie do głosowania. U kogo jeszcze z państwa posłów nie działa? Tam jeden.

Czy już działa, panie pośle? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Proszę. Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości abdykował w walce z pandemią.

Nie znalazł czasu, żeby odpowiedzieć na pytanie o największą liczbę osób na kwarantannie od początku. Czas zmienić ministra zdrowia, który przestał reagować na czynnik społeczny. Pandemia szaleje, minister milczy. Za każdą śmierć odpowiada minister, który nie potrafi reagować. Ponieważ padł wniosek o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Z wnioskiem formalnym pan poseł Wojciech Maksymowicz, Polska 2050. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wyprzedzają nas w tej chwili tylko Rosja i Ukraina. Jest to tragiczny ranking, dlatego też wczoraj posłowie lekarze ze wszystkich klubów opozycyjnych, ale przy zrozumieniu, jak dobrze wiem, również posłów lekarzy z Prawa i Sprawiedliwości, w każdym razie części z nich, zaapelowali do władz o to, żeby zintensyfikować działania, żeby zrobić wszystko to, o czym dobrze wiadomo, ponieważ takie były opinie Naczelnej Rady Lekarskiej, takie były opinie Rady Medycznej przy premierze.

Jedna z tych ustaw będzie rozpatrywana w przyszłym tygodniu, w środę, kolejne są przygotowywane. Ponieważ złożył pan wniosek o zamknięcie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zamknięciem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Wysoka Izbo! Republika Litewska podpisała memorandum, zgodnie z którym język polski miał wrócić na egzaminy maturalne na Litwie w 2022 r. Republika Litewska, jak od 30 lat ma w zwyczaju, chce przeciągnąć rozmowy ze stroną polską do takiego momentu, w którym wprowadzenie tej matury w 2022 r. będzie niemożliwe. O ile po rundzie negocjacji we wrześniu tego roku w Warszawie byliśmy na dobrej drodze do tego, żeby pokazać stronie litewskiej, że nie może kluczyć dalej, że ma zrealizować zapisy memorandum, o tyle po ubiegłotygodniowej wizycie wiceministra Rzymkowskiego ta perspektywa się oddaliła, bo przyjechał nieprzygotowany, bo działał w sposób niekompetentny.

Bardzo rzadko korzystam z takiej możliwości, ale chciałbym wyjaśnić, ponieważ pan poseł Winnicki wprowadza państwa, Wysoką Izbę w błąd.

Został też roboczo uzgodniony harmonogram ze stroną litewską. Natomiast nie będziemy ogłaszać tego roboczo uzgodnionego harmonogramu, zanim nie skonsultujemy go ze środowiskami polskimi na Litwie. I takie konsultacje w tej chwili dobiegają końca, panie pośle. One były prowadzone w ubiegłym tygodniu. Pragnę pana zapewnić, że środowiska polskie w zdecydowanej większości, w zdecydowanej większości, włącznie ze Związkiem Polaków na Litwie, opowiedziały się za przyjęciem takiego harmonogramu, są usatysfakcjonowane. Najbliższe tygodnie przyniosą dobre wiadomości w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1797. Głosujemy.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

436 - za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1799. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1803. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Przyjęcie tego wniosku spowoduje bezprzedmiotowość propozycji komisji. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1803, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wyrobach winiarskich. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1776-A. Proszę panią poseł Teresę Pamułę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Panie Premierze! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wyrobach winiarskich, druk nr 1314.

Komisje: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu tych poprawek na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r. wnoszą:

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1776. Komisje w dodatkowym sprawozdaniu przedstawiają poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1776, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o wyrobach winiarskich. Powracamy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1693, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek przyjął. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1767, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o sądach pokoju. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1760, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczać, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 1761, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1772-A. Proszę pana posła Kazimierza Chomę o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, druk nr 1772-A, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, druk nr 1694. Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w drukach nr 1694 i 1772 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1772. Komisje przedstawiają również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Konsekwencją ich przyjęcia będzie zmiana tytułu ustawy. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 3., 4. i 5., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, w brzmieniu z druku nr 1772, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Otóż w drugim czytaniu dotyczącym zmiany ustawy - Kodeks cywilny i ustawy - Kodeks postępowania cywilnego państwa klub - podpisał to pan marszałek, ale myślę, że nie mając o tym wiedzy - zgłosił poprawki, uwaga, do zmiany W drugim czytaniu. A przypomnę, że zmienialiśmy Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego. Komisja Zdrowia w ogóle nie opiniuje tego projektu ustawy. Nie ma oceny skutków regulacji. Bałagan jest taki w rządzie, że przespaliście kolejny termin. Ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości kilkanaście milionów złotych (Dzwonek) dorzuciło do ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Pan dobrze wie, że nie mogę sobie tak ściągnąć, panie pośle. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1691-A. Proszę pana posła Grzegorza Lorka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo!

Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 r., zgodnie z art. 95 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1344 do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Szanowni Państwo! Nasza rzeczywistość jest jak rozpędzony pociąg lub wyścig z czasem. Chyba wszyscy chcemy zdążyć na czas z odpowiednimi rozwiązaniami. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1691. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie zmiana tytułu ustawy. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1691, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1796-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Mariusza Goska o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sejm na 43. posiedzeniu skierował projekt ustawy do Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Widzę, że jeszcze nie ma. Widzę, proszę państwa, że nie działa, bo mam to samo u siebie.

Proszę państwa, jeszcze raz: Kto jest za przyjęciem 1. poprawki? Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? U kogo nie działa?

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy.

Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1796, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Powracamy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1809-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Pawła Hreniaka o przedstawienia dodatkowego sprawozdania komisji. Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, druk nr 1765. Jest to historyczny moment. Na tę ustawę środowisko druhów strażaków czekało 30 lat.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1809. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

W 7. wniosku mniejszości do art. 7 projektu ustawy wnioskodawcy proponują dodać ust. 3. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tego wniosku mniejszości spowoduje bezprzedmiotowość poprawek od 2. do 4. oraz 10. wniosku mniejszości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 5. i 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 435 - za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1. Sejm poprawki przyjął. 11. wniosek mniejszości stał się bezprzedmiotowy. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 15. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują nowe brzmienie art. 56 projektu ustawy. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1809, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za - 437, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o ochotniczych strażach pożarnych.

Witamy panów komendantów i komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witamy panów. Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1808-A. Proszę pana posła Jarosława Zielińskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1808, a więc pilny rządowy projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Dziękuję. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw?

odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i z panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość 5. poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 6. i 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1808, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

430 - za, 5 - przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (druki nr 1787 i 1798) Proszę pana posła Dariusza Olszewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, druk nr 1787. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 26 listopada br. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do połączonych komisji w celu rozpatrzenia. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. wnoszą, aby Wysoki Sejm raczył poprawki Senatu zawarte w 11 punktach przyjąć, a zawarte w 15 punktach odrzucić.

Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Z poprawką tą łączy się poprawka 9. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 2. i 9., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za - 1, 431 jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Senat proponuje zmiany redakcyjno-legislacyjne. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 431 posłów. Nie był nikt za, 431 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 16. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 - za, przeciw - 435, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 20. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za nie był nikt, 437 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

3 - za, przeciw - 431, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1783 i 1801) Proszę pana posła Piotra Króla o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1783.

Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie. Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Głosujemy.

Kto jest przeciw?

Nikt nie był za, 433 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Nikt nie był za, 433 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt nie był za, 427 - przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 23. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 26. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 34. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 35. poprawce Senat proponuje zmiany do art. 68 ust. 3 oraz art. 76 ust. 2 ustawy nowelizowanej. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 35. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (druki nr 1780 i 1816) Proszę pana posła Jarosława Gonciarza o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, druk nr 1780.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt nie był za, przeciw - 425, nikt się nie wstrzymał.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 3. i 5., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1781 i 1794) Proszę pana posła Jerzego Polaczka o przedstawienie sprawozdania komisji.

W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury rozpatrzyła 15 poprawek, które Senat wniósł do projektowanych przez Sejm zmian. 10 z tych poprawek komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjąć, a pięć poprawek odrzucić. Dziękuję. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

1 - za, przeciw - 430, nikt się nie wstrzymał. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Senat zgłosił do art. 2 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Senat proponuje zmiany redakcyjno-legislacyjne. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 - za, 417 - przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest odrzuceniem 14. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (druki nr 1782 i 1800) Proszę pana posła Jana Warzechę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Senat wniósł trzy poprawki redakcyjno-legislacyjne do art. 62f. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w dniu 30 listopada br. rozpatrzyła te poprawki i wnosi o ich przyjęcie w głosowaniu łącznym. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1784 i 1815) Proszę pana posła Grzegorza Lorka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, druki nr 1784 i 1815.

do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm raczył poprawkę Senatu przyjąć. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. W jedynej poprawce Senat proponuje zmianę w art. 2. Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (druki nr 1786 i 1805) Proszę pana posła Leszka Dobrzyńskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Komisja rozpatrzyła wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 30 listopada tego roku i wnosi o odrzucenie wszystkich poprawek wniesionych przez Senat. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki 4., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki 6., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki 8., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Panowie z Konfederacji, ci, którzy powinni mieć maseczki. Siedzę kilka godzin, czytam w tej maseczce, nie zdejmuję jej z szacunku dla osób, które siedzą obok mnie. Panie pośle, bardzo proszę o założenie maseczki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 9., 11. i 12., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1785 i 1804. Proszę panią poseł Danutę Nowicką o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, druk nr 1804, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1785. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 26 listopada 2021 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? U kogo nie działa? Proszę państwa, u kogo?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Senat zgłosił do art. 2 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1791 i 1807) Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo!

Komisja po dyskusji odrzuciła przedmiotową uchwałę Senatu i rekomenduje Wysokiej Izbie jej odrzucenie. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. Komisja wnosi o odrzucenie tej uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1792 i 1802) Proszę panią poseł Iwonę Arent o przedstawienie sprawozdania komisji. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1792 i 1802.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Przystępujemy do głosowania.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zieloni złożył wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, - Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolerów NIK w zakresie funkcjonowania i gospodarowania środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej; - Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem) złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie interwencji Policji w Lubinie w dniu 6 sierpnia br. i okoliczności śmierci mężczyzny zatrzymanego w czasie interwencji. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o te punkty. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Wiem, widzę, proszę państwa, widzę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1817) Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 1817, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Bardzo bym prosiła o chwileczkę uwagi. Chciałam tylko państwa poinformować, że nasi koledzy parlamentarzyści z parlamentu słowackiego podjęli uchwałę wspierającą nas, Polskę, w walce z reżimem Łukaszenki na Białorusi. Prosili o przekazanie pozdrowień, życzeń i wyrazów wsparcia. Bardzo dziękujemy.

Proszę państwa, podobne uchwały podjęliśmy wspólnie z parlamentami litewskim, łotewskim i estońskim, więc dziękujemy wszystkim naszym kolegom parlamentarzystom za tę solidarność. Dziękuję bardzo i ogłaszam 10 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 34. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 1811) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Piotra Patkowskiego o przedstawienie projektu ustawy. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej. Ta zmiana stanowi część ogłoszonego w zeszłym tygodniu pakietu zwanego tarczą antyinflacyjną albo tarczą osłonową dla gospodarstw domowych dotkniętych wzrostem inflacji. Mianowicie ten projekt nie zawiera wszystkich postulatów zawartych w tarczy inflacyjnej, ale wynika to z tej przyczyny, że części zmian, szczególnie dotyczących obniżki VAT-u na gaz, energię elektryczną i ciepło z sieci, ciepło z ciepłowni, można dokonać w rozporządzeniu. W związku z tym te zmiany zostaną dokonane w drodze rozporządzenia, nad którym Ministerstwo Finansów już pracuje.

Kilka wyjaśnień. Jeśli chodzi o akcyzę na benzynę, na paliwa - bo to obejmuje nie tylko benzynę, ale także diesel czy gaz wykorzystywany do tankowania samochodów - proponujemy obniżkę w terminie od 20 grudnia tego roku do końca maja roku przyszłego. Obniżamy tę stawkę do absolutnych minimów, na jakie pozwala Komisja Europejska. Chciałbym także zwrócić uwagę, że nie dotyczy to tylko samej akcyzy, ale także opłaty emisyjnej. W związku z tym ta przedmiotowa zmiana obniża zarówno akcyzę, jak i opłatę emisyjną do minimum, na które pozwala Komisja Europejska. Większej obniżki po prostu nie możemy zrobić z tytułu przepisów unijnych. Oprócz tego przedmiotowa ustawa zawiera zmiany i obniżkę akcyzy na energię elektryczną. Po pierwsze, obniżamy akcyzę na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Czyli od momentu wejścia w życie tej ustawy, od 1 stycznia do końca maja przyszłego roku energia elektryczna dla gospodarstw domowych nie będzie opodatkowana akcyzą.

Bo jest to absolutne minimum, na które pozwala Komisja Europejska. Natomiast obniżamy akcyzę do absolutnego minimum, na które pozwala Komisja Europejska, dla wszystkich przedsiębiorców. Ponadto, Wysoka Izbo, zawieszamy podatek od sprzedaży detalicznej na paliwa silnikowe, również od 1 stycznia do końca maja przyszłego roku, co też przełoży się na spadek cen benzyny czy szeroko pojętych paliw. Po prostu ten podatek od sprzedaży detalicznej na stacjach benzynowych dla paliw zostaje całkowicie na ten okres zniesiony. Nie walczymy, pani poseł, z problemami, które sami stworzyliśmy, bo z tego, co pamiętam, podatek akcyzowy obowiązywał także za rządów Platformy Obywatelskiej. Nie pamiętam, żeby on wtedy był obniżony.

Bo wszystkim tym, którzy mówią, że jest to rozwiązanie doraźne, rozwiązanie, które nie pomaga w walce z inflacją, przypomnę tylko słowa samej opozycji, która ostatnio nawoływała przecież do obniżenia podatków, a także Komisji Europejskiej, która jeszcze w październiku zachęcała państwa członkowskie do tego, żeby obniżać akcyzę na energię elektryczną, obniżać inne obciążenia podatkowe. Tak że to państwa ulubiona Komisja Europejska, najlepszy wyznacznik tego, co rząd polski waszym zdaniem powinien robić, to zalecała. My to wdrażamy.

Inflacja jest sytuacją bardzo poważną społecznie, bardzo też przez społeczeństwo odczuwaną. W związku z tym będziemy w I kwartale przyszłego roku patrzeć, jak ta inflacja będzie się rozwijała. I gdyby się okazało pod koniec marca przyszłego roku, czy na początku II kwartału przyszłego roku, że polskie rodziny, polskie gospodarstwa domowe dalej wymagają wsparcia i pomocy ze strony rządu właśnie poprzez obniżki podatków, to jako rząd oczywiście będziemy na to gotowi i będziemy stanowczo reagować. I kwartał przyszłego roku, ale to jest pakiet, który nie jest pakietem zamkniętym. Jest pakietem, który ma pozwolić zastanowić się, gdyby była taka potrzeba, gdyby były takie oczekiwania ze strony społeczeństwa, jak dalej pomagać polskim gospodarstwom domowym przy obecnej wysokości inflacji. W związku z tym proszę Wysoką Izbę o poparcie tego projektu ustawy. Proszę też o czytanie tego projektu ustawy właśnie z innymi rozwiązaniami, o których mówiłem. Chodzi o obniżenie VAT-u na 3 miesiące od 1 stycznia do końca marca do 5% na energię elektryczną, obniżenie VAT-u na gaz do 8% od 1 stycznia do końca marca przyszłego roku i obniżenie, bardzo dziękuję za ten pomysł panu ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu, to bardzo, bardzo dobra idea. VAT-u na ciepło do 8% na te 3 miesiące, kiedy Polacy najbardziej grzeją. Taka konstruktywna współpraca rządu z parlamentarzystami pozwala tworzyć dobre i owocne programy dla polskich rodzin i polskich gospodarstw domowych. Kolejnym projektem ustawy, który pewnie będzie prezentował minister klimatu, będzie pakiet dodatków osłonowych dla najbardziej tego potrzebujących gospodarstw domowych. Wiemy, że inflacja jest poważnym problemem społecznym. Wiemy, że gospodarstwa domowe, polskie rodziny oczekują reakcji rządu i reakcji Sejmu na ten problem. I dzisiaj mam zaszczyt przedstawić pierwszy projekt ustawy, pierwszy akt normatywny, który ten problem rozwiązuje. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół.

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec ustawy, którą przed chwilą przedstawił pan minister. Przede wszystkim dziękuję bardzo w imieniu klubu za tę ustawę i za zapowiedź innych zmian, które spowodują zahamowanie inflacji. Myślę, że społeczeństwo czekało na ten projekt. Tak, rzeczywiście na tej sali sejmowej w zeszłym tygodniu, tj. na poprzednim posiedzeniu Sejmu, dyskutowaliśmy na wniosek opozycji o inflacji.

Zarekomenduję projekt do dalszego procedowania. Zachęcam do zapoznania się z tym projektem ustawy. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość rekomenduję przyjęcie tego projektu ustawy. Bardzo proszę, pani poseł Marta Golbik, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Rozumiemy, że dopiero teraz dostrzegliście problem, skoro w tej chwili trafiła ustawa, specjalnie zwołano posiedzenie Sejmu na przyszły tydzień, ponieważ problem inflacji pojawił się nagle. Uważamy, że z tym projektem ustawy powinniście się wstydzić przychodzić do polskiego parlamentu, ponieważ ta ustawa to jest działanie propagandowe i pozorne. To jest leczenie objawów, a nie przyczyn. Panie Premierze! Taka uwaga, że najlepszą tarczą antyinflacyjną byłby niezależny bank centralny, który odpowiednio wcześnie reagowałby na problemy. Prawdziwym impulsem antyinflacyjnym byłaby obniżka VAT-u na energię, paliwa i gaz do zera. Czesi potrafią obniżyć energię elektryczną do zera, my nie potrafimy. Pytanie, czy rząd z premierem Morawieckim na czele celowo nie reagował wcześniej, korzystając z wyższych wpływów do budżetu. Inne kraje potrafiły reagować wcześniej. Wy czekaliście. Dzisiaj, kiedy wzięliście już tyle, ile chcieliście wziąć, oddajecie Polakom namiastkę, fundując im najdroższe święta w historii. Obniżka akcyzy ma wymiar symboliczny.

Megawatogodzina będzie 5 zł tańsza, czyli średnio 2-, 3-osobowa rodzina uzyska 10 zł na rok. Brawo. Powinniście państwo i pan, panie premierze, posłuchać przewodniczącego Donalda Tuska, [[Wesołość na sali]] który już w październiku mówił o tym, żeby negocjować zerowy VAT na energię i paliwa, a nie kłamać, tak jak państwo, że negocjowaliście VAT na żywność. Wtedy, gdybyście go posłuchali już w październiku, rodziny odczułyby rzeczywisty spadek cen, litr benzyny mógłby być tańszy o 1,20, a nie o 20 gr, tak jak w waszej propozycji.

Proszę to sobie przeliczyć.

Oprócz zerowego VAT proponowaliśmy państwu pilne działania: przygotowanie, wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, strategii walki z inflacją w celu ochrony przed jej skutkami najbardziej na nie narażonych grup społecznych; wykonanie rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie praworządności w Polsce oraz planowanych reform, co umożliwi uzyskanie pozytywnej opinii dla Krajowego Planu Odbudowy, a w efekcie dopływ środków na konieczne inwestycje i reformy; przywrócenie niezawisłości sędziom i niezależności sądom, co pozwoli zakończyć spór z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską i odsunie groźbę zastosowania wobec Polski mechanizmu warunkowości; zapewnienie stabilnego otoczenia prawnego dla biznesu, co podniesie rekordowo niski poziom inwestycji i wzmocni fundamenty gospodarki, zapewniając podstawę długoterminowego rozwoju. Jako cele długoterminowe proponowaliśmy: przeznaczenie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na konieczną transformację energetyczną i inwestycje w odnawialne źródła energii, co pozwoli obniżyć ceny energii w przyszłości; zapewnienie stabilnego otoczenia prawnego dla biznesu, co podniesie rekordowo niski poziom inwestycji i wzmocni fundamenty gospodarki, zapewniając podstawę długoterminowego rozwoju. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! My zrobimy wszystko w Komisji Finansów Publicznych, pracując nad tą ustawą, aby Polacy realnie odczuli spadek cen. Zrobimy wszystko, żeby te święta nie były najdroższymi świętami w historii. Ale to, co dzisiaj proponujecie, to nie jest żadna ulga dla Polaków, żadna. Skorzystaliście bardzo dużo na wysokiej inflacji i bardzo późno na nią reagujecie.

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otrzymujemy znowu w ekspresowym tempie projekt ustawy, dostaliśmy go godzinę temu. Ustawa oczywiście była zapowiedziana przez pana premiera jako działania antyinflacyjne. Pytanie się rodzi tylko takie: Czemu tak późno to wszystko się dzieje? Przypomnę, że klub Lewicy już w październiku prosił polski rząd i pana premiera o podjęcie działań w tej sprawie. Wtedy mówiliśmy o tym, że trzeba obniżać akcyzę, trzeba obniżać podatek VAT, po to żeby reagować realnie na to, co dzieje się na rynku, i na rosnącą inflację. Wtedy się okazało, że generalnie to nie są mądre propozycje. Przypomnę tylko, co mówił prezes Narodowego Banku Polskiego: mamy pieniędzy w bród i nic nam nie grozi. Przypomnę tylko nowelizację budżetu państwa na ten rok. Pan premier przecież chwalił się, że nagle się znalazło 33 mld dodatkowych środków, jeżeli chodzi o podatek VAT. Oczywiście już wtedy sygnalizowaliśmy, że te środki znajdują się ze względu na galopującą inflację, i mówiliśmy, że to nie jest żaden cud gospodarczy, tylko ceny, które rosną. I żeby była jasność: obojętnie jak będziecie zaklinać rzeczywistość i obojętnie jak propagandowo będziecie mówić, że wszystkiemu winna Unia Europejska, sytuacja gospodarcza na świecie, wojny itd., to jesteście współwinni tej sytuacji gospodarczej, tym rosnącym cenom i tej galopującej inflacji. Współwinni, podkreślam, bo rzeczywiście to, co się dzieje na zewnątrz, ma wpływ na to i co do tego nie ma wątpliwości, natomiast w dużej mierze przez mądrą politykę gospodarczą mogliście dzisiaj uniknąć tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, bo mamy wrażenie, że ta inflacja po prostu wymknęła wam się absolutnie spod kontroli. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o transformację energetyczną, można było od 2015 r. tę transformację realnie prowadzić. Co wy robiliście? Wspomniany pan minister Tchórzewski, którego bardzo szanuję, wtedy, w 2016 r., mówił: my ten węgiel będziemy przez 50 lat jeszcze wydobywać, ten węgiel to jest w ogóle podstawa funkcjonowania i bądźcie spokojni, wszystkie kopalnie będą funkcjonować. Dzisiaj oczywiście musimy w trybie pilnym tę transformację przeprowadzać. I żeby była jasność: płaci za to odbiorca, my wszyscy płacimy za te błędne decyzje. Rzecz druga. Przypomnę słynny wyborczy prezent, który zrobiliście w 2019 r. - wszyscy się dziwili, jak można płacić firmom energetycznym z funduszu rekompensat 10 czy 12 mld zł - bo zbliżały się wybory, trzeba było powiedzieć: tak, nie będziemy w tej chwili podwyższać cen energii. Wszyscy doskonale wiedzieli, że jeżeli nie podwyższy się ich o 5% w 2019 r., to w 2020 r. trzeba będzie podnosić o 15% i to będzie jeszcze bardziej bolało, ale oczywiście wybory były dużo ważniejsze. Co się dzieje ze środkami z tych słynnych świadectw emisji CO2? Tak, rzeczywiście, one wzrosły. Ale kto kazał wam jako polskiemu rządowi sprzedawać te świadectwa i zasilać budżet państwa? Paliwa? Orlen sobie kupuje jakieś zupełnie niepotrzebne zabaweczki, typu gazety regionalne, wydając na to pieniądze.

Bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Spodziewaliśmy się wszyscy, że tego typu działania będą podjęte. Trzeba je podjąć. Mamy świadomość, że ten pakiet jest początkiem szeregu działań, które po prostu muszą być przeprowadzone, aby uzdrowić sytuację, którą mamy i która jest bardzo dynamiczna.

Przede wszystkim te pierwsze propozycje to nie jest pakiet antyinflacyjny. Jest to pewnego rodzaju wstępny pakiet osłonowy. Od tego trzeba zacząć.

Właściwie teraz to też jest pewna forma nowelizacji. Pewnie będziemy podobnie podchodzić do tego w roku przyszłym. Tu nie ma dyskusji.

Myślę, że te założenia, które były w budżecie.

Teraz właściwie mamy sytuację, jaką mamy.

To się przekłada na obsługę długu.

Oczywiście to się przełożyło na wzrost zadłużenia. To też można zrozumieć.

Nie wykorzystaliśmy także wszystkich środków, które mogliśmy uzyskać z Unii na wsparcie procesów transformacji w energetyce. A więc myślę, że będziemy rozmawiać, jest o czym rozmawiać, bo tej rozmowy Polacy potrzebują.

Bardzo proszę, pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.

Wysoka Izbo! Troszkę zostaliśmy zaskoczeni tym, że dzisiaj procedujemy nad tą ustawą. Szykowaliśmy się na - i tak już zaskakujący - termin przyszłotygodniowy, ale trzeba powiedzieć, że dobrze, że ta ustawa się pojawia, ponieważ ona zdecydowanie idzie w dobrym kierunku, kierunku co prawda niewystarczającym, ale zawsze pozytywnym. Jedna rzecz, która mnie troszkę bawi w tych zapowiedziach, które są, to np. to, że będzie likwidacja opłaty emisyjnej. Tak że załatwiacie swój własny problem. Będzie też zwolnienie od podatku od sprzedaży detalicznej. Będzie opłata paliwowa jakoś ruszana. To są wasze nowe podatki, które wy wprowadzaliście. W tym momencie, jak to z socjalizmem bywa, bohatersko walczycie z problemami, które sami stworzyliście. Bardzo dobrze, że ustawa została podzielona na tę część, w której rzeczywiście dotykacie jakichś lekkich obniżek podatków, i obok tego będzie pewnie ustawa mówiąca o dodatku osłonowym, który właściwie całkowicie niszczy ten efekt, który chcieliście osiągnąć, czyli efekt antyinflacyjny. Rzeczywistość będzie taka, że po wprowadzeniu dodatku osłonowego, który de facto jest łapówką dla wyborców - doskonale o tym wszyscy tutaj, w tej Izbie wiemy - niestety nie będzie za bardzo czego zbierać. Nasza tarcza antyinflacyjna, tarcza antyinflacyjna Konfederacji, którą prezentowaliśmy wielokrotnie, to m.in. ustawa: tanie paliwo, która leży u pani marszałek Witek i czeka na wprowadzenie. Dziękuję, że ją skopiowaliście od nas, bardzo nam miło. Prąd bez VAT, likwidacja 15 podatków, w tym opłata reprograficzna, np. podatek cukrowy, który wprowadziliście na pierwszym posiedzeniu tej kadencji Sejmu, 0% VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Kłamstwem jest, że Komisja Europejska wam na to nie pozwala. Nie było w ogóle tego typu dyskusji i na pewno nie byłoby z tym problemu. No i przede wszystkim zatrzymanie dodruku pieniądza. Zatrzymanie dodruku pieniądza to jest to, co wy zrobiliście wszystkimi swoimi trzynastkami, czternastkami, piętnastkami, 500+, 1000+, RKO, 300+ i wszystkimi innymi tego typu projektami. Sprawiliście, że polski złoty w tym momencie leży, kwiczy, turla się. Inflacja w tym momencie, spirala inflacyjna, do której doprowadziliście, jest absolutnie nie do zatrzymania, jeżeli będziecie dalej zarządzać tak, jak rządzicie. Polecamy gorąco kopiowanie dobrych rozwiązań od Konfederacji, ponieważ nasze rozwiązania rzeczywiście mogą wam pomóc. Bardzo nam miło z tego powodu, a jeżeli przypadkiem uważacie, że tak się nie da, to przypomnę wam słowa waszego prezesa, który kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś nie jest w stanie (Dzwonek) zarządzać w takich warunkach, to widocznie nie nadaje się do rządzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Jeśli coś tu jest, szanowni państwo, kopiowane, to piątka Hołowni, która została ogłoszona 20 października. Ale dziękujemy, bo to naprawdę były i są dobre rozwiązania, które mogą przynieść ulgę Polkom i Polakom. Ale po kolei. Dlaczego drożyzna jest tak dotkliwa dla naszych portfeli? 8-procentowa inflacja, 8-procentowy wzrost cen oznacza, że osoba, która w tym roku nie dostała podwyżki, utraciła 1 miesiąc swoich dochodów. Do tego doprowadziliście. W ubiegłym roku przybyło w Polsce ponad 400 tys. osób żyjących w skrajnej biedzie. Inflacja, panie premierze, będzie wpychać kolejne osoby do tej grupy, grupy osób żyjących w Polsce w skrajnej biedzie. Umywacie ręce od odpowiedzialności za obecny stan, zrzucając winę na światowe trendy.

Macie w tym swój własny dorobek. To efekt nieodpowiedzialnej komunikacji prezesa Narodowego Banku Polskiego, efekt zadłużania państwa w tempie bezprecedensowym, jeżeli spojrzymy na najnowszą historię Polski. Wiecie, ile urósł dług publiczny przez ostatnie 2 lata? 33%. 1/3 długu publicznego urosła przez ostatnie 2 lata i ten dług rośnie poza kontrolą parlamentu, bo uprawiacie kreatywną księgowość. Ustawa - łaski nie robicie. Niestety, poziom jest niewystarczający. Wiecie, ile wy zarobiliście na wzroście cen i na biedzie Polaków?

Boli, wiem, boli. No, panie premierze, większego skąpca nie spotkałam. Przykładowo podatek od sprzedaży detalicznej zawieszacie, bo mówicie, że wpływa na poziom cen. No tak, wpływa, mówiliśmy to, kiedy go wprowadzaliście do systemu podatkowego. Przecież on wpływa również na poziom cen żywności, które też są horrendalnie wysokie. Idzie Gwiazdka. Dajcie ludziom spokojnie przeżyć święta. Tak jak mówiłam, ustawa jest kierunkowo zbliżona, w zasadzie jest kierunkowo interwencją tożsamą z piątką Hołowni, która proponowała obniżenie VAT, obniżenie rachunków za prąd i gaz, zawieszenie opłaty emisyjnej, ale też odłożenie Polskiego Ładu. który, panie premierze, jest kolejnym bodźcem inflacyjnym. Nie zastanawiacie się niestety ani przez moment, panie premierze.

Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania?

Wysoka Izbo!

Powiedział, że gdyby miał dwa guziki, toby wciskał ten obniżający inflację. To jest, szanowni państwo, podejście poważnego polityka, który mówi o inflacji - powiedzieć, że nie ma guzika, którym mógłby obniżyć inflację. W przypadku rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego są konkrety, a nie jakieś wyimaginowane guziki do naciskania. Przypomnijmy sobie, co mówił pan Donald Tusk, porównajmy dalej. Pan Donald Tusk po wygranych wyborach powiedział, że paliwo teraz może kosztować 7 zł. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zaprezentował zupełnie inne propozycje, które składają się na obniżenie paliwa, np. obniżenie do możliwie najniższego poziomu akcyzy na paliwo, a także zniesienie opłaty od sprzedaży detalicznej.

To są realne pieniądze, które zostaną w kieszeniach Polaków. Tak, szanowni państwo, podejmuje się działania, a nie wymyśla się, że rząd nie da rady niczego zrobić. Konkrety. Obroniliśmy miliony miejsc pracy (Dzwonek) podczas pandemii i teraz będziemy pomagali Polakom walczyć z inflacją. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Do tego mamy przerost zatrudnienia, rosnące płace, karmienie rodzin PiS-u, przyjaciół królika - można by powiedzieć - rotacyjne zarządy, gigantyczne premie.

Są zaniechania, jeśli chodzi o energetykę, jej restrukturyzację i przekształcenia.

Bardzo proszę o spokój na sali. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie widzę pana premiera. W miniony czwartek pan premier Morawiecki przekazał, że - cytuję - „Rząd zastanawiał się nad obniżką VAT do zera na artykuły żywnościowe. Komisja Europejska ma jednak inne zasady. Nie zgadza się na tego typu działania. Gdyby była zgoda po stronie Komisji Europejskiej, jest nasze zobowiązanie, zaproszenie na całe I półrocze przyszłego roku zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe. Ale takiej zgody póki co nie ma”

Polacy w grudniu, historycznie rzecz biorąc, wielokrotnie apelowali o to, aby ceny żywności były niższe. Dzisiaj pan, panie premierze, ma szansę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Proszę państwa, chciałem wrócić do spraw związanych z rolnictwem, bo sytuacja w rolnictwie jest wyjątkowo trudna.

Wiemy, jakie są ceny paliw, energii.

Co się porobiło? Kto by pomyślał, że jak będziemy drukować puste pieniądze, że jak się będziemy deficytować, jak się będziemy zadłużać, to się to skończy inflacją? Kurczę, no niemożliwe.

W objęcia hiperinflacji.

Dlaczego te rzeczy, które są dobre teraz, nie będą dobre za pół roku? Jak będziecie tak robić, to - już teraz wam to powiem - rynki będą antycypować tę przyszłą podwyżkę podatków i się na to przygotują, zamortyzują te efekty, o które wam chodzi. Bo wy próbujecie w ramach tego samego pakietu pompować dalej wydatki socjalne. Tak więc jeśli chcecie to zrobić naprawdę dobrze, to przyjdźcie do mnie, ja wam pomogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję. Panie Premierze!

Oczywiście można z tego powodu klaskać, cieszyć się, skakać tutaj, w Wysokiej Izbie, ale tę refleksję trzeba było mieć wtedy, kiedy uchwalało się wysokie podatki albo grało na obniżenie wartości złotego, bo to właśnie państwo robili, a efekty są takie, jak widzimy. Polska 2050 wielokrotnie zapraszała rząd do pracy nad takimi rozwiązaniami, które pomogą ochronić portfele Polek i Polaków. Już w październiku zaprezentowaliśmy piątkę Hołowni, czyli pięć gotowych, konkretnych rozwiązań przeciw drożyźnie. Niestety, rząd nie chciał tej współpracy i unikał tematu aż do teraz. Pan premier powinien wytłumaczyć obywatelom, dlaczego rząd nie chciał działać przeciw drożyźnie i tak długo zwlekał.

Panie Premierze!

Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Pragnę przekazać wyrazy szacunku i podziękowania panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że w swojej kancelarii, w swoim gabinecie znalazł te guziki, których nie mógł odnaleźć pan Donald Tusk. Panie Premierze!

Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków. Tylko VAT - to słowa najbliższego współpracownika pana Donalda Tuska, pana Grasia. Panie premierze, dobrze - a powtarzam za klasykiem - że nie idzie pan tą drogą. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo! Prezes Glapiński sam powiedział, że dzięki późnemu podniesieniu stopy procentowej budżet centralny zarobił 9 mld zł. W związku z tym teraz, jak rozumiem, oddajecie to, co zabraliście w postaci zbyt późnego podniesienia stopy procentowej. Oddajecie Polakom te 10 mld, więc się tym nie chwalcie. Wzrost inwestycji daje nam długofalowe zahamowanie inflacji. Pytam się: A co po 3 miesiącach? Premier Morawiecki chwali się, jaki to świetny pakiet antyinflacyjny wprowadzacie, mówiąc, że za Tuska nie było takiego pakietu. Szanowny Panie Premierze! Zwracam uwagę, że za rządów premiera Tuska nie było takiej inflacji. Mało tego, jak odchodził, była deflacja. Może pan tego nie wie. W związku z tym przedstawiam wykres. Bardzo proszę, pani poseł Wanda Nowicka, Lewica. Szanowna Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Inflacja szaleje. 2 mln ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. Polityka rządu w tym zakresie opiera się w ogromnej mierze na prognozach Narodowego Banku Polskiego i pana Glapińskiego.

Mam pytanie do pana premiera. Panie premierze, czy nadal zamierza pan opierać swoją politykę finansową na lekkomyślnych, bzdurnych, można powiedzieć, prognozach pana Glapińskiego, który tak naprawdę doprowadził w ogromnej mierze do kryzysu, jaki mamy?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Ile zaoszczędzą Polacy ze względu na obniżkę tych podatków? Bardzo proszę, pan poseł Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie ministrze, udajecie dzisiaj wybawców, którzy ratują ludzi przed drożyzną, ale prawda jest taka, że to wy jesteście za tę drożyznę współodpowiedzialni. Przez ostatnie miesiące i przez lata waszych rządów podjęliście szereg decyzji, które zwiększały i nakładały nowe podatki i opłaty. Wymienię opłatę mocową, wzrost kosztów energii, podatek handlowy, opłatę emisyjną od paliw, podatek cukrowy od napojów, wzrost akcyzy na alkohol, podatek bankowy, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, podatek od deszczu. Ponadto od stycznia wprowadzacie tzw. nowy ład, który uderzy w przedsiębiorców. A prawda jest taka, że jeżeli przedsiębiorcy będą mieli większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, to przeniosą te koszty - na kogo? - na klientów i ceny dóbr i usług znowu mogą pójść w górę.

Prawda jest taka, że trochę wygląda to tak, jakbyście pacjenta, który potrzebuje operacji, leczyli środkami przeciwbólowymi. Tak to wygląda. Ta wysoka inflacja, prawie 8-procentowa, najwyższa od 20 lat, jest wynikiem wieloletnich waszych zaniedbań.

Bardzo proszę, pan poseł Włodzimierz Tomaszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, jakie jest bezrobocie, trzeba również wiedzieć, jaki jest wzrost gospodarczy. Nawet te transfery socjalne jak wpływały? Wpływały na wzrost gospodarczy.

W związku z tym jest to opozycja, która jeszcze na domiar tego wszystkiego stwarza większe niebezpieczeństwo (Dzwonek), bo państwo chcą zagrażać polskim granicom, a nie pomagać, żeby to bezpieczeństwo w Polsce stabilizować. Proszę zobaczyć, kraje. Litwa, te kraje, które są również zagrożone tym bezpieczeństwem, mają także wyższą inflację, to wpływa na to.

No naprawdę, za wszystko w tym kraju odpowiada opozycja. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Nie wiem, dlaczego nie możemy rozmawiać merytorycznie o problemie, tylko cały czas mówimy o Donaldzie Tusku i o jakichś wyimaginowanych problemach. Dlaczego? A ja chcę mówić merytorycznie. Pytam się, dlaczego rząd nie pracuje systemowo, nie wyprzedza pewnych zjawisk, które już są, na rynkach się pojawiają, tylko czeka, kiedy sytuacja jest już dramatyczna. Proszę nie mówić, że sytuacja międzynarodowa wpływa na nasz rynek. Oczywiście w pewnym zakresie tak, ale chcę powiedzieć o cenach benzyny. Kiedy Platforma rządziła razem z PSL-em, cena baryłki kosztowała 128 dolarów. Tydzień temu, szanowni państwo, były to 82 dolary, a dziś jest to 68, ponad 15% mniej. Pytam się, dlaczego te trendy i ta sytuacja już sprawdzona, która istnieje, nie ma żadnego odzwierciedlenia na rynku krajowym. Dlaczego rząd musi o 15 gr, dokonując różnej ekwilibrystyki, obniżać cenę (Dzwonek), a Orlen nie reaguje na ceny światowe, które spadają? Bardzo proszę, pan poseł Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Pan minister przedstawił tu bardzo dobre, konkretne rozwiązania, ale nie zawsze one trafiają do opozycji.

Przypomnę w takim razie kilka faktów, żebyśmy mówili o rzeczach istotnych: Naczelną polityką mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych, dotyczy to wszystkich, tych mniej zamożnych i tych bogaczy. Kto to powiedział? Przepraszam, powiedział to w pierwszym exposé w 2007 r. Ale już w październiku 2010 r. z inicjatywy rządu przyjęta została ustawa okołobudżetowa nowelizująca ustawę o VAT, podnosząca wszystkie stawki podatku VAT o 1 punkt procentowy, wszystkie. W błyskawicznym tempie sejmowa większość przegłosowała podwyżkę składki rentowej z ilu? Rząd Donalda Tuska podniósł także akcyzę na wyroby tytoniowe oraz alkohol. Mówimy o faktach. Oczywiście, przywołajmy może inny instytut. Według licznika długu Forum Obywatelskiego Rozwoju (Dzwonek), nie naszego, pod koniec roku 2013 zadłużenie Polski wyniosło ponad 935 mld zł. Pani Marszałek! Tu panowie cały czas przeszkadzają, trudno po prostu o zmieszczenie się w czasie. Jak pan mówi tyle o Donaldzie Tusku, to brakuje panu czasu na merytoryczne teksty. W związku z tym tylko przypomnę, że właśnie według tego forum wzrost zadłużenia był nieporównywalnie większy i wynosił ponad 50%.

Panie Ministrze! Chciałbym, żebyśmy tutaj przytoczyli konkretne, bo są one bardzo konkretne, propozycje i rozwiązania, które są stosowane w tej ustawie. Bardzo proszę, pan poseł Michał Jaros, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Łatwo się rządzi, kiedy jest koniunktura. Łatwo się rządzi, kiedy jest wysoki wzrost gospodarczy, naprawdę łatwo się rządzi i łatwo się wydaje pieniądze. Na tej sali przed chwilą pan premier rozmawiał z panem posłem Tchórzewskim. Żałuję i ubolewam nad tym, że pan premier zamiast słuchać pana Tchórzewskiego, którego ostatecznie posłuchał, nie słuchał swojego przyjaciela, przyjaciela swojej rodziny, pana prof. Myśleckiego. W jakiej sprawie? Żeby nie budować elektrowni w Ostrołęce. Wiedzieliście od samego początku, bo pan prof. Myślecki od samego początku mówił, że tę elektrownię, którą chcecie budować, za chwilę będziecie musieli rozbierać. W wiele miejsc włożyliście pieniądze, które po prostu przepaliliście. I to jest najgorsze, że zmarnowaliście lata dobrej koniunktury na to, żeby oszczędzać, oszczędzać i się przygotować na trudne lata. Po tłustych latach zawsze są chude lata. Niestety, niestety. Prawda jest taka, że ta ustawa antyinflacyjna to gaszenie wywołanego przez NBP i przez rząd pożaru. Zamiast antyinflacyjnej tarczy (Dzwonek) potrzebny jest nam antyinflacyjny oszczep i miecz. Ale ani rząd, ani NBP nie wiedzą, co robią, a przed Polakami najdroższe święta od wielu lat. Wiele ciężkich miesięcy przed nami. Chcę państwu powiedzieć, że socjaliści zawsze wprowadzali podatki. Wy wprowadziliście wiele podatków. Nie rozumiecie zasad ekonomii. Państwo tego nie rozumiecie, nie znacie się na ekonomii, nie rozumiecie gospodarki.

Na prezenty, żywność, podróże i spotkania planują przeznaczyć średnio o 11% więcej środków niż rok temu. Do tej pory dochody rosły szybciej niż ceny, czyli nie spadały płace realne. Mówię o średnich.

Ostatnio amerykański ekonomista - poczytajcie trochę - oceniając sytuację gospodarczą, wprowadził nowy wskaźnik.

Natomiast w Polsce mamy wysokie tempo wzrostu gospodarczego i niskie bezrobocie. Nie ma czasu na więcej. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana ministra Piotra Patkowskiego o udzielenie odpowiedzi na pytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Były tylko słowa, opowieści.

Kilka konkretów z mojej strony.

Po prostu państwo wyszliście i nie byliście w stanie poprzeć swojego własnego wniosku. Dzisiaj mówicie o tym, że szkoda, że nie przyjęliśmy tego dezyderatu. Jak można poważnie rozmawiać o dezyderacie, którego chyba sami się wstydzicie, bo wychodzicie i nad nim nie głosujecie. Dzisiaj nam o tym przypominacie. Pojawił się zarzut, że nie byliście w stanie przygotować się do tej dyskusji, bo druk pojawił się przed chwilą. To kolejne kłamstwo. Druk na stronach sejmowych, szanowni państwo, pojawił się wczoraj.

Szanowni Państwo!

Nie pamiętam programów, które dotyczyły rozwoju energii wiatrowej czy energii solarnej. Nie było tego, ale dobrze.

W Polsce są jedne z najniższych cen.

Dzisiaj m.in. dzięki jego polityce jesteśmy eksporterem węgla i to od nas uzależnione są inne państwa. Szanowni państwo, bądźmy poważni.

Myślę, że państwo wiecie, że w tym momencie 25% dochodów z ETS trafia na fundusz rekompensat kosztów energii elektrycznej. Od przyszłego roku kolejne 40% będzie trafiało na Fundusz Transformacji Energetyki.

Wdrożyliśmy program „Mój prąd”, dzięki któremu Polacy, którzy chcą, mogą budować panele fotowoltaiczne na dachach swoich domów.

Od wielu, wielu miesięcy prowadzimy z Komisją Europejską rozmowy na temat zerowego VAT-u na przewozy kolejowe, zerowego VAT-u na książki, czasopisma. Odpowiedź Komisji Europejskiej zawsze jest ta sama - negatywna. Były także prowadzone rozmowy na temat zerowego VAT-u na żywność i tu komisja znowu rozłożyła ręce - nie. Szanowni państwo, Czesi również eksperymentowali z zerowym VAT-em i w tym momencie muszą się tłumaczyć przed Komisją Europejską, przed tą samą Komisją Europejską, która zachęca do tego, żeby obniżać podatki.

Jeśli tak, to naprawdę od razu wprowadzimy 0-procentowy VAT na żywność. Wystarczy dobra wola ze strony Komisji Europejskiej. Pojawiła się kwestia dodruku pieniądza. To jest ulubiony argument, który w tej Izbie pada. Rozumiem, że poprzez dodruk pieniądza, bo to jest pojęcie niedookreślone, rozumiecie państwo po prostu wysoki deficyt finansów publicznych. Warto w takim razie powiedzieć, że według badań Komisji Europejskiej, według publicznie dostępnych statystyk za ostatnie cztery kwartały nasz deficyt obejmujący wszystko: tarcze PFR, Fundusz Przeciwdziałania COVID wynosi 2,8%.

Państwo bardzo lubicie, jak nas pouczają państwa zachodnie, na każdy temat, także finansów publicznych. A więc według prognoz znowu Komisji Europejskiej deficyt w tym roku wyniesie 3,3%, a w przyszłym - 1,8%.

A może wzorem powinny być Niemcy, które według prognoz Komisji Europejskiej mają dług publiczny na poziomie 70%?

Warto zajrzeć na te strony i zobaczyć, że mieścimy się w kryteriach Maastricht, a kilkanaście państw Unii Europejskiej w tych kryteriach się nie mieści.

Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, bo mamy zdrowe finanse publiczne i potwierdza to Komisja Europejska. Nie powtarzajcie, szanowni państwo, nieprawdziwej tezy o dodruku pieniędzy, bo to się po prostu nie sprawdza. Trudno mi to w tym momencie powiedzieć. Bardzo dziękuję za to, że - i to jest, myślę, bardzo ważne - i Prawo i Sprawiedliwość, i kluby opozycyjne zapowiedziały albo poparcie tej ustawy, albo dalszą pracę nad nią. To jest dobry objaw.

Natomiast nie możemy poważnie rozmawiać, kiedy pojawiają się ze strony opozycji sprzeczne z przepisami unijnymi propozycje dotyczące obniżenia VAT na artykuły, na które Komisja Europejska nie pozwala obniżyć VAT-u. Ale gdyby Donald Tusk i opozycja, która ma dobre kontakty w Komisji Europejskiej, byli w stanie wpłynąć na zmianę tych przepisów, to bardzo prosimy. Jednej rzeczy, którą zrobiła Platforma Obywatelska w kryzysie w 2011 r. przy wysokiej 5-procentowej inflacji na pewno powtórzyć nie można. Zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wiem, że pana posła denerwuje to, że można się odnieść do tych nieprawd. ale naprawdę, niech pan tableteczkę.

Pan poseł zabiera głos w trybie sprostowania. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan minister oczywiście nie zrozumiał, co przedstawiciele klubów przedstawiali, i chyba to spowodowało, że wprowadził Wysoką Izbę w błąd. Pierwsza rzecz, panie ministrze Patkowski: od dbania o stabilność pieniądza jest Narodowy Bank Polski, a prezes Glapiński, który chyba kibicuje rządowi, robi wszystko, żeby polska waluta nie była stabilna, żeby cały czas osłabiała swoją wartość.

Choćby zawieszenie opłaty emisyjnej. Pan minister po prostu nie słuchał i wprowadził ludzi w błąd. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zawarty w druku nr 1811, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 2 grudnia. Czy jeszcze ktoś z pań i panów posłów chce zgłosić się do oświadczenia? Jako pierwszy głos zabiera pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Znaczenie Piotrkowa w nowo utworzonym w 1815 r. Królestwie Polskim nie było zbyt wielkie. Miasto będące kiedyś jednym z najważniejszych w Rzeczypospolitej, najpierw przez swoje tradycje parlamentarne, później dzięki odbywającym się w nim obradom Trybunału Koronnego stało się niewielką, prowincjonalną, garnizonową mieściną. W mieście i w okolicach stacjonowali strzelcy konni. Wiadomości o wybuchu rewolucji w Warszawie dotarły do Piotrkowa 4 grudnia 1830 r. Na wieść o walkach w stolicy ludność Piotrkowa oraz okoliczna szlachta rozpoczęły spontaniczną zbiórkę pieniędzy i różnych preciozów na cele powstańcze. Wśród darów były najcenniejsze pamiątki rodzinne oraz, jak pisał Krzysztof Urzędowski, historyk: obrączki i sygnety herbowe. Rozpoczęto także formowanie oddziałów regularnych, a także różnych oddziałów ochotniczych. W mieście tworzono jeden ze szwadronów jazdy kaliskiej, a także od połowy grudnia 1830 r. kompanii strzelców pieszych. Już na początku tegoż miesiąca powołano Straż Bezpieczeństwa. Jednostka ta niezależnie od pełnienia zadań porządkowych miała być także rezerwą dla wojsk liniowych. Straż liczyła niespełna 20 tys. członków i miała wyekwipować się w umundurowanie na koszt własny. Była to formacja typowo milicyjna. Jej członkowie pełnili służbę patrolową i wartowniczą w mieście niezależnie od swoich normalnych zawodowych obowiązków. Szczególnie ważne były posterunki przy odwachu, czyli więzieniu. Z nielicznych zachowanych dokumentów wynika, że mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i okolic dość skutecznie wywiązali się ze swoich nakładanych przez nich samych obowiązków. Rząd musiał sprostać, wykonując różne zadania. Natomiast rekrutów trzeba było pozyskać z regionów takich jak Piotrków Trybunalski. Był to naprawdę ogromny wysiłek finansowy dla małych miasteczek, wiosek. Aby móc mu sprostać, powołane zostały tzw. komitety żywności. Na ich czele stanęli najbardziej szacowni obywatele ziemscy. Liczono, iż uda im się sprostać obowiązkowi wyżywienia żołnierzy. Niestety komitety te nie spełniały pokładanych w nich nadziei. Piotrkowscy szewcy obniżyli samorzutnie ceny wykonywanego na potrzeby wojska obuwia. Zebrano w ekspresowym tempie prawie 4 t cennego złomu spiżowego, odesłanego następnie do warszawskiego Arsenału. Realizowano obowiązek dostarczenia pociągów, czyli podwód dla wojska. Wysiłek finansowy i gospodarczy mieszkańców regionu był wręcz tytaniczny. Odwiedzając stary cmentarz w Piotrkowie i przyglądając się omszałym nagrobkom, można dostrzec, jak wielu obywateli miasta i okolic wzięło udział w listopadowym zrywie. Wszyscy zostawili swój ślad, chcąc znów uczynić swoją ojczyznę i tę małą, i tę naszą Polskę, wolną. Bardzo proszę, pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pierwszy tydzień grudnia jest Europejskim Tygodniem Autyzmu. Święto to zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 r. uchwalił „Kartę Praw Osób z Autyzmem” Celem tego szczególnego tygodnia jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tę chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem. Autyzm należy do zaburzeń neurorozwojowych. Osoby w spektrum autyzmu mogą doświadczać trudności w sferze kontaktów społecznych, komunikacji, przejawiać przywiązanie do schematów i rytuałów, wielokrotnie powtarzać określone czynności, inaczej, często intensywniej odbierać bodźce zmysłowe. Symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu są zauważalne już od dzieciństwa, a szybka diagnoza i rozpoczęcie terapii mają istotne znaczenie dla przyszłego funkcjonowania dziecka. Zrozumienie problemów jednostki, specjalistyczna opieka i wspomaganie rozwoju dają szansę na zminimalizowanie problemów dotyczących relacji społecznych i komunikacji oraz umożliwienie samodzielnego życia w dorosłości. Ze względu na to, że osoby w spektrum autyzmu inaczej spostrzegają świat, często spotykają się z brakiem zrozumienia, a nawet z brakiem akceptacji. Reakcje te wynikać mogą z niewiedzy na temat funkcjonowania osób autystycznych, ich potrzeb i problemów. Europejski Tydzień Autyzmu ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i upowszechnianie informacji dotyczących tego zaburzenia. Wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu odbywać się będą niemal w każdym mieście, a ich organizatorami są placówki i organizacje zajmujące się diagnozowaniem i terapią zaburzeń autystycznych. Według danych organizacji Autism-Europe ok. 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest tym rodzajem niepełnosprawności i liczba ta zwiększa się. W Polsce wciąż nie wiemy, ilu ludzi dotknął autyzm. Opieramy się na nieprecyzyjnych danych szacunkowych. Autyzm w szczególny sposób obejmuje całą rodzinę i wraz z rodzinami liczba ta jest znaczna. ONZ obok AIDS, chorób nowotworowych i cukrzycy uznała autyzm za czwarte, największe zagrożenie ludzkości. Celem Europejskiego Tygodnia Autyzmu jest przedstawienie jak najszerszej liczbie osób rzetelnej wiedzy na temat tego zaburzenia, bo tylko przez zwiększenie świadomości społecznej można będzie wdrożyć programy, które pomogą rodzicom zdiagnozować swoje małe jeszcze dzieci, a tym już dorosłym autystom zapewnić bezpieczeństwo, gdy zabraknie ich rodziców. Jako wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu zachęcam wszystkich do wspierania dążeń rodziców dzieci z autyzmem oraz osób zajmujących się cierpiącymi na tę chorobę do zwiększania wiedzy na temat tego zaburzenia, do wspólnych działań, które pozwolą wypracować standardy opieki i wspomagania rozwoju osób dotkniętych autyzmem, aby mogły one samodzielnie funkcjonować, samodzielnie żyć na tyle, na ile jest to możliwe. W dniach od 1 do 7 grudnia włączmy się wszyscy w Europejski Tydzień Autyzmu. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

Odszedł od nas uroczy człowiek.

W roku 1997 Agnieszka Mikołajczyk odbyła lekcje mistrzowskie u wybitnej śpiewaczki włoskiej Renaty Scotto.

Jest godnym następcą mojego pokolenia.

We wrześniu 2002 r. została członkiem zespołu solistów Bayerische Staatsoper w Monachium i od tego czasu jej występów na najsłynniejszych scenach operowych świata, jej wyśpiewanych arii operowych i operetkowych, nazw najznamienitszych orkiestr, które jej towarzyszyły, pod batutami najwybitniejszych dyrygentów, nie sposób wymienić w krótkim wystąpieniu. Ta niebywała kariera została tak nagle, tak niespodziewanie przerwana.

Planowała kolejne występy, kolejne koncerty, pracowała nad doktoratem. Myślała, że będzie wychowywać nowe pokolenie śpiewaków, którzy przysporzą sławy Polsce i dobrze zasłużą się w historii muzyki. Miałem zaszczyt znać Agnieszkę osobiście. Była osobą wyjątkową nie tylko ze względu na kunszt artystyczny, była po prostu ciepłą kobietą, uśmiechniętą, serdeczną. Mimo licznych zajęć i artystycznych wojaży po całym świecie umiała znaleźć czas dla bliskich sobie ludzi i miejsc. W miarę możliwości odwiedzała mamę mieszkającą nadal w Kutnie, rodzinę i przyjaciół, modliła się przy grobach taty, brata i innych osób, które spoczywają na kutnowskim cmentarzu. Agnieszka Mikołajczyk już zakończyła swoją ziemską pielgrzymkę. Tak, pielgrzymkę, gdyż była osobą głębokiej wiary. Najpierw z parafią św. Wawrzyńca, a następnie z parafią św. Jadwigi Królowej Polski w Kutnie. Swoim śpiewem ubogacała oprawę mszy św., szczególnie w okresie najważniejszych uroczystości i świąt kościelnych. Dzieliła się sobą najpiękniej, jak umiała. Nadany pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, jakim uhonorował Agnieszkę Mikołajczyk prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda, niech będzie symbolem wdzięczności każdego z nas za to, kim była i jaka była. W dniu dzisiejszym odbyły się w Kutnie uroczystości pogrzebowe Agnieszki Mikołajczyk. Od teraz, kochana Agnieszko, śpiewaj już tylko Panu Bogu, śpiewaj Mu przez całą wieczność. Wierzymy, że zawsze będziesz blisko Niego. W nas pozostanie pamięć o tobie, o twoim wybitnym kunszcie artystycznym i o twoim człowieczeństwie. Będzie nam ciebie brakować, ale będziemy nadal słuchać twojego cudownego śpiewu zapisanego na płytach i różnych nośnikach pamięci. I będziemy cię pięknie wspominać, bo tylko na najpiękniejsze wspomnienia zasłużyłaś. Spoczywaj w pokoju. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 4 grudnia, czyli już w najbliższą sobotę, odbędzie się Forum Gospodarcze ruchu Polska 2050. Decyzje podejmowane są w oderwaniu od realiów gospodarczych, bardzo często na ostatnią chwilę. Decydują przypadek i wyniki sondaży politycznych, a przyjętych przepisów jest tyle, że nie jest w stanie tego przeczytać nie tylko poseł przed posiedzeniem komisji, ale także specjaliści, którzy mają to prawo później stosować. Tak dalej być nie może. Polityka gospodarcza potrzebuje świeżego, szerokiego spojrzenia. Potrzebuje wsłuchania się w głos przedsiębiorców, pracowników i innych instytucji. Dziś polityka gospodarcza potrzebuje rozsądnych propozycji. Wszystko to znajdziecie w naszym programie gospodarczym, który zaprezentujemy już w najbliższą sobotę. Zapraszam do oglądania relacji na kanałach na naszych mediach społecznościowych, do śledzenia tego, co się dzieje, za pomocą środków masowego przekazu, do komentowania i włączania się w nasze działania. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Zamierza to przedsięwzięcie zlecić dwom spółkom, przy czym prezesem jednej z tych spółek jest aktywny i prominentny działacz i funkcjonariusz Prawa i Sprawiedliwości. Według pełnomocnika rządu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej wybrano dwie polskie firmy, dlatego że są to duże polskie spółki, które dają gwarancję jakości i sprawnej realizacji tego priorytetowego zamówienia. Ponieważ 1,5 mld zł, które rząd zamierza wydać na budowę ogrodzenia, to nie są ani prywatne pieniądze pana pełnomocnika Chodkiewicza, ani prywatne pieniądze polityków PiS-u działających w zespole zatwierdzającym decyzje pana pełnomocnika, ani nawet prywatne pieniądze członków rządu, chciałbym z tego miejsca zapytać pana premiera Morawieckiego, po pierwsze, czy wybrani wykonawcy są jedynymi w Polsce dużymi polskimi spółkami, które dają gwarancję jakości i sprawnej realizacji tego priorytetowego zamówienia. Drugie pytanie: Na jakiej podstawie rząd uznał, że to właśnie te dwie spółki, a nie jakieś inne polskie firmy mają zarobić miliardy na wojnie z Białorusią? Trzecie pytanie: Czy w Polsce nie ma innych dużych spółek, które dają gwarancję jakości i sprawnej realizacji tego zamówienia? Czy może pozostałe polskie spółki są dla rządu za mało polskie lub dla polityków Prawa i Sprawiedliwości są za mało PiS-owskie? Być może wybrani wykonawcy są rzeczywiście najlepszymi spółkami do wykonania tego rządowego zlecenia. Dlatego obie firmy, a w szczególności obaj prezesi powinni być zainteresowani tym, by nie otrzymywać miliardów z państwowych zleceń w atmosferze skandalu przy zielonym stoliku zamiast w uczciwej, publicznej rywalizacji. Dziś zasady, przyczyny i okoliczności wyboru tych firm są niejasne, postrzegane przez wyborców jako towarzysko-polityczne i nie przysłoni tego żadna propaganda, nawet ta mistrzowska w wykonaniu pana premiera. Wzywam rząd do uczciwego i racjonalnego wydawania pieniędzy z budżetu państwa, ponieważ są to pieniądze wszystkich polskich obywateli. Wzywam też rząd do wyłonienia wykonawcy ogrodzenia na granicy z Białorusią w uczciwym i transparentnym postępowaniu. Tak by przy walce z reżimem Łukaszenki nie było przekrętów, wątpliwości i nieprawidłowości takich jak przy walce z pandemią. Sejm powinien oczekiwać informacji od pana premiera w tej sprawie. Bardzo proszę, pani poseł Monika Falej, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wielokrotnie mówiłam z tego miejsca o tym, że Warmia, Mazury i Powiśle są dyskryminowane niemal we wszystkich inwestycjach strategicznych i rozwojowych. Jesteśmy regionem o najsłabszej infrastrukturze drogowej i kolejowej. Mamy jedną z najsłabszych ofert medycznych, opieki medycznej. Najnowsze dane wskazują, że województwo warmińsko-mazurskie odnotowało po raz kolejny najwyższe bezrobocie w Polsce - we wrześniu 2021 r. wynosiło ono 8,7%, wobec średniej 5,6% i najniższej 3,3% w województwie wielkopolskim. Nie jest to tylko tendencja ostatnich miesięcy. Polska dwóch prędkości - uciekające marzenia i rosnące różnice to codzienny obraz północno-wschodniej Polski i powiatów warmińsko-mazurskiego. Przygranicznych miejscowości i gmin odciętych od transportu publicznego. Największym problemem regionu wciąż pozostaje ubóstwo. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. w województwie warmińsko-mazurskim wynosiło 4911,28 zł, podczas gdy w Polsce wynosiło ono 5841,16 zł. W 2011 r. wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w regionie był równy 24,2%. To drugi wynik w kraju. A w 35% gospodarstw domowych dochody były zbyt niskie, by pozwolić sobie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Choć sytuacja na Warmii i Mazurach z biegiem lat jest coraz lepsza, poprawa ta następuje wolniej niż w pozostałych regionach kraju. Pozostajemy w tyle i opadamy z sił, a reszta kraju nam ucieka. Bez strategicznych działań władz centralnych, inwestycji w infrastrukturę i transport drogowy oraz kolejowy nic się w tym regionie nie zmieni. Polska musi rozwijać się w sposób zrównoważony, a każdy obywatel i każda obywatelka powinni mieć równy dostęp do podstawowych usług publicznych. I chciałabym o to zaapelować do rządu. Bardzo proszę, pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zabiegam, jak co roku, o najważniejsze inwestycje dla mieszkańców Pomorza. Jednym z moich priorytetów jest obwodnica Kwidzyna w śladzie drogi krajowej 55. Zabiegam, składałam poprawkę do budżetu na rok następny, o 20 mln.

W związku z tym przebieg obwodnicy został już wybrany i jest on już uwzględniony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Kwidzyna i sąsiednich gmin. Powstała również wielobranżowa koncepcja budowy tej obwodnicy. Wydano wspólnie na ten cel ponad 746 tys. zł. Miasto Kwidzyn jest jednym z największych miast w Polsce bez obwodnicy, które nie znalazły się w programie budowy 100 obwodnic. Zadałam również to pytanie panu ministrowi infrastruktury. Otrzymałam dość szeroką odpowiedź, którą pokrótce zacytuję: Informuję, że inwestycja znajduje się na liście rezerwowej „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”, czyli będzie możliwa do realizacji w ramach ustalonego limitu w późniejszych latach w przypadku uzyskania oszczędności w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji, obwodnic, które zostały ujęte na liście podstawowej „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” Czyli pewnie nigdy. Apeluję więc do pana ministra o ujęcie tej ważnej inwestycji w budżecie i poparcie mojej poprawki do budżetu na rok następny, o pieniądze na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Dziękuję. Pan poseł Tomasz Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Plany budowy obwodnicy sięgają jeszcze czasów 20-lecia międzywojennego, jednak przez kolejne kilkadziesiąt lat inwestycja ta nie była realizowana. Wraz z rozwojem gospodarczym, zwiększeniem wymiany handlowej z Ukrainą Tomaszów stał się miastem tranzytowym, przez które przejeżdżało coraz więcej samochodów ciężarowych. Ruch ten był bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Zgodnie z ostatnim badaniem w ramach generalnego pomiaru ruchu przez Tomaszów Lubelski przejeżdża ok. 18 tys. pojazdów w ciągu doby. Przez szereg lat inwestycja ta pozostawała w sferze marzeń mieszkańców miasta. Przez długi czas byli oni mamieni pustymi obietnicami przez polityków, dla których budowa obwodnicy miała dostarczać tylko głosów w kolejnych wyborach. Swe prawdziwe intencje w sprawie inwestycji na Lubelszczyźnie oraz samej Polski wschodniej zawarli oni w mało parlamentarnych słowach, których na tej mównicy nie sposób przytoczyć. Wraz z objęciem władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy w 2015 r. zmieniła się polityka inwestycyjna szczególnie w odniesieniu do obszarów wschodniej Polski, gdzie występowały ogromne braki w infrastrukturze drogowej. Decyzją rządu premier Beaty Szydło budowa obwodnicy Tomaszowa otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 280 mln zł, zaś 17 listopada 2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. 20 września następnego roku podpisano aneks do umowy, którego przedmiotem było zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni.

Droga ta pozwoli połączyć południową część województwa lubelskiego z Warszawą, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg, znacząco skróci czasy dojazdów, poprawi komfort życia mieszkańców Tomaszowa oraz wpłynie na rozwój gospodarczy tej części Polski. W tym miejscu w imieniu mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i całego powiatu tomaszowskiego składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do budowy obwodnicy. Dziękuję rządowi polskiemu za podjęcie decyzji o realizacji tej inwestycji, inwestorowi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, wykonawcy - firmie Mota-Engil. Jak wynika z informacji przekazanych przez generalną dyrekcję, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę kolejnych trzech odcinków drogi ekspresowej S17 pomiędzy Zamościem a Hrebennem. Są to nie tylko kolejne bardzo dobre informacje dla wszystkich użytkowników dróg, ale także dla tych, dla których zrównoważony rozwój Polski jest gospodarczym i społecznym priorytetem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Sławomir Skwarek, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W tym tygodniu obchodziliśmy uroczyście kolejną, 191. rocznicę wybuchu powstania listopadowego.

Obecnie Dzień Podchorążego jest obchodzony szczególnie uroczyście na uczelniach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. W okolicy mojego miejsca zamieszkania, na Lubelszczyźnie, doszło do dwóch bitew. Wojska polskie pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego rozgromiły rosyjski korpus gen. Geismara. To wydarzenie zostało upamiętnione pomnikami, tablicami pamiątkowymi, m.in. na grobie nieznanego żołnierza, w wierszach Gustawa Ehrenberga i Wincentego Pola. Pamięć o zwycięskiej bitwie trwa do dziś i przejawia się w wielu imprezach organizowanych przez samorządy miasta i gminy Stoczek Łukowski. To m.in. wystawy, sesje popularnonaukowe czy biegi uliczne „Grzmią pod Stoczkiem armaty” Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ rocznica zbiegła się z 475. rocznicą nadania przez króla Zygmunta Starego przywileju lokacyjnego miastu Stoczek Łukowski. Chciałbym również wspomnieć przegraną niestety bitwę stoczoną 19 czerwca 1831 r. pod Łysobykami, dziś Jeziorzanami, znaną również w historiografii jako tzw. wyprawa łysobycka. Wśród przyczyn porażki można wskazać błędy taktyczne, złe dowodzenie, brak przygotowania, kunktatorstwo, co dało argumenty do aresztowania i oskarżenia o zdradę gen. Jankowskiego i gen. Bukowskiego. Dla lokalnej społeczności gminy Jeziorzany bitwa nie jest powodem do wstydu. Wprost przeciwnie, obchodząc uroczyście rocznicę tej bitwy, samorząd gminy upamiętnił przodków - żołnierzy, którzy walczyli i zginęli za wolną Polskę. Niech ta przegrana wyprawa i bitwy będą dla obecnych i przyszłych pokoleń nauczycielkami życia. To, co jednak nie powinno budzić naszych wątpliwości, to fakt, że mieliśmy, mamy i - mam nadzieję - będziemy mieli bohaterów narodowych, także w mundurach. Nie wszyscy zapiszą się na kartach historii imieniem i nazwiskiem, ale wszystkim należy się pamięć. W obliczu wielu zagrożeń musimy dziś pamiętać o naszych rodakach noszących mundur, broniących naszej wolności, o funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej, żołnierzach Wojska Polskiego. Stajemy murem za historią, stajemy murem za polskim mundurem, stajemy murem za ojczyzną naszą. Dziękuję, panie pośle. Wysoka Izbo! W ostatnim czasie doszło do głośnych przykładów bezprawnych zwolnień liderów i liderek związkowych. Zwolnienia Magdaleny Malinowskiej z Amazona i Mariusza Ławnika z mBanku były w oczywisty sposób bezprawne i były kolejnymi przykładami represji antyzwiązkowych. Niestety historie Magdaleny i Mariusza nie są niczym nowym ani odosobnionym. W Polsce od lat można bezprawnie i bezkarnie łamać prawa pracownicze i utrudniać działalność związkową. W 2017 r. pracownicy Kauflandu z Wrocławia dołączyli do Międzyzakładowej Organizacji Wolnego Związku Zawodowego „Jedność pracownicza” Odpowiedź pracodawcy była błyskawiczna. Dyscyplinarnie zwolniono dwóch związkowców, w tym wiceprzewodniczącego związku Przemysława Krajdę, mimo że Krajda podlegał ochronie związkowej. Było to oczywiste i rażące naruszenie prawa. Procesy o przywrócenie do pracy trwały 5 lat. Ostatecznie skończyły się w Sądzie Najwyższym skazaniem jednego z członków zarządu Kauflandu. Sąd nakazał też przywrócenie zwolnionych związkowców do pracy - po 5 latach. Mimo że Kaufland przegrał we wszystkich instancjach, udało mu się osiągnąć cel. Wielu pracowników udało się skutecznie zastraszyć, bo zwyczajnie bali się przystąpić do związku zawodowego w obawie przed zwolnieniem. Związek jednak przetrwał represje, zdołał się odbudować, ale w tym czasie sytuacja pracowników znacząco się pogorszyła. Zmniejszono zatrudnienie, obarczono tą samą ilością pracy mniejszą liczbę osób. W związku z tym związkowcy alarmują, że praca w Kauflandzie obecnie jest ponad siły. Pracowników, których firma chce się pozbyć, straszy się, mówiąc, że albo odejdą dobrowolnie, albo zostaną zwolnieni dyscyplinarnie, pomimo że nie ma ku temu żadnych podstaw. Zdaniem związków zawodowych mobbing w Kauflandzie jest powszechny, a pracodawca w żaden sposób nie próbuje mu przeciwdziałać. W związku z tym związki zawodowe przedstawiły tę sprawę, sprawę mobbingu zarządowi, ale od miesięcy nie mogą doczekać się żadnej odpowiedzi, nawet spotkania. Mimo tej ciężkiej pracy i trudnych warunków pensje w Kauflandzie są niskie i tylko nieznacznie przekraczają pensję minimalną. W związku z tymi wszystkimi okolicznościami w tej chwili w Kauflandzie trwa spór zbiorowy, referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżek i realnej walki z mobbingiem. Ponieważ zarząd Kauflandu konsekwentnie lekceważy stronę społeczną i odmawia spotkania, 6 grudnia, w najbliższy poniedziałek, zdeterminowani związkowcy organizują pod siedzibą firmy we Wrocławiu protest. Osobiście deklaruję obecność na tym proteście. Partia Razem stoi po stronie pracowników. Wspieramy związkowców, jesteśmy solidarni z tymi, którzy organizują się w miejscu pracy, i sprzeciwiamy się wszelkim represjom wobec związków zawodowych. Niestety państwo polskie nie chroni dzisiaj związkowców. Ochrona związkowa zapisana w polskim prawie jest tylko teoretyczna i nie działa w praktyce. Przepisy są martwe, jak pokazują te liczne przykłady, zwalnianie związkowców jest na porządku dziennym. Dlatego tak ważne jest w tym momencie docenienie wszystkich tych, którzy organizują się w miejscu pracy, tak ważna jest nasza solidarność ze związkami zawodowymi. Osobiście pojawię się w poniedziałek na proteście pod siedzibą Kauflandu. Dziękuję bardzo. Nie ma pana posła. Pan poseł Maciej Kopiec, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od ponad tygodnia w przestrzeni medialnej pojawiają się kolejne bulwersujące informacje na temat haniebnych biznesów wiceministra sportu i turystyki w rządzie Mateusza Morawieckiego Łukasza Mejzy. Na podstawie materiału prasowego opublikowanego przez wolne media, portal Wirtualna Polska, w dniu 24 listopada br., zatytułowanego „Jak Łukasz Mejza postanowił zarobić na cierpieniu”, autorstwa Szymona Jadczaka i Mateusza Ratajczaka wraz z posłanką Anitą Kucharską-Dziedzic złożyliśmy pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej w Zielonej Górze. 25 listopada w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy złożyłem na ręce przełożonego pana Mejzy premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o natychmiastową dymisję tego ministra oskarżonego o tak potworne czyny. Fakty, które zostały przedstawione w materiałach prasowych, są następujące. Firma wiceministra Mejzy w swojej ulotce reklamowej cynicznie obiecywała leczenie wielu nieuleczalnych chorób terapią, która zarówno w Polsce, jak i na świecie jest uznawana przez lekarzy za niesprawdzoną, a nawet niebezpieczną. Koszty takiego leczenia zaczynały się od 80 tys. dolarów, co oznacza, że zdesperowani rodzice wpłacali takie kwoty na konto pana Mejzy, motywowani miłością do swoich cierpiących dzieci, z nadzieją na ich wyzdrowienie.

Trefne kuracje bazowały na zapłodnionych komórkach macierzystych, co stanowi kompletne zaprzeczenie polityki rządu, którego członkiem jest minister Mejza. Między 16 stycznia a 17 marca 2020 r. asystenci pana Mejzy zarejestrowali aż 21 stowarzyszeń, które pomagały w pozyskiwaniu klientów, ale również miały prowadzić zbiórki na zagraniczne terapie, przypominam, oszukańczą metodą. Firma naciągająca zrozpaczonych, często nieuleczalnie chorych ludzi oraz ich rodziny na kolosalne wydatki jako podstawową działalność w PKD podaje organizację turystyki. Nie jest tajemnicą, że firma ta nie widnieje w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców prowadzonym przez marszałka województwa lubuskiego. Powyższy rejestr nadzoruje Ministerstwo Sportu i Turystyki, w którym wiceministrem od połowy października jest sam Łukasz Mejza. Spółka pana Mejzy nie złożyła jeszcze obowiązkowego sprawozdania z działalności do sądu. Tyle faktów. Panie Premierze Morawiecki! Panie Wicepremierze Kaczyński! Panie Ministrze Ziobro! Pani Marszałek Witek! Abraham Lincoln powiedział, że najpewniejszym sposobem ujawnienia charakteru ludzi nie są przeciwności losu, lecz danie im władzy. Dlaczego macie tak paskudne charaktery? Z czego wynika wasze milczenie i bezczynność, czego się boicie, bo na pewno nie boicie się stać ramię w ramię z człowiekiem podejrzewanym o antyludzkie przestępstwa motywowane chciwością. Nie ma dobrych parlamentarnych i adekwatnych słów, które zobrazowałyby poprawnie poziom obrzydliwości procederu autorstwa Łukasza Mejzy. Bezwzględne czerpanie zysków z ludzkiego nieszczęścia, dawanie z premedytacją złudnej nadziei śmiertelnie chorym ludziom to dziś moralne podsumowanie sprawowanej przez Zjednoczoną Prawicę rządów, na które się zgadzacie. Wasza władza w imię utrzymania większości bez mrugnięcia okiem toleruje w swoich szeregach każdą niegodziwość. To kolejny polityczny kameleon, którego przynależność do obozu rządzącego czy opozycyjnego zależy wyłącznie od tego, co bardziej się opłaca. Na tym polu nie wyróżnia się na tle wielu oportunistów, natomiast jego podła działalność - na pewno tak. Po opublikowanym przez Roberta Gwiazdowskiego wpisie na jednym z portali społecznościowych nie mogliśmy pozostać obojętni, skoro w przestrzeni publicznej mówi się o jawnym łamaniu zasad demokracji i fałszowaniu list poparcia. Dlatego z Anitą Kucharską-Dziedzic, posłanką ziemi lubuskiej, złożyliśmy drugie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Łukasza Mejzę, z art. 248 Kodeksu karnego, dotyczące podejrzenia fałszowania podpisów pod listami poparcia. To kolejne podejrzenie, za które minister Mejza powinien natychmiast otrzymać dymisję, zniknąć z życia publicznego, a także stać się obiektem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości. Fakty dotyczące działalności Łukasza Mejzy są skrajnie szokujące, i to nie tylko dla opinii publicznej, opozycji, ale również dla samych posłów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Pokazały to dzisiejsze i wczorajsze głosowania. Podziały polityczne w tej sprawie nie powinny i nie mają znaczenia. Chodzi o zwykłą, ludzką przyzwoitość. Mejza jest ode mnie rok młodszy. Reprezentuje wszystko to, z czym ja i większość młodych polityków i polityczek walczymy na co dzień - z polityczną patologią. Skumulował w sobie, mając 30 lat, całą patologię III Rzeczypospolitej Polskiej. Hańbą dla polskiego rządu i parlamentu jest każdy następny dzień, w którym ten człowiek sprawuje swoją funkcję. Parlamentarzyści mówią dziś jasno: nie chcemy pracować, debatować i głosować w obecności człowieka podejrzewanego o tak wstrętne czyny. To całkowity upadek parlamentaryzmu. Polki i Polacy, a przede wszystkim ofiary wypowiadające się w przestrzeni publicznej na was patrzą, a wy uśmiechnięci i pełni frazesów na ustach zacieracie ręce, bo jeszcze tym razem, bo jeszcze na chwilę macie w parlamencie dwa niemoralne głosy przewagi. Do czasu. Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Zwracam się do pana w imieniu wielu rodziców, dzieci i młodzieży cierpiących na depresję. Depresja jest chorobą, która może zagrażać życiu. Jest to długotrwały, szkodliwy i poważny stan nadmiernie obniżonego nastroju oraz objawami psychicznymi, behawioralnymi i fizycznymi. Według Światowej Organizacji Zdrowia ok. 1,5 mln Polaków cierpi na depresję, a za kilka lat będzie to najczęściej występująca choroba na świecie. Wszystko na to wskazuje, że zajmie ona drugie miejsce wśród chorób będących najczęstszymi przyczynami przedwczesnej śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. A co robi rząd w Polsce? Serwuje niestety tylko kampanię nagłaśniającą ten problem, zamiast realnie pomóc w leczeniu. Tanim kosztem i szumem wokół tego tematu nie rozwiąże się tego problemu. A w efekcie nie przybyło psychologów, psychiatrów czy specjalistycznych oddziałów. Nawet na prywatną wizytę dzieci czekają kilka miesięcy. Czy to ma im pomóc? Depresję da się wyleczyć, tylko do tego nasze państwo powinno podejść poważnie. Bo to jest bardzo poważna sprawa dla osób cierpiących na nią i dla najbliższych, którzy cierpią razem z nimi. Dodam, że ten problem dotyczy również wielu dorosłych, którzy znajdują się w tej samej sytuacji. A co państwo zrobiliście z tym tematem? Niestety nic. Potrzebni są specjaliści, a plakaty, szkolenia czy kampanie powinny być kontynuacją i dodatkiem do zabezpieczonych już podstawowych potrzeb, a nie ich zastąpieniem. Dlatego proszę z tego miejsca o pilne i rzetelne zajęcie się tym tematem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Teresa Glenc, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mieszkańcy Górnego Śląska i całej Polski w dniu 20 listopada br. przeżywali wielką radość z beatyfikacji śląskiego kapłana Jana Franciszka Machy, który całym swoim życiem służył Bogu, ludziom i ojczyźnie. Życie i patriotyczna postawa błogosławionego pozostaną na kolejne lata świadectwem prawdy i umiłowania ojczyzny, a także dowodem zbrodniczej hitlerowskiej okupacji w Polsce. Niech bohaterska postawa ks. Machy oraz wielu mniej lub bardziej znanych bohaterów, którzy przelewali krew za naszą umiłowaną ojczyznę, będzie dla nas wzorem i inspiracją w codziennej trosce o Polskę. Dzisiejsze czasy są dla nas wyzwaniem, by okazywać szczególny szacunek kapłanom oraz uczyć nasze dzieci i młodzież poszanowania dla duszpasterzy w obliczu narastającej w ostatnich latach agresji wobec Kościoła katolickiego i duchowieństwa. Jest to powód do głębokiej refleksji, która budzi niepokój o przyszłość naszej ojczyzny, która jest naszym wspólnym dobrem. Błogosławiony ks. Franciszek Macha uczy nas odwagi i ogromnego szacunku do Kościoła. Zadaniem rodziców, wychowawców, ale również nas, polityków, jest nie tylko rzetelne przekazywanie wiedzy, w tym wiedzy historycznej, ale przede wszystkim odpowiedzialność za przyszłość Polski. Widzimy, co się dzieje na zachodzie Europy. Kościoły katolickie są podpalane, zamykane czy przerabiane na dyskoteki bądź bary. Nigdy nie możemy dopuścić, by nurt laicyzacji i ateizacji przeniósł się do Polski. Naszą powinnością jest stać na straży naszych świętych wartości, takich jak wiara, ojczyzna, patriotyzm, w duchu wierności ponad 1500-letniemu dziedzictwu Rzeczypospolitej. Bardzo proszę, pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewica. Wysoka Izbo! 12 grudnia zmienia się rozkład jazdy pociągów, na który to rozkład czekają tysiące pasażerów kolei. Dla części z nich to wyczekiwanie jest jednak przepełnione strachem, ponieważ wprowadzone zmiany stanowią dla nich wyrok. To wyrok odebrania pociągów, którymi na co dzień dojeżdżają do pracy, do szkoły, do lekarza, rodziny czy przyjaciół. Są zmuszeni do zmiany swoich planów, dostosowania godzin pracy do nowego rozkładu, co przecież nie zawsze jest możliwe, przeorganizowania swojego życia, a w skrajnych przypadkach muszą nawet zrezygnować z pracy. Te osobiste tragedie dzieją się w całej Polsce. Nie ominęły także mojego rodzinnego Kutna. Docierają do mnie bowiem głosy mieszkańców, którzy są rozczarowani proponowaną ofertą dotyczącą przewozów kolejowych, którzy są zaniepokojeni tym, co ich czeka. W Warszawie pracuje wiele kutnianek i wielu kutnian, a także sporo osób z okolicznych miejscowości. Pracują na różne zmiany, dlatego potrzebne są połączenia odpowiadające na ich realne potrzeby. Niestety nowy rozkład kolejowy na nie nie odpowiada. Przeciwnie, sprawia, że piętrzą się kolejne kłopoty. Kontaktują się ze mną pracowniczki i pracownicy, którzy już niebawem nie będą mieli jak dojechać na poranną zmianę rozpoczynającą się o godz. 7, ponieważ pierwszy pociąg z Kutna przyjeżdża do Warszawy kilka minut po tej godzinie. Jak będzie wyglądać to w rzeczywistości? Poranny pociąg TLK z Kutna będzie wyjeżdżał o godz. 5.08, aby znaleźć się o godz. 7.03 na Dworcu Centralnym w Warszawie. Podróżujący z Kutna mieli wcześniej możliwość podróży z przesiadką, aby zdążyć. Ale i ta możliwość została im z tym nowym rozkładem odebrana. Problemy dotyczą także godzin wieczornych. Piszą do mnie pasażerowie, którzy kończą zmianę o godz. 22, a ostatni pociąg do domu, do Kutna odjeżdża kilka minut po godz. 20. Później nie ma już żadnego bezpośredniego połączenia. Chciałabym więc zapytać, co mają zrobić ci mieszkańcy. Czy mamy kazać im przesiąść się do samochodów? Przecież nie tak buduje się sprawny system komunikacji zbiorowej. Nie tak zachęca się pasażerów do korzystania z komunikacji zbiorowej. Takie zmiany rozkładu jazdy na kolei, zmiany na gorsze, poważnie podważają zaufanie do transportu publicznego. Dla mnie jako przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym taka sytuacja jest nie do pomyślenia. Jako rodowita kutnianka jestem zbulwersowana lekceważącym traktowaniem pasażerów, którzy dotychczas podróżowali właśnie pociągami relacji Kutno - Warszawa. W ich sprawie interweniuję, w ich sprawię wysyłam interpelacje i zapytania. Apeluję do ministra infrastruktury o racjonalną politykę transportową, która uwzględnia potrzeby podróżujących. Bardzo proszę, pani poseł Wanda Nowicka, Lewica.

Szanowna Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pragnę poinformować, że zwróciłam się z gorącem apelem do pani marszałkini Witek o to, by jak najszybciej podjęła prace nad uchwałą Sejmu jednoznacznie potępiającą skandaliczne, antysemickie wydarzenia w Kaliszu podczas obchodów święta niepodległości, kiedy w czasie wiecu publicznie nawoływano do nienawiści wobec społeczności żydowskiej oraz ją znieważano.

Dokonano też publicznego spalenia statutu kaliskiego z XIII w., który zagwarantował Żydom prawo do mieszkania i przebywania w ówczesnej Polsce. W tej sprawie nie może zabraknąć głosu polskiego Sejmu, głosu jednoznacznie i zdecydowanie potępiającego te zamieszki. W czasie posiedzenia wysłuchaliśmy informacji prokuratora generalnego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji i innych osób.

Niestety, wszystkie źródła wskazują na to, że antysemici czują się, można powiedzieć, zupełnie bezkarni i w związku z tym zamieszki tego typu mają miejsce i są coraz częstsze. Ta sprawa ma ogromny wydźwięk międzynarodowy dla postrzegania Polski jako kraju otwartego, tolerancyjnego i szanującego prawa mniejszości narodowych i etnicznych, mniejszości wyznaniowych. Dlatego my, parlamentarzyści, nie możemy milczeć. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinien dać jasny sygnał opinii międzynarodowej, że w Polsce nie ma przyzwolenia na antysemityzm i ksenofobię. Dlatego też apeluję do pani marszałkini Witek o to, żeby te prace nad uchwałą zostały podjęte jak najszybciej i żeby ta uchwała została przez Wysoką Izbę jak najszybciej przyjęta.

Słuszną sprawą jest poprawa sytuacji ochotniczych straży pożarnych, wzmocnienie ich roli, uhonorowanie wieloletniej i ofiarnej służby. Wprowadzenie świadczenia ratowniczego w wysokości 200 zł dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet brali czynny udział w działaniach, to sprawa niepodlegająca dyskusji.

Z jednej strony w maju pojawił się projekt utworzenia formacji obrony cywilnej z ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP RP. Z drugiej strony we wrześniu zaczęły napływać informacje o toczących się w tajemnicy pracach nad ustawą o OSP, bez konsultacji z tymi, których ma ona dotyczyć. Uregulowania wprowadzane są odgórnie, bez konsultacji ze strażakami ochotnikami. Taki tryb działania jest niebezpieczny, bo ochotników nie da się do niczego zmusić. W efekcie można ich po prostu stracić, tak jak tracimy kadrę Państwowej Straży Pożarnej, w której ludzie po prostu nie chcą już pracować. Nie można organizacji, jaką jest Związek OSP RP i stowarzyszeń, jakimi są OSP, wprost zamieniać w formację obrony cywilnej. Gwarantuje to konstytucja. A jeżeli już mówimy o służbie w obronie cywilnej, to reguluje to ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 142 wskazuje, kto podlega tej służbie, a kto może być z niej zwolniony.

Strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest ok. 30 tys. a członków OSP - ok. 700 tys. Nie wolno ich lekceważyć. Członkowie ochotniczych straży pożarnych jak wszyscy inni ratownicy i społeczni działacze oraz pasjonaci pożarnictwa wchodzili w szeregi stowarzyszenia mającego szczytne cele. Nikt z nich nie podpisywał zgody na to, aby go zmilitaryzowano. Oczywiście są sytuacje nadzwyczajne, w których wszystkie służby działają razem, ale stowarzyszenia, które w statutach mają zapisane ratowanie, pomaganie, edukację, kulturę, nie mogą być odgórnym nakazem wcielane do formacji zmilitaryzowanej. Gdy zagrożone jest życie i zdrowie w czasie pożarów, podczas powodzi czy w wypadkach, strażnicy ochotnicy spieszą z pomocą, ale formacja obronna w sytuacji stanu wojennego czy wyjątkowego może zostać wykorzystana np. do tłumienia strajków czy ulicznych protestów. Nie jestem pewien, czy ok. 700 tys. strażaków ochotników marzyło o tym, wstępując w szeregi OSP. Dziękuję, panie pośle. I bardzo proszę, pani poseł Maria Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Szanowna Wysoka Izbo!

Zanim to się stało, z woli większości posłów i senatorów naszego parlamentu zostało wystosowane pismo, list do kustosza Sanktuarium Narodowego św. Andrzeja Boboli w Warszawie Waldemara Borzyszkowskiego, w którym posłowie i senatorowie napisali: Czcigodny Księże Kustoszu! Jako parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się z prośbą do księdza kustosza o przekazanie relikwii św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, do kaplicy sejmowej znajdującej się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Św. Andrzej Bobola urodził się w 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka w województwie podkarpackim. Był polskim duchownym katolickim, jezuitą, gorliwym misjonarzem zwanym apostołem Polesia, autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.

Od tego czasu był uważany za patrona Polski, ale wybuch II wojny światowej przeszkodził i odsunął na wiele lat oficjalne stanowisko Kościoła w tej sprawie.

Postać św. Andrzeja Boboli, pierwszego patrona Polski, stanowi bezkompromisowy przykład walki o wiarę i wartości z nią związane. W czasie kiedy coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem deprecjonowania znaczenia religii katolickiej w przestrzeni publicznej oraz podważania wielowiekowego fundamentu, na którym budowana jest historia naszej ojczyzny, a którym jest cywilizacja chrześcijańska, my, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, chcemy stawić opór wszystkiemu, co do tego prowadzi. Wpatrując się w życiową postawę tego męczennika, pierwszego patrona Polski, uważamy, że obecność Jego relikwii w kaplicy sejmowej Jego kult będzie wywierał istotny wpływ na parlamentarzystów, którzy w kaplicy modlą się i prowadzą duchowe życie, oraz na pracę całego parlamentu. W związku z powyższym kierujemy naszą prośbę do księdza kustosza o przekazanie do kaplicy sejmowej relikwii głównego patrona Polski, św. Andrzeja Boboli. Szanowni Państwo! To jest wizerunek św. Andrzeja Boboli, którego relikwie od dzisiaj znajdują się w kaplicy sejmowej. Ten największy męczennik Kościoła, co dziwne, musiał się upominać o to, abyśmy go czcili, abyśmy go uznali, a ksiądz kustosz w Słowie Bożym, które było dzisiaj na porannej mszy świętej, przypomniał nam tę niezwykłą historię. Św. Andrzej Bobola jest patronem Polski i jest patronem jedności.

I mam takie marzenie, i życzę państwu i sobie, aby stopniowo wprowadzana była jedność w tej Izbie parlamentarnej, abyśmy się zaczęli nawzajem szanować, dyskutować o Polsce, a nie partyjnie przeciwstawiać się i budować dalsze podziały. Św. Andrzeju Bobolo, strzeż Polski. Dziękuję, pani poseł. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.